Liczymy, że dogodne formy organizowania się i swoboda ich wyboru będą stymulowały większą aktywność społeczną na obszarach wiejskich. Projekt nowelizacji zapewnia kompleksowe regulacje kwestii związanych z tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół. Zmieniamy przepisy określające przekazywanie pomocy finansowej kołom gospodyń wiejskich, przenosimy kompetencje w zakresie udzielania pomocy z ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Następuje też decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich. Wysoki Sejmie! Kołom gospodyń wiejskich pomaga w działalności również Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, którego zadaniem jest m.in. wspieranie tradycyjnej kultury ludowej i odrębności regionalnych. Instytut ten podjął szeroką współpracę z kołami gospodyń wiejskich, doceniając ich bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim. Na przestrzeni lat organizacje te pielęgnowały polską tradycję, promowały sztukę ludową i jednocześnie wywierały silny wpływ na rozwój polskiej wsi. Dziś jest podobnie, chociaż krąg zainteresowań i obszar działania tych organizacji znacznie się poszerza. Obecnie koła gospodyń wiejskich (Dzwonek) angażują się w decyzje na szczeblu lokalnym, wpływają na problemy społeczne, inicjują wydarzenia kulturalne. Szanowni Państwo! Ustawa, jak najbardziej oczekiwana przez środowiska wiejskie, spełniła swoje zadanie, spowodowała, iż środowiska się aktywizują. Wracamy do kultywowania lokalnych tradycji, do organizowania imprez. Ustawa jak najbardziej została dobrze przyjęta przez koła gospodyń wiejskich, przez środowiska wiejskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Bardzo szczegółowo tutaj je przedstawił. Bez wątpienia taka pomoc była niezbędna, bo to spowodowało, że działaczki, a także - co koleżanka przede mną powiedziała - działacze, którzy przystępują teraz do tych zrzeszeń, są bardziej aktywni. Może inaczej, poczuli autonomię, poczuli, że to, co robią, jest wspierane również finansami, o które sami zabiegają, a nie tylko tymi, które otrzymują od włodarzy.

Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Ale teraz powie na pewno. Wysoka Izbo! Tak, postaram się przekazać te informacje.

Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Fryderyk Kapinos i Teresa Pamuła z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie sposobów wspierania rodzinnych gospodarstw rolniczych w kontekście nowej perspektywy finansowej oraz planów promowania w Polsce i za granicą produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych. Pytanie to zostanie skierowane do obecnego tu ministra. Proszę bardzo, pan poseł Fryderyk Kapinos zadaje pytanie. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Podczas wystąpienia na konferencji Europa Karpat pan minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wypowiadał się o rodzinnych gospodarstwach rolniczych. Powołując się na raport ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, mówił, iż dostarczają one światu 80% żywności, wykorzystując 75% gruntów. Według ekspertów FAO tylko rodzinne gospodarstwa rolnicze są w stanie sprostać coraz większym potrzebom żywnościowym przy kurczących się zasobach gruntów, upraw i wody. Odnosząc się do tej wypowiedzi, mam do pana ministra pytanie: Jak w Polsce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza wspierać rodzinne gospodarstwa rolnicze w kontekście nowej perspektywy finansowej? Bardzo proszę, panie ministrze. Zapraszamy. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie!

W projekcie „Planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027” przewidziano różnorodne instrumenty wsparcia dedykowane rodzinnym gospodarstwom. Analizy SWOT i diagnoza sektora rolno-spożywczego wskazały na duże potrzeby związane z zapewnieniem odpowiednich dochodów gospodarstw rolnych, a także na potrzebę budowania odporności i konkurencyjności tych gospodarstw.

Wsparcie inwestycyjne będzie realizowane w ramach interwencji pod nazwą „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” Zakłada się, że celem interwencji będzie zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność gospodarstw poprzez racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji, zmianę profilu produkcji, poprawę jakości produkcji, zwiększenie wartości dodanej produktu. W ramach interwencji możliwa będzie realizacja operacji polegającej na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji zwierzęcej z wykorzystaniem nowych technologii oraz realizacja operacji w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną. Inwestycje będą musiały doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie. Ponadto w projekcie planu strategicznego dla WPR przewidziano realizację interwencji „Premia na rozwój małych gospodarstw” Ona w tej chwili również jest realizowana. Celem ww. interwencji jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, w szczególności poprzez powiązanie produkcji ze sprzedażą, upowszechnianie krótkich łańcuchów, zmianę profilu produkcji, poprawę jakości produkcji. Dodatkowo planuje się, że premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w wyniku którego powinien nastąpić wzrost orientacji rynkowej gospodarstwa wyrażony w szczególności w osiągnięciu określonego wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. O pytanie dodatkowe poproszę panią poseł Teresę Pamułę. Panie Ministrze! Wiemy, że produkcji żywności w Polsce jest coraz więcej, o czym świadczy również eksport produktów rolno-spożywczych.

Głównymi partnerami są nadal kraje Unii Europejskiej. W 2020 r. wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych na unijny rynek wzrosła o 5% - do 27,2 mld euro, co daje 80% przychodów z eksportu towarów żywnościowych. Pozostałe kraje, czyli Rosja, Ukraina, Arabia Saudyjska to 20%.

Panie ministrze, bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest promowanie polskiej żywności zarówno na rynku krajowym, jak też na rynkach zagranicznych. Celem prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w tym obszarze jest zwiększenie konkurencyjności polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległy mu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizują wspólną, dynamiczną i ukierunkowaną politykę promocji produktów żywnościowych dostosowaną do aktualnych potrzeb sektora rolno-spożywczego. Resort rolnictwa wdraża spójne działania informacyjne i promocyjne dotyczące polskiej żywności o wysokiej jakości oraz polskich produktów, w tym produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ich przetworów, które mają na celu przede wszystkim kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności w kraju, na rynkach Unii Europejskiej i rynkach krajów trzecich, zwiększanie rozpoznawalności marki polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, zwiększanie wartości eksportu, w tym dywersyfikacja i otwieranie nowych rynków zbytu ze szczególnym uwzględnieniem rynków państw trzecich o największym potencjale wzrostu. W celu kreowania pozytywnego wizerunku polskiej żywności, a także zwiększania konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego ministerstwo rolnictwa oraz KOWR realizują m.in. działania mające na celu promocję produktów rolno-spożywczych przez organizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń wystawienniczo-targowych. Dzięki temu zarówno w kraju, jak i za granicą budowana jest silna i rozpoznawalna marka polskiej żywności. W kraju pod jednym hasłem „Kupuj świadomie” prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne dotyczące oznaczenia „Produkt polski”, rolnictwa ekologicznego, znaku „Poznaj dobrą żywność”, unijnych znaków: „Chroniona nazwa pochodzenia”, „Chronione oznaczenie geograficzne” i „Gwarantowana tradycyjna specjalność”, a także „Integrowana produkcja roślin”, [[Dzwonek]] oraz oznaczenia przez GMO - „Wyprodukowano bez stosowania GMO” Ta kampania skierowana jest do krajowego odbiorcy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jednostka nadzorowana przez ministerstwo wdraża instrumenty polityki promocyjnej także w sektorze rolno-spożywczym. Oferta KOWR-u jest dla wszystkich branż tego sektora. Promujemy też akcję „Kupuj świadomie” Znaczny nacisk położony jest tutaj na działania w obszarze oznaczenia „Produkt polski” w związku z koniecznością wsparcia wewnętrznego popytu na krajowe produkty rolno-spożywcze oraz rolnictwa ekologicznego w związku ze strategią Europejski Zielony Ład. Ponadto ministerstwo organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego m.in. celem omówienia i przedstawienia planowanych działań informacyjno-promocyjnych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, panie ministrze. Przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Mariusz Trepka i Waldemar Andzel z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zadadzą pytanie w sprawie programu „Moja woda” Odpowiedź będzie ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Ireneusz Zyska. Bardzo proszę, panie pośle. Pan poseł Mariusz Trepka ma głos. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Program „Moja woda” to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczenie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać do 5 tys. zł. Wiemy, że wielu właścicieli domów już z tego skorzystało. To jest bardzo cenna inicjatywa. Panie Ministrze! Chciałbym się dowiedzieć, ile wniosków i na jaką kwotę wpłynęło w tym roku do wojewódzkich funduszy, jaki budżet został przeznaczony na obecny, już drugi nabór do programu „Moja woda” oraz do kiedy można składać wnioski w ramach obecnego naboru. Myślę, że ta inicjatywa jest bardzo cenna, będzie kontynuowana w następnych latach i wielu mieszkańców domów z tej „Mojej wody” skorzysta, podlewając ogródki czy działki przy swoich domach - a w ten sposób będzie też ta oszczędność i ogródki będą piękne - deszczówką, którą zatrzymają przy swoich posesjach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze, ma pan głos. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Bardzo dziękuję za to pytanie. Chcę powiedzieć, że program retencjonowania wody, który został uruchomiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku, osiąga bardzo dobre rezultaty i jest niezwykle potrzebny. Otóż, szanowni państwo, program „Moja woda” ma na celu właśnie zwiększenie retencjonowania wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, jak też zwiększenie właściwego wykorzystania wód w okresach suszy. Stąd też pan Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, realizując szeroki program polityki klimatyczno-energetycznej w zakresie swojego resortu, zainicjował wielki program „Miasto z klimatem”, ale także program budowy infrastruktury zielonej i infrastruktury niebieskiej w miastach, a także na obszarach wiejskich.

Proszę państwa, te wnioski są weryfikowane przez służby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpowiadając na pytanie, może też powiem, szanowni państwo, że w roku 2020, roku ubiegłym, budżet tego programu był nieco większy, bo program spotkał się z niesłychanie wielkim zainteresowaniem beneficjentów.

Warunki uzyskania dofinansowania: maksymalnie do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów realizacji projektu.

Wnioski w tym roku można składać do 10 czerwca drogą elektroniczną, z podpisem elektronicznym.

Jeżeli wcześniej zostanie wyczerpany budżet 100 mln zł, to te wnioski, które wpłyną, niejako nie zostaną rozpatrzone czy uwzględnione w budżecie, który mamy określony na ten rok. Z uwagi na to, że jest to program wieloletni, one uzyskają dofinansowanie w kolejnym roku, po uruchomieniu kolejnej edycji. Tak że, szanowni państwo, panie pośle, bardzo dziękuję za to pytanie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę pana posła Waldemara Andzela o pytanie dodatkowe. Miałem napisane, że pan poseł Andzel, ale coś. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę informację.

Jeszcze zostało 18 mln, można powiedzieć, tak?

I mam nadzieję, że po 2024 r. ten program będzie kontynuowany, bo naprawdę to jest duża oszczędność wody, której nam brakuje. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana ministra. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie pośle, akurat nie dysponuję dzisiaj informacją szczegółową o alokacji środków w województwie śląskim - tutaj deklaruję, że taką informację przekażę panu posłowi na piśmie - natomiast chcę przy okazji powiedzieć też o bardzo ważnym problemie, z którym stykamy się przy okazji realizacji tego programu.

Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju o wydanie wiążącej interpretacji w tym zakresie. Mam nadzieję, że w tej nowej edycji w tym roku z takimi przypadkami obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie będą musieli się borykać. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję za zadanie pytania. Przechodzimy do następnego pytania. Otóż posłanki Urszula Zielińska i Klaudia Jachira zadadzą pytanie w sprawie pomysłów rządzących na prywatyzację polskich lasów. Odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Edward Siarka. Bardzo proszę panią posłankę Klaudię Jachirę o zabranie głosu i zadanie pytania. Panie Przewodniczący Komitetu Kaczyński! Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W związku z pracami nad poselską nowelizacją ustawy o lasach pozwalającą na zamianę gruntów, także tych cennych przyrodniczo, będących w zarządzie Lasów Państwowych na inne tereny, niższej jakości, chciałabym spytać pana ministra, jaka jest opinia odnośnie do tego projektu ustawy. Jak pan ocenia fakt, że posłowie składają ustawę, potem nagle z niej się wycofują, a potem, wczoraj, składają poprawki na ostatnią chwilę, które i tak niewiele zmieniają, i za chwilę będziemy w komisji nad nią pracować? Czy ministerstwo widzi zagrożenia płynące z zaproponowanych zmian? Czy chcemy doprowadzić do tego, że zamiast lasów będziemy mieć fabryki, kopalnie albo wysypiska śmieci? I wreszcie czy nie obawiacie się, że otworzy to furtkę do cichej prywatyzacji lasów, kawałek po kawałku? Poza tym jak to możliwe, że pracujemy nad dokumentem, który traktuje las jak każdy inny teren inwestycyjny, nie zważając na aspekt przyrodniczy, zniszczenie bioróżnorodności, przerwanie korytarzy ekologicznych pozwalających na migracje zwierząt, i pana ministerstwo, które ma przecież chronić przyrodę, a nie ją niszczyć, na to nie reaguje? W projekcie jest napisane, że będą to inwestycje służące ochronie powietrza, ale czy naprawdę ktoś uwierzy, że będziemy wycinać starodrzew, żeby poprawiać jakość powietrza? Czy pan minister wie, dlaczego w takim tempie przeprowadza się tak niebezpieczne zmiany? Są proponowane jako projekt poselski, bez możliwości konsultacji społecznej, z negatywną opinią leśników, „Solidarności”, NGOs. Jakie inwestycje są tak pilne? Komu i gdzie konkretnie obiecaliście tereny leśne, że tak się spieszycie, [[Dzwonek]] by w świetle prawa uwłaszczyć się na państwowym? Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, czas na konkrety. Zapraszam pana. Wysoki Sejmie! Należy stwierdzić, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o lasach szczegółowo regulują kwestie dotyczące obrotu gruntami leśnymi. Jest temu poświęcony cały rozdział zatytułowany: Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych. Ustawa ta i zapisy tego rozdziału przewidują szereg rozwiązań prawnych i instrumenty uprawniające Lasy Państwowe do rozporządzania i gospodarowania lasami będącymi w zarządzie, a mówimy tutaj rzeczywiście o dobru narodowym.

Rzeczywiście Lasy Państwowe zarządzają 30% powierzchni naszego kraju. Rozdział ten kształtuje również całą sytuację prawną, w której zarząd nad lasami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Uprawnienia w zakresie rozporządzania tym mieniem obejmą zarówno sytuacje związane z nabywaniem, jak i ze zbywaniem nieruchomości. W tym miejscu chciałem przypomnieć kilka ważnych kwestii, które związane są właśnie z obrotem tymi nieruchomościami. Uprawnienia Lasów Państwowych to przede wszystkim nabywanie lasów i gruntów, gdy jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza to interesu Skarbu Państwa. Ostatnio zostało do tego uprawnienia dopisane również prawo pierwokupu gruntów, które są zbywane przez osoby fizyczne. Lasy Państwowe również z tego uprawnienia w ostatnich latach korzystają.

W wyniku tego nabyto grunty o powierzchni prawie 400 ha. Ustawa reguluje również kwestię sprzedaży gruntów i innych nieruchomości w ściśle określonych przypadkach. Jeżeli idzie o zbywanie nieruchomości leśnych, które stanowią własność Skarbu Państwa, to zbywanie odbywa się tylko wtedy, kiedy mówimy o pozbywaniu się, zbywaniu współwłasności czy jeżeli regulowana jest granica polno-leśna lub kiedy nadleśniczy stwierdzi, że dana nieruchomość leśna ze względu na jej charakter jest zbędna dla gospodarki leśnej, a nabywca chce ją pozyskać z tytułu ważnych interesów społecznych czy gospodarczych. Oczywiście grunty przekazywane są też krajowemu ośrodkowi wsparcia w sytuacjach, kiedy mamy grunty leśne w jakichś dużych obszarach rolnych i te enklawy leśne nie do końca spełniają warunki do tego, aby prowadzić tam racjonalną gospodarkę leśną.

Każdy z nas widzi, jak dużo linii energetycznych, linii gazowych jest umieszczonych na terenach leśnych. Również z tego tytułu lasy ponoszą bardzo duże koszty związane z lokalizacją linii energetycznych czy gazowych. Wreszcie chcę powiedzieć, że duże obszary lasów przekazywane są w wyniku ustawy jednostkom wojskowym, ale najpoważniejsze wyzwanie, które stoi przed lasami, to przekazywanie gruntów pod budowę dróg krajowych i autostrad. Niewiele osób w kraju wie, że wiele tysięcy hektarów jest związanych z budową dróg, jest przekazywanych pod budowę dróg. Te grunty są po prostu przekazywane za darmo. W świetle tego, co państwo mówicie, iż procedowana jest ustawa poselska, w tej chwili trudno jest do niej się odnosić, dlatego że zawiera ona szereg poprawek. Dziękuję, panie ministrze. O pytanie dodatkowe poproszę panią posłankę Urszulę Zielińską, Zieloni. Pan przez 5 minut lał wodę, a wody w kraju mamy mało, więc ja proszę: konkretnie, przestańmy owijać w bawełnę. Ten projekt jest po to, żebyście mogli wyciąć w pień tysiące hektarów lasu, zalać to betonem i oddać pod inwestycję za bezcen i z naruszeniem, panie ministrze, interesu państwa, właśnie z naruszeniem interesu państwa w wielu aspektach. Wiemy, że na pierwszy ogień pójdzie 240 ha lasu w Jaworznie pod budowę fabryki Izery. To piękna kampania wizerunkowa dla pierwszego polskiego samochodu elektrycznego, panie ministrze. W kraju, w którym dziesiątki tysięcy osób umierają z powodu smogu, wyrżnąć kilkaset hektarów lasu pod samochód. Gratulacje! Wtedy może okazałoby się, że do jej lokalizacji da się wykorzystać tereny pokopalniane. Zabrze, są przykłady. Ale może macie w planach kolejne takie inwestycje. Jakie konkretnie inwestycje macie państwo w planach? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana ministra. Wysoki Sejmie!

Odnosząc się do tego przedłożenia poselskiego, chcę wyraźnie powiedzieć, że wszystkie obecnie obowiązujące instrumenty prawne, które są w ustawie o lasach, i te, które tworzone są przez rząd Zjednoczonej Prawicy, nie mają możliwości, nie dają takiej możliwości, żeby dochodziło do jakiejkolwiek prywatyzacji. Po prostu jest to niemożliwe na gruncie obowiązującego prawa i mam nadzieję, że tak również będzie. Czasami jest tak, że odpowiedzi nie satysfakcjonują pytających, ale taka jest sytuacja w demokracji. Następne pytanie będą zadawali. Następne pytanie będą zadawali posłowie Tadeusz Tomaszewski oraz Paweł Krutul z klubu parlamentarnego Lewica. Będzie to pytanie w sprawie planowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji niekorzystnych zmian prawnych w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych jako jednostek ochrony przeciwpożarowej zawartych w projekcie ustawy z dnia 26 kwietnia 2021 r. o ochotniczej straży pożarnej. Odpowiadał będzie pan minister Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Panie Komendancie! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło konsultacje dotyczące nowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. I dziś chcę, aby pan minister zechciał nam odpowiedzieć, odpowiedzieć rzeszy prawie 700 tys. strażaków zrzeszonych w 16,5 tys. ochotniczych straży pożarnych, gdzie na zasadzie partnerstwa między OSP, Państwową Strażą Pożarną i gminą 4,5 tys. z nich służy w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ustawodawca proponuje, szanowni państwo, podział tego pięknego zbioru ludzi szlachetnych, walczących ramię w ramię z państwowcami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o życie, zdrowie oraz mienie ludzi. Mówi o tym w art. 15 ust. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Do tej pory jednostkami ochrony przeciwpożarowej są ochotnicze straże pożarne.

Natomiast pozostałe 12 tys. będą zwykłymi stowarzyszeniami, w których ochotnicy, uwaga, będący nawet ratownikami, spełniający kryteria ustawy, mający wyszkolenie itd., itd., którzy dzisiaj [[Dzwonek]] biorą udział w akcjach ratowniczych, nie będą mieli uprawnień przewidzianych w ustawie. A więc nie będą mieli prawa do rekompensaty pieniężnej za czas niezdolności do pracy, świadczenia ratowniczego, ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, środków ochrony i umundurowania. Znosi się też zapisy, które zobowiązują dzisiaj gminę do obowiązku ponoszenia kosztów umundurowania ochotniczych straży pożarnych, finansowania ich gotowości. Wszystko to traktujemy jako element konsultacji. Mam nadzieję, że w wyniku tych konsultacji doprowadzimy do takiej sytuacji, że ochotnicze straże pożarne nadal będą jednorodnym systemem zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, proszę bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Chciałbym panu, panie pośle, bardzo podziękować za to pytanie, bo uważam, że to jest właśnie moment, żeby przeciąć te wszystkie spekulacje. Część ludzi, polityków, którzy wiele, wiele lat obiecywało złote góry strażakom, dzisiaj, kiedy zobaczyło tę ustawę, chce ją skompromitować. Szanowny panie pośle, chciałem panu powiedzieć, że głównym celem tej ustawy jest wprowadzenie oczekiwanych od dawna dodatków emerytalnych dla ratowników OSP, [[Oklaski]] dla strażaków, którzy przez 25 lat ratowali życie, zdrowie i mienie ludzkie. To jest główny cel. Obiecywano im to od dawna. My chcemy to zrealizować. Druga rzecz. Mówi pan o podziale środowiska. To jest ten podział czy go nie ma? Jakiś jest.

Obecny tutaj komendant główny PSP jeździ po województwach, powiatach, rozmawia. Byliśmy na Mazowszu, Podlasiu, pojedziemy do Wielkopolski, panie pośle, do pana. Wszędzie rozmawiamy, słuchamy i przedstawimy raport z tych konsultacji. Pokażemy, co chcą ochotnicy. Chciałbym podkreślić, że niektóre środowiska są przerażone tą ustawą, bo wreszcie zrozumiały, że ktoś jest w stanie spełnić ich obietnice.

To jest główny cel tej ustawy. Nie, my to spełnimy, bo my dotrzymujemy słowa. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy pracować w Sejmie nad tą ustawą. Pana uwagi są cenne, będziemy się im przyglądać, będziemy je omawiać. Jestem przekonany, że pan jako ochotnik na pewno będzie miał duży wkład w dobrą jakość tej ustawy. Jestem przekonany, że zagłosuje pan za tą ustawą. Chciałbym przeciąć wszystkie wątpliwości.

Jeżeli ochotnicy powiedzą, że chcą mieć w ustawie napisane, że to ma być formacja umundurowana, to my to napiszemy, chociaż nigdzie nie zakazujemy tego, panie pośle.

Jeśli pan poseł pozwoli, mówił pan minutę za długo, ja jeszcze nie dokończyłem. Panie ministrze, przepraszam pana bardzo, że się wtrącę, ale o tym, czy ktoś mówi za długo czy nie, decyduje marszałek Sejmu. Jak pan będzie mówił za długo, to też panu pozwolę. Natomiast mam nadzieję, że zwrócił pan uwagę, że ani razu nie przerwałem panu posłowi, czego nie można powiedzieć o zachowaniu pana posła. Ale wracam do jakże ciekawego tematu. To ustawa, która docenia strażaków ochotników. To ustawa, która wprowadza po raz pierwszy legitymację. Na podstawie legitymacji minister spraw wewnętrznych i administracji może osobie legitymującej się legitymacją strażaka OSP wykupić np. zniżki komunikacyjne. Ta ustawa daje ministrowi takie prawo. Nigdy czegoś takiego nie było. Ta ustawa jest o przywilejach dla strażaków, nie o zakazach dla strażaków. Jestem przekonany, panie pośle, że w toku prac parlamentarnych wyjaśnimy sobie wszystkie wątpliwości i zagłosuje pan tak, jak powiedziałem, za tą jakże dobrą i długo oczekiwaną przez środowisko ustawą. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Paweł Krutul, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Komendancie! Wysoka Izbo!

Tak że klub Lewicy jest za dobrymi poprawkami, na pewno będzie głosował. Tak jak powiedział przed chwilą poseł Szczepański, zagłosujemy zgodnie z własnym sumieniem. Tak że klub Lewicy na pewno to poprze. Właściwie dodatkowego pytania nie było, ale ma pan, panie ministrze. To niech mnie też pan pozwoli mieć swoje zdanie w tej sprawie, dobra? My na Lewicy tak robimy, że robimy to, co uważamy za stosowne i ważne, i sami o tym decydujemy. Proszę bardzo, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Pozwolę sobie skomentować to wystąpienie pana posła i podziękować mu za to. Ja jestem przekonany, że cały parlament zagłosuje za tą ustawą, bo to będzie dobra ustawa i to będzie ustawa, której de facto twórcami są ochotnicy. Rozmawiamy z nimi codziennie, konsultujemy z nimi, słuchamy ich, przyjmujemy ich postulaty. To będzie ustawa, która wzmocni ruch ochotniczych straży pożarnych w Polsce. Bardzo dziękuję za tę deklarację poparcia i pracy nad tą ustawą.

Jakbym mógł prosić pana posła Tomaszewskiego, jest pan minister, spotkajcie się na chwilę i pogadajcie, bo widzę, że pan ma konkretne pytania co do dokładnie jednego czy drugiego zapisu. Tak że Tadeusz, jest pan minister. Pan minister nie boi się posła.

Proszę państwa, przechodzimy do następnego pytania. To dojdzie do spotkania, może będziemy więcej wiedzieli. Proszę państwa, przechodzimy do następnego pytania. Posłowie Andrzej Grzyb, Stefan Krajewski i Jarosław Rzepa z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska mają pytanie w sprawie wzrostu cen paliw, do prezesa Rady Ministrów. Na to pytanie odpowiedzą podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Jan Sarnowski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Rafał Weber. Bardzo proszę pana posła Andrzeja Grzyba. Proszę bardzo, panie pośle. Dziękuję, panie marszałku. W istocie, podobnie jak w sprawach ochotniczych straży pożarnych i tej noweli ustawy, tak również w sprawie rosnących cen paliw docierają do nas liczne interwencje ze strony obywateli, którzy pytają, jakie są przyczyny tak istotnego wzrostu cen paliw.

Jednocześnie pan prezes Narodowego Banku Polskiego, pan prezes Glapiński, stwierdza: Inflację podbijają czynniki, które są poza zasięgiem NBP-u i polityki pieniężnej, a zwłaszcza wzrost cen paliw oraz cen żywności.

Są również epidemiczne zjawiska, chociażby grypa ptasia. To wszystko sprawia, że one bardzo istotnie rosną. Opłaty dodatkowe w cenie litra np. benzyny to jest prawie 60% dodatkowych opłat.

Zatem pytam jeszcze raz: Czy rząd rozważa w tej sprawie jakieś elementy, które pozwolą na obniżenie cen paliw? Tak jak powiedziałem - czy akcyza, czy VAT, czy rezygnacja z okresowej opłaty paliwowej, czy inne elementy, które m.in. są kosztotwórcze w tej cenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana ministra. Proszę bardzo. Czyli jako drugi. Pan minister. Proszę. Przede wszystkim chciałbym gorąco podkreślić: ceny detaliczne paliw należą do kategorii cen umownych ustalanych przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe.

wątpliwości, pamiętajmy: kwotowe stawki akcyzy na olej napędowy i benzyny silnikowe nie były podwyższane od bardzo długiego czasu, odpowiednio od roku 2012 - to już jest 9 lat - i od roku 2007 - to już nawet więcej. Tak że polityka podatkowa rządu w stosunku do tych paliw i do tego obciążenia nie jest pod żadnym pozorem przyczyną wahań poziomu cen tych paliw. Powiem więcej: wysokości stawek akcyzy wraz z opłatą paliwową na benzynę i olej napędowy należą do najniższych w Unii Europejskiej. Kształtują się na poziomie minimów dopuszczalnych prawem wspólnotowym. Patrząc również na ceny - według danych za maj 2021 r. benzyna silnikowa była tańsza jedynie w Bułgarii i w Rumunii, olej napędowy był tańszy jedynie w Bułgarii, w Rumunii i na Litwie. Ewentualne obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe nie będzie jednoznacznie równało się obniżeniu cen detalicznych. Obniżka akcyzy może być przechwycona przez producentów, dystrybutorów i już mieliśmy z tym do czynienia w roku 2005, kiedy próbowaliśmy robić taki ruch.

Tak że pojawia się pytanie, czy nas na to w tej sytuacji stać.

Najprawdopodobniej nic, ponieważ według prognoz Ministerstwa Finansów wzrost gospodarczy w tym roku będzie sięgał ok. 3,8%, w przyszłym - 4,3%, a to jeszcze bez wpływu KPO. Dzięki pieniądzom z tego źródła wzrost powinien przyspieszyć jeszcze o dodatkowe 0,5 punktu procentowego albo i więcej.

Co do opłaty paliwowej - poproszę pana ministra. Dziękuję serdecznie.

Jeżeli chodzi o opłatę paliwową, to jest to główny składnik wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, a Krajowy Fundusz Drogowy służy do tego, aby realizować najważniejsze, strategiczne wręcz inwestycje drogowe, które polegają na budowie dróg szybkiego ruchu, autostrad i dróg ekspresowych. Tak że jeżeli ktoś wzywa do tego, aby czasowo zawiesić czy obniżyć opłatę paliwową, to de facto wzywa do wycofania tych inwestycji, do niebudowania dróg szybkiego ruchu, do niebudowania obwodnic w ciągach dróg krajowych, bo Krajowy Fundusz Drogowy właśnie do tego służy. Przypomnę, szanowni państwo - zresztą o tym mówił pan minister Jan Sarnowski - że ostatnie podwyżki czy to akcyzy, czy to opłaty paliwowej miały miejsce odpowiednio w 2010 i 2012 r. Wtedy nie słyszałem z państwa ust jakiejś wielkiej troski o to, że Polacy za paliwo muszą płacić bardzo dużo, a najwyższe koszty paliwa w ostatnich 10 latach to styczeń i luty 2012 r. Akurat pewnie przypadkowo tak się zbiegło, że byliśmy po wyborach, druga kadencja waszej koalicji dopiero się rozpoczynała i być może faktycznie było to pokłosie słów Donalda Tuska, który w rozmowie z ówczesnym prezesem Orlenu powiedział, że po wyborach paliwo może być i po 7 zł za 1 l. Tak że reasumując, nie podnosimy opłaty paliwowej, nie będziemy też jej obniżać z tego względu, że zależy nam na tym, aby inwestycji infrastrukturalnych, inwestycji drogowych, budowania, łączenia brakujących odcinków autostrad, budowania dróg ekspresowych było w Polsce jak najwięcej, i będzie jak najwięcej. Dziękuję serdecznie.

Panowie Ministrowie!

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Ale w 2011 r. to prezes Kaczyński mówił, że można obniżyć te opłaty, żeby cena paliwa była niższa.

Dziękuję. Proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, szanowni państwo, że ustaliliśmy jedno: za rządów Prawa i Sprawiedliwości opłata paliwowa nie wzrosła, a akcyza została obniżona. To jest fakt, który miał miejsce. To za waszych rządów zostały podniesione i akcyza, i opłata paliwowa.

Minimalne wynagrodzenie w roku 2011 to 1386 zł, średnie wynagrodzenie to 3400 zł. W 2021 r., kiedy paliwo jest w podobnej cenie, minimalne wynagrodzenie to 2800 zł, a średnie wynagrodzenie to 5200 zł. Tak że nie mówcie, szanowni panowie, że dzieje się coś złego na rynku paliw, bo się nie dzieje.

Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do następnego pytania. Poseł Waldemar Andzel oraz posłanka Barbara Bartuś. pani poseł Barbara Bartuś. z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zapytają się, pytanie będzie w sprawie porównania polskiego Krajowego Planu Odbudowy z planami obowiązującymi w innych państwach oraz środków dla województw śląskiego i małopolskiego. Odpowiadał będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pan minister Waldemar Buda. Bardzo proszę, pierwsze pytanie zadaje pan poseł Waldemar Andzel, a drugie pytanie będzie zadawała pani poseł Barbara Bartuś. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Premier Mateusz Morawiecki wynegocjował gigantyczne środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski, to jest 23,9 mld euro w formie grantów oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek. Według obliczeń Komisji Europejskiej Polska jest na trzecim miejscu jako beneficjent funduszu naprawczego Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać, które z państw członkowskich otrzymają równie wysokie wsparcie, a które relatywnie niewielkie. Po drugie, jakie środki otrzyma województwo śląskie w tym podziale? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie ministrze. Tak sobie myślę, panie pośle, że jeżeli Polska jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, to wszystkie państwa, które są poniżej trzeciego miejsca, dostały mniej. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Dziękuję, panie pośle, za to pytanie.

Elementy negocjacyjne miały tu bardzo duże znaczenie.

22 kraje ratyfikowały decyzję Rady o systemie zasobów własnych, która umożliwia uruchomienie tych środków, a dokładniej pozyskanie środków na rynkach finansowych.

Jeżeli dzisiaj samorządowcy pytają, kiedy będą środki, to ja mogę powiedzieć tylko, że będą miesiąc później.

Chyba nikomu nie zleży na tym, żeby tych środków nie było albo żeby ich przekazanie się opóźniło. Tym bardziej, że system, to też jest wynikiem zabiegów pana premiera, jest tak zbudowany, żeby bardzo szybko uruchomić środki.

To jest kwota wspólna dla całego kraju. Jest 5 komponentów i w ramach tych komponentów będą realizowane konkursy.

To jest najwyższa w Polsce alokacja.

Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe zada pani poseł Barbara Bartuś. Proszę bardzo.

Natomiast chciałabym dopytać o te środki, które popłyną. Środki, w tym środki unijne, płyną do nas od dawna i budzą wiele emocji: dlaczego ktoś dostaje, a ktoś nie dostaje.

I jeszcze jedno: Na co te środki będzie można przeznaczać?

Bez pomocy zewnętrznej samorządy tego nie udźwigną. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Największym zarzutem kierowanym wobec obecnego rządu, jeśli chodzi o dysponowanie środkami na inwestycje, zarówno europejskimi jak i krajowymi, jest zarzut odejścia od polityki dyfuzyjno-polaryzacyjnej, czyli od polityki, która koncentrowała się na założeniu, że wzmacnianie dużych ośrodków przyniesie ostatecznie spójność terytorialną i rozwój całej Polski. Efekty tego możemy przejrzeć w danych statystycznych: GUS-owskich, Eurostatu, które pokazują budowanie coraz większej rozpiętości między bogatszymi a biedniejszymi regionami, między miastami a regionami wiejskimi, obszarami wiejskimi.

To budzi wiele emocji, dlatego że przyzwyczajenia były inne.

Proszę mi wierzyć, że przy konstruowaniu założeń Krajowego Planu Odbudowy mieliśmy na względzie właśnie uwzględnienie małych miast, których problemy wykluczenia komunikacyjnego, albo też w zakresie służby zdrowia, braliśmy pod uwagę. Ale trzeba też powiedzieć o rozmowach z Lewicą, która również zwracała nam uwagę na to, żeby koncentrować się na problemach chociażby zdrowotnych w małych ośrodkach, i to też trzeba docenić.

Dziękuję serdecznie. Posłowie Izabela Leszczyna i Sławomir Nitras z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska zadadzą pytanie w sprawie planu dramatycznego zwiększenia obciążeń podatkowych i składkowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Pytanie to będzie skierowane do ministra finansów, a będzie odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan minister Jan Sarnowski. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku! Przedstawiliście państwo w zeszłym tygodniu Nowy Ład.

A ludzie się tych rozwiązań boją, bo uważają, że z całego Nowego Ładu, z tych wszystkich obietnic zostanie tylko jedna rzecz: podwyżka podatków. Najbardziej boją się tego przedsiębiorcy. Najbardziej boją się tego przedsiębiorcy samozatrudnieni. Boją się, że wprowadzicie nowy 9-procentowy podatek, który zapowiedzieliście.

Dlaczego polska gospodarka mogła latami się rozwijać? Dlatego że polscy przedsiębiorcy mieli dwie rzeczy: po pierwsze, byli przedsiębiorczy, pod drugie, Polska proponowała im niskie, proste podatki. Uważacie, że wyjście z COVID-u, który przetrwaliście dzięki przedsiębiorcom. To polski eksport, polscy przedsiębiorcy uratowali budżet. To nie jest wasza zasługa, to jest zasługa przedsiębiorców. Co dostają w zamian? Drastyczną podwyżkę podatków. Będziecie uszczelniać, ale oni znajdą furtkę. Pan Kaczyński obiecał nam kiedyś europejskie zarobki, a wprowadził nam europejskie podatki. Proszę zwrócić uwagę, że przy podatkach. W Niemczech za 6 tys. zł, za 1300 euro nie płaci się żadnych podatków, jest zwolnienie z PIT, a u nas za te same kwoty płaci się 30%. Chcecie, żeby przedsiębiorcy płacili 30% podatków. Charakterystyczne, że pan Morawiecki, który przepisał praktycznie cały swój majątek na żonę, latami jako prezes banku nadużywał tego systemu. System dla fryzjerów, dla kosmetyczek, dla kierowców transportowców wykorzystywał prezes banku. Mógł mieć umowę o pracę. Wykorzystywał system.

W ten sposób zarżniecie polską gospodarkę. Oczekuję od państwa tutaj pełnej informacji dotyczącej wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, szczególnie samozatrudnionych, po wprowadzeniu tzw. Nowego Ładu. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, panie ministrze.

Jesteśmy teraz u progu jednej z największych obniżek podatków obserwowanych w ciągu ostatnich dwóch dekad i całkowicie zadziwiające jest to, że jest to podsumowywane przez państwa posłów jako ogromna podwyżka. Już teraz efektywna stawka podatku ogółem w Polsce jest zdecydowanie niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej i w innych krajach naszego regionu.

Przeciwnie, pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie, czego efektem jest relatywnie wyższe opodatkowanie osób mniej zarabiających. Szanowni państwo, przede wszystkim obniżka podatków dla 18 mln osób.

Pani kasjerka w supermarkecie - 1800 zł rocznie. Robotnik - 1400 zł.

Jest to również pakiet, który zdecydowanie poprawi ich sytuację poprzez poprawę sytuacji na rynku pracy oraz globalnej sytuacji gospodarczej. To bardzo pozytywne zjawisko, ale przedsiębiorcom sprawia bardzo duże problemy związane z niedostatkiem rąk do pracy. Znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku to przede wszystkim ogromna zachęta do wejścia na rynek pracy.

To jest sprawdzone rozwiązanie, które sprawdziło się w wielu innych krajach świata. Pamiętajmy również, że im więcej pieniędzy w kieszeniach pracowników, tym lepsza sytuacja na rynku, tym więcej pieniędzy idzie do gospodarki, tym większy popyt, tym więcej klientów mają polscy przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że wysokość środków, które zostają przedsiębiorcy na koniec dnia, jest determinowana nie tylko stawką podatku, ale przede wszystkim szerokością bazy podatkowej i tym, przez co przemnażamy tę stawkę podatku. To jest inwestycja, a nie wydatek, i zawsze tak to rozpatrujmy. Ostatni element. Mówią państwo o Polskim Ładzie, koncentrując się tylko i wyłącznie na zmianach dotyczących składki zdrowotnej.

A ja odpowiadam, jeśli chodzi o podatki. Ulga na ekspansję i zwiększenie sprzedaży produktów, ulga na pierwszą ofertę publiczną, ulga konsolidacyjna, poszerzenie zakresu zastosowania estońskiego CIT-u, ulga w VAT dla pozyskiwania usług finansowych.

Przecież te projekty będziemy realizowali wspólnie, nie tylko z kolegami ministrami, ale również z przedsiębiorcami, z branżą doradczą... i nawet z państwem. Oczywiście. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę panią poseł Izabelę Leszczynę o zadanie pytania dodatkowego. Dziękuję, panie marszałku.

Panie ministrze, dobrobyt bierze się z pracy, z inwestycji, z przedsiębiorczości. Tymczasem po roku pandemii, po roku recesji, kiedy przedsiębiorcy liżą rany i chcą wrócić do pracy, wychodzicie i mówicie: Podnosimy wam podatki.

Proszę odpowiedzieć nam, jak macie zamiar zatrzymać lekarzy, którzy też często są na samozatrudnieniu i których brakuje. Pielęgniarki. Jak chcecie im po roku walki z COVID-em, kiedy oni ledwie żyją. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź na pytanie pani poseł. Wysoka Izbo! Chciałbym gorąco przypomnieć, że na zmianach, nawet w tej formie, która była przedstawiana w drodze szerokich założeń, zyskuje aż 40% osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

To jest właśnie to płacenie pod stołem, zatrudnianie osób za płacę minimalną. Im niższe podatki w wydolnych sekcjach dochodowych, tym mniejsza opłacalność zatrudniania tych osób za płacę minimalną i płacenia im części środków pod stołem.

Dziękuję. Posłowie Mariusz Gosek i Piotr Sak zadadzą pytania w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą w rodzinie. To pytanie jest skierowane do ministra sprawiedliwości, a odpowiadać będzie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan minister Marcin Romanowski. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Odbywa się w zaciszu domowym i z tego powodu jest trudna do wyeliminowania.

Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Rzeczywiście głównym instrumentem ustawy, o której mówimy, ustawy z 30 kwietnia ub.r., jest tzw. natychmiastowy nakaz opuszczenia przez sprawcę wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się do tego mieszkania i jego najbliższego otoczenia. Zaleta tego rozwiązania to natychmiastowa wykonalność. Wcześniej, bez tego rozwiązania, procedura wyłącznie sądowa, cywilna powodowała, że opuszczanie przez sprawcę mieszkania trwało średnio 143 dni. Obecnie to trwa między 50 a 90 minut, bo rzeczywiście natychmiastowość i prostota tego rozwiązania, stosowanego przez Policję i Żandarmerię Wojskową, jest kluczowa, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie przemocy i zwalczanie jakże szkodliwego i dolegliwego zjawiska przemocy domowej. Jeżeli chodzi o monitorowanie skuteczności tej ustawy, to już od samego początku Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło specjalne rozwiązania. Chciałbym też bardzo podziękować za działalność Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, MON-u, przede wszystkim funkcjonariuszy, bo rzeczywiście ta współpraca układa się bardzo dobrze. Monitorujemy na bieżąco sygnały pochodzące od funkcjonariuszy w związku ze stosowaniem nakazu, również ze środowiska sędziowskiego.

Jeżeli chodzi o dalszy etap, czyli postępowanie sądowe, to w omawianym czasie wniesiono do sądu 52 wnioski o przedłużenie stosowania tego środka, 6 w ubiegłym roku i 46 w tym roku. Mamy dane do końca marca, ponieważ tutaj dane zbierane są kwartalnie.

Jeżeli chodzi o skuteczność stosowania tej ustawy, to oczywiście mamy do czynienia z przypadkami łamania nakazu lub zakazu orzeczonego przez funkcjonariuszy Policji względnie Żandarmerii Wojskowej. Tutaj przewidzieliśmy postępowanie wykroczeniowe, odpowiedzialność wykroczeniową za takie przypadki. W pierwszym miesiącu było 25 takich postępowań.

Jeżeli chodzi o postępowania wykroczeniowe, to dane są zbierane w systemie półrocznym.

To też pokazuje, że to rozwiązanie działa (Dzwonek) w tym sensie, że te przypadki łamania są rzeczywiście identyfikowane, co przewidzieliśmy również w ustawie. Na koniec może ostatnie dane, które też bardzo dobrze pokazują skuteczność tej ustawy. Mianowicie osobie, w stosunku do której wydano nakaz lub zakaz, przysługuje zażalenie. Takich zażaleń w czasie obowiązywania ustawy jak na razie złożono jedynie 20 i tylko w dwóch przypadkach to zażalenie, można by powiedzieć, zostało uwzględnione, czyli ten nakaz lub zakaz został uchylony. Czyli, szanowni państwo, to oznacza, że z jednej strony mamy 1326 przypadków zastosowania nakazu i zakazu i tylko dwa przypadki, w których sąd orzekł, że właśnie ten zakaz lub nakaz był zastosowany nieprawidłowo.

Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe zada pan poseł Piotr Sak. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź i przedstawienie kompleksowych informacji i danych statystycznych. Nie chcę tutaj prawić komunałów i banałów, ale oczywistym jest, że przemoc rodzinna to poważny problem społeczny, taka anomalia w środowisku rodzinnym, bo jest przede wszystkim trudno uchwytna, z tego względu, że odbywa się w miejscu, które tak naprawdę powinno być jakimś takim swoistym asylum, taką oazą spokoju, a tak naprawdę jest miejscem niejednokrotnie gehenny i kaźni.

Dlatego też pozwolę sobie zadać pytanie panu ministrowi: Czy według ministerstwa obecny stan prawny, ten system ochrony rodziny w tej materii jest wystarczający? Czy w tym zakresie ministerstwo ma w zanadrzu jakieś nowości (Dzwonek) legislacyjne, które jeszcze bardziej wzmocnią i poprawią bezpieczeństwo? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! My przede wszystkim na bieżąco analizujemy skuteczność tych nowych regulacji, które, tak jak powiedziałem, są kluczowe, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie, bo ta skuteczność opiera się na prostocie i natychmiastowości. Rzeczywiście z tych analiz i naszych wcześniejszych zapowiedzi wynika, że w przypadku kiedy te rozwiązania zafunkcjonują, będziemy starali się rozszerzać instrumenty cywilnoprawne, bo to jest ważne, że to są instrumenty nie karne, tylko cywilnoprawne. Myślę, że ta wcześniej wskazana analiza pokazuje, że te instrumenty rzeczywiście działają, w związku z tym będziemy proponować rozszerzanie tych instrumentów właśnie wobec sprawców przemocy w rodzinie stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia członków rodziny właśnie w kierunku tej efektywnej izolacji. Mówię tutaj oczywiście o zakazie zbliżania się do osoby.

Tutaj dostrzegamy również potrzebę wprowadzania zakazu zbliżania się do osoby, ale też są innego typu rozwiązania, takie jak kwestia pełniejszego zagwarantowania osobom niepełnosprawnym intelektualnie, osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez wzbogacenie procedury karnej o jeszcze bardziej szczególny tryb przesłuchania, jeżeli zajdzie taka potrzeba, jakichś alternatywnych, wspomagających metod komunikacji. Oczywiście chodzi również o usprawnienie postępowania cywilnego w tym zakresie, a także rozstrzygnięcie różnego rodzaju wątpliwości interpretacyjnych, które siłą rzeczy w trakcie stosowania obecnych regulacji się pojawiają. Ale wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tym momencie, jeżeli chodzi o skuteczność systemu, to jest stałe nadzorowanie i doskonalenie stosowania obecnych regulacji. Tutaj jeszcze przed wejściem w życie ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości przeszkoliło 30 tys. funkcjonariuszy, kilkaset osób pierwszego kontaktu z ośrodków z Funduszu Sprawiedliwości. Tutaj też muszę powiedzieć, że miesięcznie ok. tysiąca nowych osób korzysta z pomocy Funduszu Sprawiedliwości, osób będących ofiarami przemocy domowej.

W planie mamy - właśnie są przygotowywane i prace są na finiszu - szkolenia dla kuratorów i prokuratorów wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Na koniec czerwca będziemy mieli już gotową analizę dotyczącą stosowania obecnej ustawy, co oznacza kilka tysięcy kwestionariuszy skierowanych do funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej, ośrodków pomocy społecznej oraz samych osób pokrzywdzonych.

Bardzo dziękuję. Przechodzimy do następnego pytania. Powiem panu szczerze, że wielką przyjemność mi robicie, zadając to pytanie, gdyż wczoraj toczyła się dyskusja na ten temat.

To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, w którego imieniu odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Piotr Dziadzio. I zaraz panu powiem, panie ministrze, dlaczego to pytanie sprawiło mi przyjemność. A więc jeżeli dzisiaj będziemy wiedzieli coś więcej, to będzie super. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 17 maja o godz. 16.30 10 z 11 bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów przestało wytwarzać prąd. Ubytek produkcji był znaczący, objął bowiem prawie 20% całej energii produkowanej przez elektrownie w Polsce i wyniósł 3900 MW. Przyczyną wyłączenia produkcji, jak podaje PGE, była awaria stacji Rogowiec.

Dojdą dodatkowe koszty rozruchu wyłączonych bloków, szacowne na kilkanaście milionów. Po pierwsze, czy polski system energetyczny w związku z tymi powtarzającymi się awariami jest bezpieczny? Czy polski system energetyczny jest zarządzany przez kompetentnych ludzi? Czy polski system gwarantuje gospodarstwom domowym dostarczanie prądu? Czy prąd dotrze do polskich firm? Czy polecą głowy za awarię? Bo ktoś źle odczytał wskazania na stacji Rogowiec i nie zareagował w porę, co spowodowało gigantyczne koszty. Prosimy o konkretne odpowiedzi. Jednocześnie pytam, czy Bełchatów został ujęty w planie sprawiedliwej transformacji? Bo nie ma do tej pory potwierdzenia, że tak się stało. Dziękuję serdecznie.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postaram się przedstawić państwu historię tego wydarzenia, żebyśmy powiedzieli sobie o faktach, które zaistniały, i przyczynach tak naprawdę, co jest istotne, żebyśmy prowadzili dalszą rozmowę w tym zakresie.

Przechodzę do faktów.

Dokładny mechanizm zaistnienia tej sytuacji obecnie jest przedmiotem badania specjalnej komisji powołanej przez PSE.

Komisja zbada i na pewno zabezpieczy, czyli poczyni wszelkiego rodzaju starania w tym zakresie, żeby ten błąd się nie powtórzył. Jeszcze druga sprawa - co również chciałem podkreślić, żeby było to jednoznaczne - z zebranych do tej pory informacji wiemy, że nie było to efektem działań podmiotów trzecich ani też żadnej aktywności w cyberprzestrzeni, żebyśmy mieli taką jasność. Krajowy system elektroenergetyczny został niezwłocznie zbilansowany przez PSE poprzez uruchomienie generacji w elektrowniach szczytowo-pompowych należących do PGE Energia Odnawialna. Te elektrownie w ciągu kilku minut od polecenia operatora przesyłowego uruchomiły swoje jednostki produkcyjne.

Pozostała część pochodziła z wirtualnej rezerwy cieplnej w pracujących elektrowniach: Ostrołęka, Kozienice, Opole, Połaniec, Turów, Jaworzno, Rybnik, Dolna Odra. Tak, z Niemiec, niewiele. W związku z tym system funkcjonował bez problemów. Dzięki tej szybkiej reakcji służb PSE stacja Rogowiec była gotowa do przyłączenia nowych bloków w ciągu godziny.

Reasumując to, co chciałem państwu powiedzieć, podsumowując, chciałbym stwierdzić, że to zdarzenie było w pewnym senesie takim testem dla krajowego systemu elektroenergetycznego. System zadziałał, wszystko pracuje prawidłowo oraz nie było zagrożenia w zakresie odłączenia odbiorców.

Dobrze? Panie pośle, bardzo proszę. Pan poseł Krzysztof Gadowski. Panie Ministrze! Oczywiście awarie się zdarzają i to jest rzecz normalna, że co pewien czas coś się może zdarzyć, ale rolą rządzących czy zawiadujących systemem jest być zabezpieczonym na takie ewentualne sytuacje.

Te bloki, tak jak pan minister powiedział, zasiliły system, właściwie uratowały nas przed tym, co nam zagrażało.

Bo dzisiaj mówimy o sieciach przesyłowych, gdzie te duże moce są podłączone do jednej sieci przesyłowej do transformatorów. Czy w tym zakresie ta polityka [[Dzwonek]] się zmieni czy nie? Czy państwo macie już konkretny projekt, żeby to zrobić? I ostatnie pytanie: Ile środków finansowych zabezpieczacie na system przesyłowy w swoim ładzie, Polskim Ładzie, który dzisiaj w Polsce mocno promuje pan premier?

Co do pytań, które. Nie potrafię teraz powiedzieć, jakie, ale to nie są takie koszty uruchomienia, które by wpłynęły na koszty ceny energii elektrycznej, w żaden sposób. To raz.

Czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji? Myślę, że nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie panu posłowi. Dobrze. Przechodzimy do następnego i ostatniego w tej rundzie pytania w sprawie planów dotyczących utworzenia koncernu multienergetycznego. To pytanie zada pan poseł Andrzej Gawron z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pan minister Maciej Małecki. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Mamy do czynienia z dużymi podmiotami, z rozpoznawalnymi markami.

Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie pana posła, w pierwszym zdaniu poinformuję, że Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN Orlen, Grupa PGNiG i Grupa Lotos potwierdziły strukturę połączenia spółek w taki sposób, aby utworzyć jeden narodowy koncern multienergetyczny. W planowanej konsolidacji wiodącą rolę będzie odgrywał PKN Orlen i dzięki temu Polska zyska silny, narodowy podmiot, który będzie konkurencyjny także na rynkach międzynarodowych. Połączenie Orlenu z Lotosem oznacza wejście do najbardziej liczących się koncernów paliwowo-energetycznych w Europie, takich jak austriacki OMV, francuski Total, brytyjsko-holenderski Shell czy hiszpański Repsol. W momencie zrealizowania wszystkich fuzji, wszystkich połączeń powstanie grupa o rocznych przychodach na poziomie 200 mld zł i zróżnicowanej EBITDA liczonej na poziomie 20 mld zł rocznie. Tak zbudowany koncern będzie miał przed sobą otwartą ścieżkę do dalszego wzrostu. I trzeba mocno powiedzieć, że konsolidacja gwarantuje wejście Orlenu do ekstraklasy firm paliwowo-energetycznych w Europie. Polska potrzebuje silnego koncernu multienergetycznego, który będzie kołem zamachowym naszej gospodarki. Koncernu, który będzie miał środki na inwestycje i który z powodzeniem będzie konkurował na zagranicznych rynkach. Chcemy mieć markę rozpoznawalną na świecie. Orlen po połączeniu z PGNiG, Lotosem stanie się polskim czempionem, polską światową marką i jednym z największych w Europie koncernów multienergetycznych. Stworzenie koncernu multienergetycznego jest konieczne z punktu widzenia wszystkich firm tworzących ten koncern, budowania ich wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz bezpieczeństwa naszej części Europy, a także interesu klientów indywidualnych i lokalnych społeczności. Dziś mamy sytuację, w której Orlen i Grupa Lotos wzajemnie ze sobą konkurują, mimo że obie spółki są w portfelu Skarbu Państwa. Takie zjawisko jest niespotykane w innych krajach europejskich. Dodatkowo konsolidacja znajduje tu silne uzasadnienie biznesowe. Polski system energetyczny, jak pan poseł raczył wspomnieć, wymaga fundamentalnej transformacji ze względu na wiek aktywów i ze względu na ambitne cele klimatyczne. Koszty transformacji to jest ponad 450 mld zł i gros zadań w tym procesie weźmie na siebie nowy, silny koncern multienergetyczny zbudowany wokół Orlenu. Ale korzyści będą też takie: większy potencjał rozwoju w kontekście oczekiwanej w dłuższej perspektywie marginalizacji branży rafineryjnej oraz wzrostu znaczenia petrochemii, rynku gazu czy OZE, wzmocnienie pozycji na europejskim i globalnym rynku, zwiększenie konkurencyjności polskiego podmiotu, dywersyfikacja przychodów i większa odporność na fazy cyklu gospodarczego. Połączony podmiot będzie oparty o w pełni zintegrowany łańcuch wartości: od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę, aż po sprzedaż detaliczną. To oznacza długoterminowe zyski dla firm oraz ich akcjonariuszy, ale też oznacza stabilne ceny energii dla polskiej gospodarki i atrakcyjny pakiet kompleksowych usług dla klientów. Patrząc na wszystkie procesy akwizycyjne, które przewidujemy, można wyobrazić sobie jeden rachunek, na którym znajdą się paliwa, gaz czy energia elektryczna. Dla klientów to jest większa wygoda, ale i oszczędność czasu. Ważne, że połączony koncern będzie miał silniejszą pozycję negocjacyjną w odniesieniu do dostawców surowców - czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Rosji. Przejęcie Lotosu przez Orlen nie spowoduje też wzrostu cen paliw na stacjach. Temat cen paliw jest bardzo wrażliwy, ale pamiętajmy o tym, że spółki nadal będą działały w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, a ceny paliw są kształtowane też przez inne zewnętrzne czynniki, przede wszystkim przez ceny surowców czy kursy walut. Optymalizacja procesów zachodzących pomiędzy tymi spółkami, wykorzystywanie synergii nie oznacza zwolnień, bo nie tu koncern będzie poszukiwał oszczędności. Nie są prowadzone żadne prace związane z redukcją zatrudnienia. Ważnym aspektem, to podkreślam, jest wzmocnienie pozycji Skarbu Państwa w akcjonariacie skonsolidowanego podmiotu. Obecnie Skarb Państwa ze względu na posiadany udział ma władztwo korporacyjne w Lotosie i PGNiG i mniejszościowy udział w Orlenie. Zwiększenie udziału Skarbu Państwa w skonsolidowanym podmiocie zwiększy władztwo korporacyjne w multienergetycznym koncernie i zminimalizuje ryzyko wrogiego przejęcia, zagwarantuje też bezpieczeństwo energetyczne Polski i umożliwi właściwe kontrolowanie strategicznych aktywów zgodnie z interesem gospodarczym Polski. Dziękuję serdecznie. Pytanie dodatkowe, bardzo proszę. Panie ministrze, mówił pan o celach. Rzeczywiście można powiedzieć, że te cele są w dalszej perspektywie pozytywne dla gospodarki, dla pracowników, co pan podkreślił, ale też dla Skarbu Państwa, który w tym ładzie korporacyjnym polepszy jak gdyby swoją pozycję, ale na pewno będzie to proces długotrwały i skomplikowany.

To są, tak jak powiedziałem, duże firmy. To są spółki Skarbu Państwa o różnym kapitale własnościowym i nie będzie to łatwe, ale myślę, że determinacja ze strony PKN Orlen jest dosyć istotna. Ministerstwo akceptuje ten proces. Tak że proszę o określenie tych poszczególnych etapów konsolidacji. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgodnie z czterostronnym porozumieniem zawartym w Ministerstwie Aktywów Państwowych połączenie zostanie zrealizowane poprzez przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos i Grupy PGNiG. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Lotosu i akcjonariusze PGNiG otrzymają nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tejże nowej struktury, tego nowego podmiotu. Połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji. Umożliwi to pełną i szybką integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia. Wygenerowane w ten sposób środki będą wspierać prowadzony przez połączony koncern program rozwojowy i transformacyjny. Konsolidacja jest procesem bardzo skomplikowanym, a harmonogram konsolidacji zależy także od decyzji administracyjnych organów antymonopolowych. I tu się toczą dwa postępowania: w sprawie konsolidacji Orlenu i Lotosu przed Komisją Europejską, a w sprawie konsolidacji Orlenu i PGNiG przed polskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie przed Komisją Europejską będzie... ta konsolidacja będzie uzależniona od dalszych decyzji Komisji co do wykonania wynegocjowanych w 2020 r. środków zaradczych. Wykonanie tych środków zaradczych przez Orlen i Lotos ma na celu zapewnienie konkurencji i ochrony konsumentów w sytuacji, kiedy obydwa podmioty będą działały łącznie.

Jego akceptacja umożliwi podjęcie dalszych czynności, w tym zaplanowanie harmonogramu odpowiednich decyzji korporacyjnych. Z kolei połączenie Orlenu i PGNiG, tak jak powiedziałem, podlega postępowaniu przed UOKiK-em. Spodziewamy się, że decyzja co do zgody na konsolidację powinna zapaść w II połowie br. I wtedy będą możliwe dalsze czynności, w tym również zaplanowanie harmonogramu odpowiednich decyzji korporacyjnych. Czyli - odpowiadając już wprost na pytanie pana posła - najbliższe miesiące będą kluczowe dla możliwości precyzyjnego określenia terminu powstania skonsolidowanego podmiotu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że intencją Skarbu Państwa jako akcjonariusza wszystkich tych spółek jest, aby zasoby majątkowe i ludzkie każdej z nich przyczyniły się do stworzenia silnego koncernu multienergetycznego o zdecydowanie większych możliwościach rozwoju. Przyjęta formuła gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej, silnej firmy, uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Zagwarantowana została wiodąca rola PKN Orlen w tej transakcji. Podkreślam: z punktu widzenia ministerstwa aktywów, polskiego rządu konsolidacja Orlenu, Lotosu, PGNiG jest korzystna dla polskiej gospodarki, dla klientów i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dziękuję serdecznie. Pytanie to kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie działań podejmowanych na rzecz seniorów, w szczególności zmierzających do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 5 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut. Bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców panią poseł Barbarę Bartuś. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Wniosek o przedstawienie informacji w sprawie działań podejmowanych na rzecz seniorów, a w szczególności zmierzających do poprawy warunków życia i aktywności społecznej osób starszych, rozpocznę od takiej ogólnej deklaracji, że problemy osób starszych powinny być rozwiązywane przez rząd, samorządy, a nie tylko spoczywać na barkach rodzin. Biorąc pod uwagę rolę seniorów w naszym społeczeństwie, ich zasługi oraz bieżące potrzeby, jesteśmy zobowiązani podejmować wszelkie możliwe aktywności na rzecz poprawy sytuacji osób starszych. Uwzględnianie w polityce społecznej spraw seniorów jest wyzwaniem i zobowiązaniem dla rządu, jest podziękowaniem dla naszych seniorów za ich dotychczasową pracę i obywatelską postawę. O tym też wielokrotnie mówiliśmy, będąc w opozycji za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wtedy też zgłaszaliśmy propozycje, postulaty, jak również gotowe projekty ustaw, które miały pomóc w sytuacji, pomóc seniorom.

Chcemy żyć jak najdłużej, ale wszyscy się starzejemy. My też jesteśmy coraz starsi, liczba seniorów w naszym kraju stale rośnie. Do końca roku 2050 będzie to najliczniejsza grupa społeczna. Dlatego jest to olbrzymie wyzwanie i olbrzymie zadanie dla rządu i całego naszego państwa, aby o tę grupę zadbać. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Ważne jest też zwrócenie uwagi na fakt, że seniorzy to grupa nie tylko liczna, ale i niejednorodna. Innych działań potrzebują młodzi seniorzy, którzy chętnie biorą udział w różnego rodzaju inicjatywach, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, a innych - osoby w wieku sędziwym, w przypadku których najczęściej najważniejsze są pomoc w codziennych czynnościach i pieniądze na leki. Trzeba też brać pod uwagę to, że znaczna grupa seniorów to samotne kobiety, wdowy, które albo nie mają dzieci, albo których dzieci mieszkają w innych miejscach, a często, tak jak na moim terenie - poza granicami kraju. Pragniemy więc, panie ministrze zapytać: W jaki sposób rząd Rzeczypospolitej Polskiej dba o interes seniorów? Które kwestie są dla rządu priorytetowe w tej szczególnej społecznej sytuacji, w odniesieniu do zmiany proporcji pomiędzy generacjami, wzrostu populacji seniorów względem pozostałych grup społecznych? Rząd ma partnerów do realizacji działań społecznych. Rośnie liczba organizacji seniorskich, wiele zadań realizują samorządy. A jeżeli tak, to jak wygląda ta współpraca z samorządami? Oczekiwania społeczne dotyczą wielu aspektów życia. Niektóre z nich są ściśle związane z bieżącymi problemami, w tym szczepieniami przeciw COVID-19, adekwatną opieką zdrowotną, sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, aktywnego starzenia się. Działania rządu na rzecz osób starszych są przewidziane w planowanych programach społeczno-gospodarczych, takich jak Polski Ład. Prosimy więc o pełną informację, jakie rozwiązania prawne i systemowe proponuje ministerstwo, jakie też programy rząd już realizuje. Dziękuję serdecznie za pytanie. Panie ministrze, bardzo proszę. Bardzo proszę o odpowiedź. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję klubowi Prawo i Sprawiedliwość za to, że wniósł o informację bieżącą dotyczącą polityki senioralnej, bardzo ważnej dla nas wszystkich, dla naszego kraju, ale również dla naszego rządu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy od samego początku bardzo mocno wspiera działania wspomagające seniorów. Oparliśmy te nasze działania na dwóch filarach. Pierwszy filar to poprawa bezpieczeństwa materialnego seniorów, a drugi filar to poprawa zarówno usług dotyczących seniorów i ich rodzin, jak i aktywizacji. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo materialne, to rozpocznę od dwóch najważniejszych chyba działań, które podejmowaliśmy w ostatnim czasie. Ale trudno nie przypomnieć najważniejszego działania, które podjęliśmy zaraz na początku naszej kadencji, czyli przywrócenia wieku emerytalnego mężczyznom i kobietom. Przypomnę: 65 lat - mężczyźni, 60 lat - kobiety. To był postulat obywatelski, był też projekt obywatelski w tym zakresie złożony przez związek zawodowy „Solidarność”, który także domagał się przywrócenia wieku emerytalnego, i to spełniliśmy.

W tym zakresie bardzo ważne działanie, które podjęliśmy, dotyczyło wzrostu najniższej emerytury.

Bardzo ważnym instrumentem, który wprowadziliśmy w życie, była tzw. trzynasta emerytura, czyli świadczenie, które już w tej chwili jest na stałe wpisane, ustawowo. Przyznaliśmy każdemu emerytowi i renciście w naszym kraju dodatkowe świadczenie w postaci najniższej emerytury. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w ciągu 3 lat funkcjonowania programu prawie 36 mld zł trafiło do naszych emerytów i rencistów, bo wszystkie grupy bez wyjątku tym programem są objęte.

Czyli to dziesięciokrotny wzrost nakładów na politykę senioralną. W tym zakresie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, warto jeszcze przypomnieć o naszym bardzo dobrym programie, jakim jest emerytura mama 4+, czyli emerytura przeznaczona dla tych mam - i ojców - które wychowały co najmniej czwórkę dzieci, a które nie nabyły prawa do świadczenia emerytalnego. Z tego rozwiązania korzysta dzisiaj ponad 71 tys. mam i nieliczna grupa ojców. Łącznie przeznaczamy na to ponad 880 mln zł. Także w stosunku do osób związanych z osobami represjonowanymi takie rozwiązanie wprowadziliśmy - dodatkowe świadczenie do kwoty 2500 zł, również jako uzupełniające świadczenie wyrównawcze. Tutaj są dwa bardzo ważne programy, które realizujemy. To jest program, który realizujemy wspólnie w ostatnim czasie.

Dzisiaj mamy ponad 1000. Czyli nastąpił olbrzymi wzrost liczby tych jednostek i z tego się cieszymy, bo seniorzy chętnie z tego korzystają - ponad 23 tys. uczestników zajęć w tym okresie.

Przez kolejne lata to jest wsparcie na poziomie 500 mln zł.

On z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem.

To jest nowe rozwiązanie, które wprowadziliśmy. Z niego korzysta w tej chwili 588 tys. osób.

Na resztę odpowiem państwu po pytaniach. Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Powiedzmy, do 1 minuty. Do 1 minuty? Półtorej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy realizuje kompleksową politykę senioralną. Seniorzy i rodzina są dla nas szczególnie ważni, co udowadniamy od momentu przejęcia odpowiedzialności za Polskę w 2015 r., dobrze realizując umowy społeczne. Przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn - to obietnica, z której się wywiązaliśmy w trybie błyskawicznym. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma imposybilizmu. My nie mówimy, że nie ma i nie będzie pieniędzy, szczególnie wtedy, kiedy trzeba realizować cele społeczne, kiedy trzeba wspierać tych, którzy tego wsparcia potrzebują najbardziej, a tą grupą są właśnie seniorzy. Świadczenia seniorów najniżej uposażonych wzrosły za naszych rządów o ponad 42%.

Bardzo cieszę się z tego, że w naszym kolejnym programie dla Polski, programie Polski Ład, w naszej strategii, nowej strategii [[Dzwonek]] dla seniorów znajduje się również kwestia emerytury bez podatku do kwoty 2,5 tys. zł.

Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rzeczywiście najniższe świadczenie wzrosło, ale nie mówicie już państwo o tym, że liczba emerytów, którzy pobierają głodowe emerytury, również drastycznie wzrosła. Na dzisiaj to jest ok. 350 tys. osób. Mówicie państwo o wzroście emerytur, ale prawda też jest taka, że jest duża inflacja. A więc za te same pieniądze można było kupić więcej produktów, niektóre nawet taniały. Dzisiaj mamy do czynienia z drożyzną. Za prąd trzeba zapłacić nawet o 14% więcej. Szanowni Państwo! Co zrobiliście z głodowymi emeryturami? Nic nie zrobiliście. Wśród tych emerytów 80% to kobiety. Niestety tak to wygląda. Mówicie państwo o opiece nad seniorami, a przecież tak naprawdę nie wprowadziliście żadnego systemu opieki nad seniorami - żadnego. Żadnej ustawy nie wprowadziliście. Mało tego, np. pieniądze, które były przeznaczone na opiekę w 2020 r., w stosunku do 2019 r. były mniejsze. Niestety tak to wygląda. Zadłużenie emerytów.

Dziękuję. Pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Rząd wspiera i finansuje tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To jest nowy typ placówki w polskim systemie. Bardzo ciekawy program, oczekiwany. On jest przeznaczony dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Realizuje się opiekę i pomoc osobom z takim właśnie stopniem niepełnosprawności w ramach albo dziennego, albo całodobowego pobytu w tych placówkach. Chciałbym zapytać pana ministra, w jakim procencie czy w jakiej liczbie już utworzone centra opiekuńczo-mieszkalne i te planowane będą świadczyły opiekę na rzecz niepełnosprawnych seniorów, niepełnosprawnych osób starszych.

Jakie są kryteria kwalifikowania tych osób do tych placówek? Czy są uwzględnione kryteria socjalne, dochodowe, wiekowe?

Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Obowiązkiem władzy publicznej jest aktywna polityka senioralna.

Pan minister mówił - jak przedstawiał swoje osiągnięcia - o wzroście o ponad 40% emerytury minimalnej. Ale dzisiaj mamy problem dotyczący 350 tys. tzw. emerytów, którzy nie mają prawa do minimalnej emerytury, czyli 1250 zł brutto. Tym problemem trzeba się zająć od zaraz, to jest kwestia godności człowieka. W tej sprawie klub Lewicy nie czeka. Złożyliśmy stosowny projekt ustawy, który jest już na stronach internetowych Sejmu. Warto do niego wrócić, warto, aby rząd chciał konstruktywnie, wspólnie z parlamentem poszukiwać rozwiązania tego problemu społecznego. Drugi problem to bieżący problem dotyczący szczepienia osób po 70. roku życia, które są niesamodzielne. Niestety nadal to nie funkcjonuje, w wielu miejscach nie odzywają się telefony i trzeba szukać innych rozwiązań. Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Nie ma pana posła.

Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ta dyskusja zazwyczaj ogranicza się do tego, co tu i teraz, co dzisiaj. Natomiast ja chciałem prosić pana ministra o kilka słów o tym, co w przyszłości, co dla kolejnych pokoleń, ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, że społeczeństwo się starzeje, emerytów będzie coraz więcej, coraz więcej osób będzie przechodziło w stan emerytalny i będzie ich znacznie więcej w stosunku do pracujących niż ma to miejsce dzisiaj. Tymczasem w parlamencie leży projekt ustawy, który przewiduje, że 15% środków zgromadzonych w OFE zostanie zagrabionych w formie takiego, powiedziałbym, podatku.

W związku z tym, panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy rząd wycofa się z tego projektu i pozostawi te środki w gestii emerytów, tak żeby one mogły pracować na emerytury kolejnego pokolenia w perspektywie (Dzwonek) wielu dziesiątek lat do przodu. Dziękuję. Nie ma pani poseł. Pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Można powiedzieć, że dzisiejszy dzień zaczyna literka „i” Najwyższa od 20 lat, w kwietniu wyniosła 5,1% rok do roku - to są dane Eurostatu. Szanowni państwo, co to oznacza? To oznacza, że emerytów czeka niewyobrażalna drożyzna. A jeżeli czeka drożyzna, to potrzebne są dodatkowe środki w portfelach emerytów. Wtedy Sejm głosował nad dwoma projektami: emerytura bez PIT-u, projekt Platformy Obywatelskiej i emerytura bez podatku, projekt PSL-u. W obydwu przypadkach 237 posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości głosowało przeciw. Przypominajmy te dane. Druga sprawa to ochrona zdrowia. Najdłuższe w historii kolejki do specjalistów. To pokazuje, że muszą wydawać na prywatne usługi medyczne, prywatne wizyty, prywatną rehabilitację. Kolejna sprawa to narodowy plan alzheimerowski. Tego programu cały czas nie ma. I ostatnia sprawa - zakłady opiekuńczo-lecznicze. Stawka, którą płaci NFZ za osobodzień, [[Dzwonek]] jest niedoszacowana na skalę 40%. Weźcie się wreszcie do roboty, bo polscy seniorzy na to liczą. Pani poseł Wanda Nowicka, klub Lewicy.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Mianowicie bardzo ważne jest, żeby na problem seniorów patrzeć nie tylko jako na problem do rozwiązania, ale również potencjał do wykorzystania. Brakuje mi tego w tym, co słyszę, że macie w ogóle takie podejście do kwestii osób starszych. Wiemy, że seniorzy to jest grupa zróżnicowana, ma różny potencjał i możliwości, ale ma właśnie potencjał. Zwłaszcza chciałabym zwrócić uwagę na potencjał intelektualny seniorów, zgromadzony przez lata kapitał wiedzy i doświadczenia powinien mieć szansę na realizację. Czy macie jakieś plany i programy, żeby pójść w tym kierunku?

Pani poseł, bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Trwająca już od roku pandemia dotknęła wszystkich. Nie ma zapewne w naszym kraju rodziny, której skutki pandemii nie dotyczą - strata bliskich, śmierć, utrata rodzinnych firm, choroba, strach. Pamiętajmy, że grupą najbardziej narażoną od początku trwania pandemii, ale i nadal są osoby starsze, schorowane, dotknięte niepełnosprawnością, które przez ten czas były często odcięte od rodziny. Mam na myśli osoby przebywające w ośrodkach i domach pomocy społecznej. Wiele z tych osób odeszło, wiele wyzdrowiało, wiele zostało zaszczepionych. W tej grupie od początku pandemii zachorowania odnotowano u ponad 80% pensjonariuszy. Panie Ministrze! Czy prowadzone są na bieżąco statystyki? Czy odpowiednio monitorowana jest sytuacja osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach dla ludzi z niepełnosprawnością? Jaka jest dzisiaj skala zachorowań? Jaki jest procent wyszczepialności? Teraz, kiedy trzecia fala poniekąd odpuszcza, tym bardziej nie możemy stracić tej czujności, jeżeli chodzi o osoby starsze, schorowane. Skutki niedopatrzenia mogą być katastrofalne. Są to wciąż środowiska bardzo wielkiego ryzyka. Dlatego pytam: Czy ta sytuacja jest na bieżąco monitorowana? Dziękuję. Pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! O obszarze społeczno-socjalnym mieliśmy okazję usłyszeć. Natomiast chciałabym wspomnieć o aspekcie zdrowotnym. Wiemy, że dobra jakość życia to dobry stan zdrowia. Dlatego chciałabym podkreślić, że te działania rządu, które były podejmowane w ostatnich latach, były nakierowane na zwiększenie liczby świadczeń udzielanych seniorom, jak również na zwiększenie finansowania.

Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Warto podkreślić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jedynym, który tak mocno wspiera seniorów. W mojej ocenie najważniejsze w szerokim spektrum działań na rzecz seniorów było wprowadzenie trzynastej, czternastej emerytury. Obecnie na pierwszy plan ochrony senioralnej wysuwają się przedstawione w zeszłą sobotę przez premiera Mateusza Morawieckiego elementy Polskiego Ładu i emerytury bez podatku.

Po wprowadzeniu zmian zyska 180 zł na rękę, finalnie otrzymując 2275 zł. Nasuwa się pytanie: Która partia zrobiła tak wielki ukłon w stronę emerytów i rencistów w czasach światowej pandemii? Przeciwnie, pandemia byłaby pretekstem do tego, by jeszcze bardziej zubożyć klasę niższą oraz pogrążyć w ubóstwie emerytów i rencistów. Dlatego chciałbym zapytać, czy rząd nadal będzie prowadzić [[Dzwonek]] wsparcie narodowego programu szczepień i jakie są rekomendacje rządu w tym zakresie. Pani poseł Paulina Matysiak, klub Lewicy. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Szczególnie interesują mnie sposoby aktywizacji społecznej seniorów, którzy dotąd izolowali się w związku z pandemią. Warto dodać, że seniorzy byli tą grupą, która była w największym stopniu odizolowana ze względu właśnie na wysokie ryzyko zakażenia i ciężki przebieg COVID-19. W tym zakresie kluczowe wydaje się przyspieszenie szczepień w tej grupie wiekowej i zachęcanie do szczepienia osób, które do tej pory tego nie zrobiły. Tu pojawia się pytanie o działania międzyresortowe, przede wszystkim działania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia w kontekście ciągle niewystarczającego wyszczepienia społeczeństwa w grupie wiekowej 60+. 2 dni temu, podczas posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej, dowiedzieliśmy się o liście ministra zdrowia do realizatorów świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Mogą oni w systemie wygenerować listy pacjentów swoich placówek z informacją na temat zaszczepienia, także z informacją o terminie umówionych szczepień. Lekarz porozmawia z tymi pacjentami, którzy jeszcze się nie zaszczepili, przedstawi korzyści płynące z uzyskania odporności przeciw COVID. Problem polega na tym, że minister Niedzielski prosi, minister Niedzielski zachęca, ale minister Niedzielski nie wymaga. Lekarze nie muszą nawet odnotować tej informacji, którą uzyskają podczas rozmowy. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, by realnie zwiększyć liczbę zaszczepionych seniorów? Bardzo proszę. Panie Ministrze! Rada Ministrów w październiku 2018 r. przyjęła dokument: Polityka społeczna wobec osób starszych z perspektywą 2030. Po 3 latach myślę, że warto zapytać o realizację tego dokumentu. W tym dokumencie sformułowano pięć programów celowych, tzw. priorytetowych. Chciałbym prosić o odpowiedź na pytanie o realizację przynajmniej dwóch tych priorytetów. Mianowicie pkt 4 to stworzenie kompleksowego systemu wsparcia niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów, np. poprzez uregulowanie prawne ryzyka niesamodzielności, określenie kryteriów i stopnia niepełnosprawności. Jeśli pan w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, to prosiłbym o odpowiedź pisemną. Jest też priorytet piąty, mianowicie: zastosowanie nowych technologii w opiece nad osobami starszymi i kompleksowe monitorowanie ich poziomu zdrowia, np. przez rozwój telemedycyny i teleopieki. Mam nadzieję i takie wrażenie, że nie chodziło o te teleporady, które wynikały z pandemii, a które przyniosły wiele zła, nie tylko zresztą dla osób starszych. Pytanie aktualne, które tu już padało - inflacja, wszechogarniająca drożyzna. Wzrost cen. Myślę, że to niestety - trzeba tu dodać (Dzwonek) - nie ostatnie słowo.

Dziś rozmawiamy o seniorach, osobach, które przez wiele lat swojej aktywności zawodowej wspierały budowę gospodarki polskiej.

Zaczęliśmy prowadzić spójną politykę senioralną, wprowadzać różnego rodzaju programy, o których już dzisiaj rozmawialiśmy: trzynasta, czternasta emerytura, kwota wolna od podatku. Naprawdę bardzo wiele dobrych rzeczy zaczęło się dziać. O tym dziś należy pamiętać i o tym mówić. Niestety opozycja - dziś słucham jej w tej dyskusji - zapomina, co było wcześniej. Bez pewnego wstydu zaczyna krytykować to, co dziś robimy. Trzeba pamiętać, z czym kojarzy się dzisiejsza opozycja w czasach poprzednich, a kojarzy się w wymiarze polityki senioralnej wyłącznie z podwyższeniem wieku emerytalnego. Dziś chciałbym panu ministrowi bardzo serdecznie podziękować za to, co rząd robi od roku 2015 dla seniorów. Pani poseł Joanna Frydrych, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Działania rządu w obszarze emerytur przez ostatnie 5 lat sprowadzają się do podważania zaufania do państwa. Najpierw obniżyliście wiek emerytalny, skazując kobiety na głodowe świadczenia, później mówicie o konieczności dłuższej pracy. W ciągu 5 lat liczba emerytów wzrosła o 1 mln osób, a ponad 350 tys. osób otrzymuje głodowe emerytury. Czy interesuje was ich los? Od 5 lat zapowiadacie likwidację OFE. Mieliście oddać pieniądze ludziom, a cały czas próbujecie tak zorganizować nowy system, żeby dzięki przekształceniu OFE znacjonalizować prywatne spółki i zabrać Polakom zaoszczędzone pieniądze. To też się nie udało. Aż 80% osób zrezygnowało z tej formy oszczędzania, bo nie wierzą one w przygotowaną przez was politykę inwestycyjną. Drenujecie Fundusz Rezerwy Demograficznej, bo brakuje wam środków na wypłaty trzynastych i czternastych emerytur, a dzięki kreatywnej księgowości obniżacie bezpieczeństwo finansowe państwa. Nie macie planu aktywizacji osób w wieku 60+, zniechęcacie ludzi do dłuższej pracy i skłaniacie do szybszego przejścia na emeryturę, fundując im niższe świadczenia. Zamierzacie wprowadzić niekorzystne rozwiązania podatkowe dla emerytów, którzy otrzymują wyższe świadczenia. W tym roku nie dostaną czternastej emerytury, a w przyszłym roku zapłacą wyższą składkę zdrowotną. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! To jest niepokojące, że w ogóle nie pojawił się ten temat w pana wystąpieniu, a tymczasem jest to temat palący. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze powinny mieć możliwość niezależnego życia, co przewiduje m.in. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Deinstytucjonalizacja oznacza rezygnację z dużych molochów, dużych DPS-ów i realne wsparcie w ramach społeczności lokalnej. Oznacza mieszkania chronione z prawdziwego zdarzenia, dobrą siatkę asystentów osobistych, tworzenie małych ośrodków w lokalnych społecznościach po to, żeby seniorzy jak najdłużej mogli cieszyć się w miarę niezależnym życiem na jak najwyższym poziomie, w lokalnej społeczności, tam gdzie mieszkają wśród swoich sąsiadów.

Moje pytanie brzmi: Dlaczego? Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Nasi seniorzy są często skarbnicą wiedzy, doświadczenia życiowego, są skłonni do dużych poświęceń, pomagają bliskim. W miarę upływu czasu to oni wymagają pomocy i opieki osób drugich. Jedną z form pomocy seniorom, a także osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom są rodzinne domy pomocy społecznej.

Rodzinne domy pomocy tworzone są dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy w tej formie.

Panie ministrze, czy jest rozważane rozszerzenie listy podmiotów, które mogą tworzyć takie domy, i czy rozważana jest możliwość stworzenia dodatkowych zachęt do ich tworzenia? Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Dyskutując na temat opieki nad seniorami, nie sposób nie odnieść się do kwestii opieki zdrowotnej. Chciałabym poruszyć temat mieszkańców domów pomocy społecznej jako osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby, a korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na ogólnych zasadach. Co prawda od lat funkcjonuje podwyższona stawka kapitacyjna, zwiększany jest współczynnik, jednak jak pokazuje doświadczenie, w dalszym ciągu jest to kwota niedoszacowana, co często powoduje, iż znalezienie lekarza, który zdecydowałby się na opiekę medyczną nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, nie jest łatwe. Obecna stawka jest niewspółmierna do nakładów pracy i zaangażowania lekarzy związanych z opieką nad pacjentami z różnorakimi chorobami w tego typu placówkach. Podobna sytuacja dotyczy pielęgniarek środowiskowych, które mają zapewnić opiekę medyczną w domach pomocy społecznej i których brakuje, o czym powszechnie wiadomo. Dotyczy to głównie małych miejscowości. Kiedy rządzący zainteresują się tym problemem? Kiedy zostanie rozwiązana sprawa zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej tak, aby nie traciły uprawnień [[Dzwonek]] i były wynagradzane podobnie jak pielęgniarki pracujące w szpitalach. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jak wynika z przedstawionych w mediach informacji o zamiarach rządu, emeryci i renciści, którzy przejdą na te świadczenia 1 stycznia 2022 r., będą mogli otrzymywać emerytury wyłącznie na konta bankowe, chyba że w drodze wyjątku otrzymają specjalną zgodę ZUS na przekazywanie gotówki pocztą. Emeryci i renciści, także niepełnosprawni, będą musieli o taką zgodę specjalnie zabiegać, często udając się do urzędu osobiście. ZUS może łaskawie taką zgodę wydać, ale nie musi. Mam pytanie do pana ministra. Na podstawie jakiego programu dla polskich seniorów rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zamierza zmuszać seniorów do opłacania kosztów obsługi kont bankowych, które obecnie rosną tak samo gwałtownie, jak rosną koszty jedzenia i koszty utrzymania mieszkania? Zdaniem emerytów i rencistów rząd robi to dla wygody rządowych urzędników, a nie dla wygody seniorów. Uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź w tej sprawie na piśmie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Beata Strzałka, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pani poseł? Jest, przepraszam. Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi szeroką politykę senioralną. Należy zauważyć, że od 2017 r., gdy obniżono wiek emerytalny, rozpoczął się proces wspierania seniorów w różnych aspektach życia społecznego. Oprócz waloryzacji rent i emerytur, wypłaty dodatkowych świadczeń, trzynastej, czternastej emerytury mamy również świadczenie przewidziane programem „Mama 4+” Otrzymują je kobiety, które wychowały czworo dzieci lub więcej. To świadczenie mogą pobierać również ojcowie. To wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenie normuje dochód i pozwala na polepszenie bytu seniorów, a nie na skazywanie wielu z nich tylko na zasiłki z pomocy społecznej. Dla wielu kobiet, matek, które z różnych względów - nie tylko wynikających z posiadania potomstwa, ale również czynników życiowych - nie wypracowały emerytury lub zabrakło im kilku miesięcy składkowych do naliczenia choćby kwoty minimalnej emerytury, właśnie świadczenie „Mama 4+” stało się gwarancją stabilizacji i niezależności finansowej. Program funkcjonuje niespełna od 2 lat, bo od marca 2019 r. Wspomniał pan minister, że już ponad 70 tys. osób korzysta z tego programu. W pełnej wysokości świadczenie pobiera jednak tylko 35% świadczeniobiorców. Dla pozostałych to świadczenie było uzupełnieniem do kwoty najniższej emerytury. Można powiedzieć: tak wiele i tak niewiele, a jednak liczby jasno wskazują, jak niskie były dochody polskich emerytów. To oświadczenie [[Dzwonek]] to wyraz szacunku wobec polskich seniorów. To gest solidarności społecznej. Moje pytanie.

Bardzo konkretna kwestia - budownictwo senioralne. Jaki mieliśmy postęp i jakie są plany? Bo w Polskim czy w Nowym Ładzie słowa na ten temat nie ma, a rzecz jest niebagatelna, bo chodzi właśnie o warunki życia seniorów w okresie starości. A więc pytam: Jak się rozwinął system mieszkań wspomaganych albo serwisowanych? Co ze zrównoważonymi strukturami mieszkaniowymi, czyli sytuacją, kiedy są gwarantowane mieszkania dla osób starszych w normalnej strukturze demograficznej, tak żeby ludzie mieli wsparcie? Budownictwo dla seniorów typu apartamentowce, enklawy senioralne - jakie plany, jakie osiągnięcia, co z tym? Jak wiemy, DPS jest tą formą, gdzie powinni być ludzie najstarsi, już niesamodzielni, bo inaczej mamy mieszkania wspomagane, których jest tak mało. W okresie pandemii okazało się, że DPS-y były miejscem masowych zakażeń. Pytanie dlaczego. Przypuszczalnie również dlatego, że to są obiekty nienowoczesne. Czy przewidziany jest monitoring? Analiza sytuacji? Ile osób zmarło, ile osób było zakażonych, jaki to był odsetek? Jak było w domach zarządzanych przez rękę publiczną, a jak w prywatnych?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To daje 17%, a więc będzie ich przybywać, ten problem będzie narastał. Przed każdym człowiekiem, który wchodzi w wiek senioralny, nowe wyzwania, przede wszystkim wyzwania zdrowotne, wyzwania ekonomiczne. Licząc bazę od 2015 r. do 2020 r., inflacja wzrosła o 9, szanowni państwo, a najniższa emerytura o 42%. Bez tego roku, zaznaczam. Chodzi o kluby seniora i dzienne domy pobytu seniora.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rząd obiecuje seniorom złote góry. W strategii odpowiedzialnego rozwoju promocja aktywności zawodowej i społecznej. Ale strategii odpowiedzialnego rozwoju nie wykonaliście. W najnowszym planie 5-letnim, hasło „Złota jesień życia”, czyli zachęcenie seniorów do pracy po ukończeniu 65. roku życia. A jaka jest rzeczywistość? Wczoraj ekspresem przeszła przez Sejm ustawa o służbie zagranicznej. Ta sama fatalna ustawa, którą trzeba poprawiać, którą trzeba uchwalać jeszcze raz, zanim w ogóle weszła w życie. Art. 4 tej ustawy: stosunek pracy dyplomaty wygasa z mocy prawa w momencie ukończenia przez niego 65. roku życia. W praktyce oznacza to po prostu, że tych ludzi wyrzucacie, pozbywacie się ich. Łaskawie pozwalacie dostojnym jubilatom odwołać się do ministra, który w oparciu o swoje widzimisię może przedłużyć okres powołania. Taki prezent urodzinowy na 65. urodziny. Ten przepis jest niezgodny z polskim Kodeksem pracy, ten przepis urąga normom polskiej konstytucji. Nikt w Polsce nie może być dyskryminowany, przede wszystkim ze względu na wiek, ale ze względu na jakąkolwiek okoliczność. To jest piętnowane i wytykane palcami we wszystkich rozwiniętych krajach. Pan poseł Marek Polak, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Ja, korzystając z okazji, chciałem podziękować obecnemu rządowi i pracownikom resortu rodziny i polityki społecznej za dostrzeganie potrzeb i oczekiwań naszych seniorów, a także za podejmowanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę ich bytu. To w 2019 r. po raz pierwszy w historii polscy emeryci i renciści otrzymali trzynaste emerytury, których nie zaoferowały im nigdy ani władze PRL-u, ani też żadna inna władza po okresie transformacji ustrojowej. Dziś mają to wszyscy zagwarantowane ustawą, a znaczna z nich część może liczyć również na czternaste świadczenia. Ale środki finansowe, choć niezwykle ważne, to jednak nie wszystko, czego potrzebują nasi seniorzy. Walka z osamotnieniem, potrzeba kontaktów międzyludzkich, a także aktywność fizyczna i społeczna to potrzeby, naprzeciw którym wychodziły bardzo dobre w mojej ocenie rządowe programy takie jak „Senior+” i ASOS, które pozwalały realizować się naszym seniorom w całej swojej okazałości. Dlatego chciałbym zapytać pana ministra, czy te i podobne im rządowe programy wspierające naszych seniorów są i będą nadal realizowane, a jeżeli tak, to jakie środki rząd zamierza w nie zaangażować. Dziękuję bardzo. Pan poseł Stanisław Bukowiec, Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma pana posła? Pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wiemy, jak bardzo rząd Prawa i Sprawiedliwości pomaga seniorom, tę politykę senioralną bardzo mocno wspiera. Pamiętamy chyba wszyscy, a szczególnie emeryci rolnicy, rolnicy, którzy są emerytami, jaka niska była emerytura za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu ubolewam, że również Polskiego Stronnictwa Ludowego - to podkreślam. I wiemy, jaką podwyżkę emeryci dostali za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, które wiele lat było w różnych rządach, proponuje zniesienie podatku od emerytur. Ale, drodzy państwo, od wszystkich emerytur, a to znaczy, że ci, którzy mają 10 tys. emerytury, a są tacy w Polsce, skorzystaliby najwięcej.

emerytów, przepraszam, zwolnić emerytów z podatku.

Panie pośle, pan wyczerpał czas. Pan poseł Władysław Kurowski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W 2012 r. rząd koalicji PO i PSL podniósł kobietom i mężczyznom w naszym kraju wiek emerytalny. Zmiana ta była szczególnie drastyczna w przypadku kobiet, które zamiast 60 lat miały pracować 67. Na szczęście rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2016 r. znowelizował tę ustawę, przywracając poprzednio obowiązujący wiek emerytalny, a więc wspomniane 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Za to działanie szczególnie dziękowały kobiety, które wykonywały wymagające fizycznie prace, a dla których nie do przyjęcia było wymaganie od nich jeszcze dodatkowych 7 lat pracy. Obecnie praca po 60. roku życia jest dla nich możliwością, a nie obowiązkiem. Bardzo istotnym programem realizowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest „Senior+”, dzięki któremu jednostki samorządu terytorialnego otrzymują wsparcie na tworzenie dziennych domów i klubów „Senior+”

Korzystając z okazji, chciałbym również serdecznie podziękować za wzrost najniższej emerytury o 42% za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a także za trzynastą i czternastą emeryturę. Co istotne, w założeniach Polskiego Ładu (Dzwonek) znalazła się propozycja, aby emerytury większości polskich seniorów nie były opodatkowane. Nie ma pani poseł. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd Prawa i Sprawiedliwości, powiedziałbym, jako jedyny wprowadził kompleksową opiekę nad seniorami, bo jest wzrost emerytur i są programy pomocowe. W małych, niedużych miejscowościach głównym problemem jest samotność.

Z tego miejsca apeluję do pana ministra, byśmy przyjrzeli się tym programom. Jako osoba uczestnicząca w wielu otwarciach takich domów, miejsc, gdzie mogą się spotykać, wiem, że jest duża potrzeba kontynuowania tego typu wsparcia, bo ci ludzie czują się osamotnieni.

Pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Polacy pracują najkrócej w Europie. Nie oceniam tego. Być może tak jest obiektywnie. Praca jest naturalną wartością, ale jeżeli kolejne setki tysięcy naszych rodaczek i rodaków przechodzą, osiągają wiek emerytalny, to państwo powinno zapewnić przestrzeń systemowej opieki. Opieki liczonej przede wszystkim możliwością tworzenia dziennych domów senioralnych, domów pomocy społecznej, także tych, które są w ustawie - mówię o rodzinnych domach pomocy społecznej - przestrzenią aktywności, wychodzenia z samotności, z depresji.

Polityka senioralna stanie się za chwilę, z uwagi na starzejącą się populację naszych rodaków, jednym z najważniejszych zadań państwa polskiego.

Dlatego apeluję gorąco o zmianę tych zapisów i pomoc w polityce senioralnej państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze przedstawiciel wnioskodawców pani poseł Barbara Bartuś. Dziękuję. Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie najniższych emerytur i rent, trzynasta emerytura corocznie, w tym roku czternasta emerytura, emerytura „Mama 4+”, świadczenia dla osób represjonowanych, zajęcia dla seniorów w ramach programów „Senior+” i „Aktywni+”, program „Opieka 75+”, świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych, to są te elementy, które wypisałam sobie na szybko z wypowiedzi pana ministra i o których wszyscy wiemy.

Tak jak powiedziałam w swoim pierwszym wystąpieniu, starzejące się społeczeństwo jest dla nas wszystkich wyzwaniem. Jest wyzwaniem dla rządu.

Nie potrzebują, żeby ich straszyć, co będzie złego. Państwo mówiliście, że ten okres dla starszych często jest okresem depresyjnym, że nie można wyjść z domu. Dlatego mam apel do opozycji: jeżeli nic dobrego nie zrobiliście przez lata, nie robicie teraz, to przynajmniej nie straszcie, nie uderzajcie w seniorów. Oni naprawdę tego nie potrzebują.

Za naszych rządów walczyliśmy o to, żeby tam w ogóle była opieka zdrowotna.

Po 5 latach traciły uprawnienia do wykonywania zawodu.

Dlatego też bardzo cieszymy się z zapowiedzi, które są w Polskim Ładzie, że nie będzie limitów, że będzie łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Dzisiaj, kiedy to zwolnienie będzie realne, znowu jest narzekanie.

A więc to jest nasz wspólny interes, wszystkich, jako polityków i jako Polaków. Proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo!

Rozpocznę może od tego dzisiejszego, bardzo ważnego tematu dotyczącego szczepień osób w wieku senioralnym. To było priorytetowe działanie, jeżeli chodzi o narodowy program szczepień.

Ale pojawił się tutaj wątek domów pomocy społecznej.

W tym programie wzięło udział - bierze udział, bo program jest kontynuowany - ponad 2 tys. gmin w naszym kraju. Przeznaczaliśmy też dodatkowe środki. Ponad 38 tys. osób z tego programu skorzystało, nie tylko osób w wieku powyżej 70. roku życia.

Pojawił się tutaj wątek dotyczący tzw. emerytur groszowych.

Do tego momentu, żeby otrzymać emeryturę, trzeba było mieć odpowiedni staż emerytalny.

Po prostu tych osób przybywa z racji wieku.

Tych osób jest ponad 71 tys. Polski Ład. Chcemy pomagać tym osobom, które mają słabsze świadczenia.

To też jest rozwiązanie, które będzie wspierać aktywność osób, które chcą dłużej pracować.

Osoba, która chce dalej pracować, pracuje.

Bardzo dziękuję panu ministrowi. Ta wypowiedź kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1200.

Marszałek Sejmu proponuje, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o rządowych projektach ustaw: - o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1176, - o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1117. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1070 i 1176) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wczoraj Komisja Infrastruktury przeprowadziła szczegółowe prace nad rządowym projektem ustawy, który ma powołać nowy byt - społeczne agencje najmu. Sprawozdanie komisji ma nr 1176. Zostało przyjęte 31 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i bez głosów wstrzymujących. W trakcie szczegółowych prac nad projektem komisja przyjęła 28 uwag i poprawek o charakterze legislacyjnym, a także rozpatrzyła dwa pakiety poprawek merytorycznych złożone przez posłów do projektu.

Generalnie materia jest bardzo delikatna.

Te poprawki w głosowaniu zostały przyjęte. Wysoka Izbo!

Dotyczy on stosowania przepisów innych ustaw w odniesieniu do innych rodzajów działalności objętych regulacją tej ustawy. Poprawka ma na celu umożliwienie inwestorom korzystającym z łącznego wsparcia na podstawie omawianej ustawy zawierania z najemcami umów na czas nieoznaczony w przypadku, gdy z najemcą zawarta została jednocześnie umowa partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, a partycypacja ta wynosi minimum 15% kosztów przedsięwzięcia. Ponieważ w zasobie realizowanym wyłącznie z udziałem finansowania zwrotnego taka właśnie możliwość już istnieje, jest uzasadnione umożliwienie stosowania jednego typu umów najmu w ramach jednej inwestycji mieszkaniowej.

Z uwagi na brak czasu nie mogę jej omówić. Dodam tylko, że komisja przytłaczającą większością przyjęła projekt ustawy i apeluje do Wysokiej Izby o to, żeby projekt ustawy przepracowany przez komisję został w głosowaniu przyjęty.

Jako pierwsza pani poseł Anna Paluch, Prawo i Sprawiedliwość, tym razem w imieniu klubu. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Jak już wspominałam jako sprawozdawca, celem omawianego projektu ustawy jest poradzenie sobie z zastojem na rynku najmu mieszkań. Przez zatrzymanie rynku usług turystycznych rynek długoterminowych i krótkoterminowych najmów bardzo na tym cierpi.

Jest to działanie nie tylko gospodarcze, ale także, proszę państwa, działanie społeczne, które wpływa na ubogacenie tkanki miejskiej, bo w jednej przestrzeni będą mogli zamieszkiwać nie tylko ludzie bogaci, ale także ludzie o mniejszych dochodach. Ma to swoje uzasadnienie, zarówno takie dotyczące rozwoju gospodarczego, jak i rozwoju społecznego. Pozwolę sobie tylko w imieniu kluby Prawo i Sprawiedliwość na złożenie poprawek. Otóż przypominam, proszę państwa, że w ustawie zawartej w druku nr 985, czyli ustawie o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, zawarliśmy przepisy, które umożliwiają przeniesienie funduszy, czyli zasilanie zarówno Funduszu Dopłat, jak i Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Chwilę temu mówiłam, że jest bardzo mocna oferta skierowana do gmin, żeby wesprzeć je w realizacji polityki mieszkaniowej. Popularność tych rozwiązań jest tak duża, że te fundusze są bliskie wyczerpania, a sezon inwestycyjny zaczyna się teraz. Chodzi o to, żeby była ciągłość finansowania, żeby gminy, które się zdecydowały na zaangażowanie w realizację polityki mieszkaniowej w mniejszych miejscowościach, to wsparcie miały ciągłe. Chodzi o zasilenie tych dwóch funduszy środkami publicznymi. Właśnie taki przepis znajduje się w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Niemniej jednak Senat po 30 dniach złożył poprawkę, która te przepisy wyrzuca. Stąd też poprawka mojego klubu, żebyśmy mogli jednak utrzymać spójność ustaw, jednej ustawy, czyli tej o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, jak i ustawy zawartej w druku nr 1070. Składam w imieniu mojego klubu poprawki, które są pewnego rodzaju bezpiecznikiem, gdyby się nie udało utrzymać tego kształtu ustawy o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i ochronie praw nabywcy lokalu, domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego. Gdyby się jej nie udało utrzymać w kształcie przedłożenia sejmowego, będzie szansa na to, żeby w obecnie procedowanych przepisach zawrzeć te zapisy dotyczące przeniesienia finansów. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Sibińska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani poseł sprawozdawca mówiła o tym, że poprawki zgłaszane na posiedzeniu komisji przez posłów opozycji wykraczały poza uzgodnienia z samorządami, podczas gdy sama przedstawiała obszerne poprawki.

I dziwnie brzmi troska o samorządy w ustach posłanki PiS-u, podczas gdy wprowadzane są chociażby regulacje wynikające z Nowego Ładu. To jest fałszywa troska o samorządy. Natomiast lepiej nie posługiwać się takimi argumentami, bo trzeba mieć przejrzysty przekaz. Nie lubicie samorządów, ale będziecie robili wszystko, żeby teraz to odczarować.

To, co chcieliście zrobić przez 6 lat, nie wyszło. Nie ma dodatkowych mieszkań mimo zmieniających się ministrów, przepisów i wprowadzanych ustaw, które miały rozwinąć budownictwo. Nic się nie dzieje. Dzisiaj chcemy w przypadku tej ustawy zaangażować do współpracy organizacje pozarządowe i stronę społeczną. Mam takie przeświadczenie, że jeśli pójdzie to w tym kierunku, to organizacje pozarządowe i społecznicy sobie z tym doskonale poradzą. Żeby wzmocnić ich rolę i żeby w lepszy sposób usamodzielnić SAN-y, składam poprawki w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, które doprowadzą do tego, żeby SAN-y, jeśli w porozumieniu z gminami powstaną, miały realny wspływ na politykę mieszkaniową, oczywiście w pełnym porozumieniu z gminami.

W związku z tym SAN-y na podstawie tych kryteriów, które zostaną jako prawo miejscowe ustalone przez gminy, będą mogły podpisywać umowy. Tak jak powiedziałam, element ekonomii społecznej. Jestem przekonana, że będzie to możliwe. W związku z powyższym klub Koalicji Obywatelskiej projekt popiera.

Przepraszam, Wiesław Szczepański, klub Lewicy. W imieniu klubu koalicyjnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec omawianego dzisiaj projektu zawartego w drukach nr 1070 i 1176. W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury rozpatrzyła ten projekt i przyjęła kilka poprawek, oczywiście poprawek koalicji rządzącej. Projekt ten dotyczy wprowadzenia instrumentów mających na celu podtrzymanie funkcjonowania rynku najmu i złagodzenie skutków ograniczeń administracyjnych spowodowanych epidemią COVID-19 dla sektora mieszkaniowego. Ale jest to projekt, który nie rozwiązuje problemu budowy tanich mieszkań. Ten projekt wychodzi naprzeciw właścicielom mieszkań, którzy mają dwa lub trzy mieszkania, a którzy boją się dzisiaj wynająć swoje mieszkanie z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie chronienia lokatorów. Z drugiej strony to możliwość wynajmu tych mieszkań przez osoby, które nie mają możliwości kupna własnego mieszkania, ze społecznej agencji najmu po cenie rynkowej lub cenie z dopłatą, którą określi gmina w obowiązujących przepisach.

Ale trzeba powiedzieć wprost, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi budować mieszkań. Krajowy Zasób Nieruchomości dotychczas nie skorzystał z żadnego prawa pierwokupu, a jego pracownicy odpisują tysiącami na pisma od notariuszy, że nie korzystają z prawa pierwokupu. Dziś Polska boryka się z deficytem ilościowym i jakościowym mieszkań. Brakuje 1,9 mln mieszkań, 5,3 mln Polaków mieszka w mieszkaniach będących w złym stanie technicznym i przeludnionych. Zajmujemy dopiero 24. miejsce w Unii Europejskiej pod względem powierzchni użytkowej i liczby na osobę.

Otóż nie wiemy, dlaczego rząd nie chce, aby tym samym zajmowały się spółdzielnie mieszkaniowe.

A więc proponujemy, aby taka poprawka tam się znalazła, dlatego że jeżeli dajemy taką szansę fundacjom, stowarzyszeniom, które - w przypadku, kiedy będzie dzisiaj możliwość niepłacenia czynszu - będą miały katastrofalną sytuację, jak poradzić sobie z płatnościami na rzecz wynajmującego i jak poradzić sobie z brakiem środków od tego najemcy. Spółdzielnia przy zarządzaniu kilkoma tysiącami mieszkań z takim problemem sobie po prostu poradzi. W związku z tym składamy tę przedmiotową poprawkę i, jak już mówiłem, zagłosujemy za tą ustawą, choć nie jest to ustawa panaceum, która ma rozwiązać problem polskiego budownictwa mieszkaniowego. Głos ma pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1070 i 1176. Model SAN z założenia ma pozwolić gminom zwiększyć ofertę mieszkaniową na swoim terenie bez konieczności ponoszenia przez nie wydatków na budowę mieszkań. Nawiązanie przez samorząd współpracy z SAN umożliwi bowiem wykorzystanie w tym celu istniejących już lokali pozyskiwanych np. z komercyjnego rynku najmu. Ta działalność może ponadto przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności obrotu mieszkaniami na wynajem, w tym w kontekście wyzwań związanych z epidemią COVID-19 na rynku najmu krótkoterminowego oraz spadkiem liczby osób zainteresowanych najmem długoterminowym.

A więc zasadniczo działanie jest potrzebne, konieczne, natomiast pokazuje jedno: Prawo i Sprawiedliwość przekonuje dzisiaj Polaków, że mieszkania, tanie mieszkania, ale będące ich własnością, nie są im potrzebne, bo przecież można wynająć i całe życie przemieszkać w mieszkaniu wynajętym.

Trzeba w tej chwili włączyć do działania te samorządy, które w wielu miejscach, i na tej sali, i w innych miejscach, były krytykowane. Było mówione, że samorządy nie dają rady, a to właśnie opierając się na samorządach i organizacjach pozarządowych, które współpracują z samorządami, będzie można jakąś część tego najmu uporządkować.

Jest nadzieja, że to się uda, bo jeśli włączycie w to samorządy - oby chciały samorządy w to wejść, oby chciały działać wspólnie - to jest szansa na jakieś powodzenie tego przedsięwzięcia. Chociaż samorządy też w wielu miejscach mówiły o tym, że to wcale nie jest program, który mocno ich interesuje i przyciąga. Ale wiemy, jak ważne jest to, żeby zwłaszcza młodzi ludzie mieli możliwość korzystania z tych mieszkań, może w nie najlepszej formule, ale w takiej, która dzisiaj jest dostępna i możliwa, traktując to działanie, tak jak tutaj już padło, jako swego rodzaju pilotaż.

Chciałoby się, żeby też poprawki zgłaszane przez opozycję częściej przechodziły. Natomiast dzisiaj, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem już na wstępie, czyli potrzebę zwiększenia tej liczby mieszkań, my jako posłowie Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego będziemy głosować za tą ustawą. Oczywiście będziemy się też przyglądać, jak to będzie funkcjonować, bo to jest znowu pakowanie w nowe opakowanie tego, co miało działać już wcześniej w innej formule. Dziękuję. Pan poseł Michał Urbaniak, koło Konfederacja.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Z punktu widzenia państwa i jego budżetu to w zasadzie nie są duże pieniądze. Na rynku ma się pojawić planowo ok. 2 tys. mieszkań. W porządku. Zakładamy, że to będą mieszkania dla osób najbardziej potrzebujących, więc z uwagą i sympatią też przyjrzałem się temu projektowi.

Niestety trzeba też przypomnieć kilka nieprzyjemnych rzeczy. Otóż państwo stworzyli program „Mieszkanie+” Niestety ten program to jeden wielki niewypał. Nie rozwiązaliście tym samym problemu dotyczącego potrzeby mieszkaniowej młodych Polaków. Wiemy, że brakuje tysięcy mieszkań na rynku, a ceny rosną i właśnie będą rosnąć, czy wyspowo, czy ogólnie w Polsce.

Wielkie spadki. Szanowni Państwo! Nie wiem, czy to ma być w takim razie w interesie tylko deweloperów i banków, bo być może w interesie Polaków wcale nie będzie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Cieszę się też, że mogliśmy wnieść merytoryczne poprawki i uwagi, przede wszystkim te, które zapowiadaliśmy tutaj, na sali plenarnej, dotyczące wzmocnienia roli organizacji pozarządowych albo innych podmiotów, które będą prowadzić społeczne agencje najmu. Otóż jest gmina, która ma niedobór mieszkań, ma problem z tym, żeby znaleźć mieszkania socjalne i wygospodarować ten zasób, często dla ogromnej, wielotysięcznej kolejki. Teraz, kiedy mamy boom w nieruchomościach, to będzie oczywiście zjawisko nadpodaży mieszkań na wynajem. On zapośrednicza nie tylko wynajęcie, ale też pomaga później, kiedy lokatorzy już wprowadzą się do tych mieszkań.

Po co? Żeby oni nie tylko w tych mieszkaniach mieszkali, ale żeby mieszkania były zadbane, żeby tym osobom, często z niepełnosprawnością lub niesamodzielnym, pomóc w reintegracji, żeby czynsz był płacony, bo to jest bardzo ważne.

Czyli ta ustawa leży gdzieś pomiędzy dwoma sektorami oddzielonych polityk społecznych, czyli między polityką mieszkaniową, która, uprę się na tej Sali, jest jak najbardziej polityką społeczną, i usługami społecznymi, które należy do tej polityki mieszkaniowej dołączyć.

Kto ponosi wszystkie koszty?

Panie Ministrze! Pani Poseł! Koncept społecznych agencji najmu wydaje się trafiony, bardzo sensowny, chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewną kwestię, a mianowicie to, że on w całości zależy od samorządu. Społeczna agencja najmu nie jest pomyślana jako instytucja zaufania publicznego, jako coś, co mogłoby działać, nawet gdyby gmina nie wyraziła takiej woli. Wskazuję na to uzależnienie od samorządów celowo, bo np. na obszarach wiejskich, jak się okazuje, bardzo dużo mieszkań jest wynajmowanych, bardzo dużo, przez rzeczywiście skromnie zarabiających ludzi. Oni są bez żadnej osłony. Imigranci, którzy pracują - legalnie pracują, to są nieraz w niektórych regionach tysiące ludzi. Na przykład kępiński klaster drzewny. Pytanie: Czy ta formuła jest również dla nich? Można by było uporządkować tę trudną sytuację, kiedy okazuje się, że ludzie funkcjonują tam w zasadzie w bardzo złych warunkach. Raz na kadencję może pan. Chodzi też o aspekt integracyjny, bo jeżeli ci ludzie spotkają się z dobrą wolą ze strony państwa polskiego, będą w dobrych warunkach tu funkcjonować i pracować.

Wysoka Izbo! O nieudanych pomysłach rządu PiS-u na tanie mieszkania dla Polaków można by było napisać książkę. A teraz nadszedł czas na społeczne agencje najmu, dzięki którym gminy za pośrednictwem spółek i organizacji społecznych będą mogły zapewnić tanie mieszkania na wynajem. Współpraca samorządów i właścicieli nieruchomości przeznaczonych na najem komercyjny może zasługiwać na aprobatę. Szkoda tylko, że 6 lat zajęło wam, żeby skorzystać z rozwiązań, które z sukcesem przyjęły się w innych europejskich państwach. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie: W jakim czasie od wejścia ustawy w życie należy oczekiwać na znaczną i szybką pomoc adresowaną do właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem? Chciałabym jeszcze zapytać, dlaczego umowy najmu będą zawierane tylko na 5 lat. Czy gminy otrzymają dofinansowanie w związku z tą ustawą i jaka to będzie wysokość? Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Wśród podmiotów, które mogą prowadzić - zgodnie z ustawą - społeczne agencje najmu, są spółki kontrolowane przez samorządy, organizacje pozarządowe, fundacje i spółdzielnie socjalne. Klub Lewicy złożył wniosek, żeby były to również spółdzielnie mieszkaniowe. To ruch o ponadstuletniej tradycji, o dobrze wykształconej kadrze, dzisiaj również zarządzający wspólnotami mieszkaniowymi, a więc dobrze przygotowany do prowadzenia społecznej agencji najmu. Drugą formą, która może prowadzić tę społeczną agencję, jest organizacja pozarządowa. Organizacja pozarządowa dzisiaj, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może prowadzić działalność odpłatną, nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Czy prowadzenie społecznej agencji najmu może odbywać się w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizację pozarządową? Dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewicy. W procedowanej ustawie ani słowem nie odnosimy się do kosztów działalności statutowej społecznych agencji najmu. Jedynym dochodem SAN-ów wymienionych w dokumencie jest dochód z czynszu. Natomiast SAN ma mieć obowiązki sprawozdawcze, musi mieć prezesa, zatem księgowego, pracowników zajmujących się zawieraniem umów. SAN-y mają też odpowiadać za remonty tych lokali, czyli będą pokrywały koszty funkcjonowania całej rzeszy pracowników. Projektodawca przewiduje zawieranie umów gminy z SAN-ami. Zatem w ustawie powinny być wymienione środki dla gmin, a niestety takie środki w ustawie nie są wymienione.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Największym dramatem polskiego rynku mieszkaniowego jest brak przystępnych cenowo mieszkań na wynajem. Winny jest temu brak podaży takich mieszkań i wysoka cena rynkowa tych mieszkań, które są. Ten projekt wychodzi naprzeciw temu, ażeby tę cenę rynkową, różnicę między ceną rynkową a możliwą do zapłacenia, płaciła społeczna agencja najmu.

Dziękuję, pani poseł. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Art. 5 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy jest absolutnie fundamentalny z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb milionów Polaków. Jestem, nie ukrywam, zwolennikiem tego, żeby - po pierwsze - zakazać prywatyzacji tego mieszkaniowego zasobu gminy, tak aby nie sprzedawać mieszkań komunalnych za 5, 10, 15, 20% wartości, z drugiej jednak strony, żeby uelastycznić umowy o odpłatne użytkowanie lokalu, ponieważ można zgodnie z tym artykułem zawierać je wyłącznie na czas nieokreślony. To powoduje, że dzisiaj np. świetnie zarabiający prawnik ma lokal komunalny w mieście X, natomiast rodzina wielodzietna na ten lokal od gminy czeka.

Apeluję do pana ministra jednak o rozważenie zmiany art. 5 ust. 2, korzystając ze swoich doświadczeń jako wiceprezydenta Opola, który zarządzał mieszkaniowym zasobem gminy. Pani poseł Wanda Nowicka, klub Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tanie mieszkania na wynajem dla najuboższych mieszkańców są bardzo ważne i dobrze, że ustawa podejmuje ten problem i stwarza ramy prawne do tego, żeby powstały społeczne agencje najmu. Natomiast same ramy prawne i chęć szczera nie wystarczą, bo za tą chęcią szczerą powinny iść odpowiednie fundusze, które sprawią, że rzeczywiście ten program obejmie o wiele większą populację niż w przypadku tych funduszy, które są asygnowane. Jeżeli w pierwszym roku przeznaczone jest na to 200 tys. zł, co oznacza de facto wsparcie 40 mieszkań, to umówmy się, to nie jest program, który rozwiąże problem. Moje pytanie jest takie: Czy są szanse na to, żeby jednak ten budżet był zwiększony? Bo inaczej rzeczywiście będzie to tylko piękny program, ale bez treści. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Oczywiście program wynajmu mieszkań dla ludzi najmniej zasobnych jest szczytnym programem i na pewno trzeba go rozwijać, ale jakby teraz spytać Polaków, jakie dobro materialne chcieliby mieć od razu na własność czy na jakie dobro materialne by pracowali, to wszyscy powiedzą, że chcą mieć mieszkanie lub dom. Polacy chcą posiadać, chcą być właścicielami mieszkań, chcą być właścicielami domów i państwo powinno im w tym pomóc. Moje pytanie jest takie, panie ministrze: W jakich i w ilu programach państwo uczestniczy, programach, które mają na celu pomóc Polakom i Polkom w kupieniu lub wybudowaniu, kupieniu mieszkania lub wybudowaniu własnego domu? Chciałbym poznać ilość programów i ilość pieniędzy na to przeznaczonych. Proszę o odpowiedź na piśmie. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Uprzejmie dziękuję. Wysoka Izbo!

Otóż taki remont jest możliwy, natomiast później w ramach umowy z właścicielem można rozliczyć koszty w zamian za obniżenie lub czasowe zaniechanie poboru czynszu dzierżawy, ale są różne programy, które umożliwiają choćby termomodernizację, wymianę różnych urządzeń, pieców itd.

Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy listę posłów. Teraz wystąpi podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pan minister Marek Niedużak. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Myślę, że najważniejsza kwestia, która jest istotna, i ważne, żeby tutaj wybrzmiała, jest następująca. Te szacunki, które widzimy w OSR tego projektu, to są właśnie szacunki, a nie limity górne.

Było pytanie o to, czy SAN-y mogą się sprawdzić na terenach wiejskich, czy mogą być odpowiedzią na problemy zamieszkania, jak rozumiem, pracowników, którzy przyjechali do Polski z innych krajów. Teoretycznie tak, oczywiście, to jest jakby po stronie gminy.

W toku konsultacji i uzgodnień spółdzielnie nie wyrażały zainteresowania, nie chciały taką działalnością, przynajmniej wedle naszej wiedzy, się zajmować, tym bardziej że one się jednak zajmują czymś trochę innym, większość spółdzielni zarządza własnym zasobem, stawia też nowe budynki, w których z kolei sprzedaje lokale spółdzielcze. Znaczy, to, co mogę powiedzieć, to jest to, że projekt był szeroko konsultowany. I chciałbym jednak sprostować jedną z wypowiedzi, która nie była pytaniem. Strona organizacji pożytku publicznego jak najbardziej była, wielokrotnie się z nimi spotykano, rozmawiano. Mówię w takim trybie, ponieważ to nie ja prowadziłem ten projekt, tylko pani minister Kornecka, ale wiem, że były takie spotkania. A więc to nie jest tak, że myśmy zupełnie nie rozmawiali ze stroną organizacji pożytku publicznego. To chciałbym też sprostować.

I ostatnie pytanie - dosyć trudne, być może też do szczegółowej odpowiedzi na piśmie - o możliwość korzystania z programów pomocowych. Zasadniczo SAN będzie działał tak, że rzadko, myślę, będzie miał cały budynek, częściej będzie po prostu dysponował czy wynajmował jakiś lokal.

Natomiast trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której.

Natomiast jeżeli cały budynek (Dzwonek), to absolutnie będzie mógł korzystać. Tak że to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Teraz w imieniu sprawozdawców pani poseł Anna Paluch. Wysoka Izbo! W niektórych wypowiedziach podawano w wątpliwość kwestię równoprawnego traktowania poprawek składanych przez różne podmioty. Chcę zaakcentować, że jeśli chodzi o poprawki, które złożyłam w drugim czytaniu, które zostały przyjęte przez komisję, pierwsza i trzecia z tych poprawek miały charakter porządkujący i legislacyjny, a w przypadku drugiej poprawki źródłem jej finansowania jest wsparcie rządowe. A więc tutaj nie ma jakichkolwiek zagrożeń. Druga kwestia, którą też poruszano w wystąpieniach - rozwiązania wprowadzane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, dotyczące normalizacji, normowania sytuacji na rynku mieszkań. Przypominam, że to jest ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, druk nr 985, ustawa lokal za grunt, druk nr 766, ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, druk nr 534, ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane, druk nr 121. To są pierwsze z brzegu projekty, które były procedowane w tej kadencji. Czyli, proszę państwa, rząd konsekwentnie dąży do tego, żeby stworzyć taki system, w którym są poszczególne rozwiązania, jest szeroki wachlarz rozwiązań, jest szansa na synergię pomiędzy różnymi działaniami. To dopiero stworzy takie otoczenie prawne, że polityka mieszkaniowa będzie mogła się rozwijać.

Wszystkie te kwestie służą temu, żeby Polacy mieli więcej mieszkań. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przestawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1086 i 1117) Proszę pana posła Marka Asta o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka mam przyjemność przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1086 i 1117. Powyższy projekt ustawy komisje rozpatrzyły w dniu dzisiejszym. W trakcie prac nad projektem były zgłaszane poprawki, głównie porządkujące, legislacyjne, ale też - przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość - poprawki, które przesuwały terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów projektowanej ustawy. Była też poprawka pana posła Tomasza Zimocha, która nie została przyjęta, a którą w sprawozdaniu przedstawiamy jako wniosek mniejszości. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trakcie prac komisji i prac parlamentu, moim zdaniem, zdaniem klubu Prawo i Sprawiedliwość, zostało wykazane, że ta ustawa jest zasadna i potrzebna, wbrew stanowisku klubów i kół opozycyjnych, które twierdzą, że jedyną intencją tej ustawy jest tzw. skok na kasę, czyli zagarnięcie przez państwo tych pieniędzy, które są w depozytach z tytułu postępowań prokuratorskich. Jest to oczywistą nieprawdą, ponieważ wystarczy, że przypomnę, że to poprzedni rząd, rząd koalicji PO-PSL w 2014 r. wprowadził przepisy, które w podobny sposób uregulowały sprawę depozytów sądowych. Każdy sąd w zasadzie w innym banku, na różnych warunkach te depozyty, które były w gestii sądów, trzymał i wtedy to uregulowano, ustalono, że prowadzi to Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunkach ministerstwa finansów i ministerstwa - już teraz - rozwoju.

Takie argumenty były przedstawiane i my podchodziliśmy do nich pozytywnie, a w tej chwili państwo podchodzicie do tego, że tak powiem, demagogicznie, tylko i wyłącznie politycznie, więc nawołuję do tego, żebyście jednak spojrzeli na to racjonalnie. Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera projekt, wraz z wniesionymi poprawkami.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Mam przyjemność w zastępstwie pana posła Arkadiusza Myrchy zaprezentować stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1086. To jest zresztą kolejna taka ustawa. Pierwszy obszar to jest centralizacja i tutaj też państwo nas niczym nie zaskoczyliście. Centralizujemy kwestie związane z depozytami wpłacanymi w trakcie postępowania przygotowawczego. Do tej pory dysponowały nimi poszczególne prokuratury, w tej chwili ma tym dysponentem być minister finansów.

Nie wiem, czy to ma być jakaś taka forma chwilówki, nie wiem, zarabiania na odsetkach czy też kwestia inwigilowania tego, kto wpłaca, z jakich źródeł wpłaca, skąd pochodziły środki na te depozyty - to już pozostawiam do przemyślenia opinii publicznej. Natomiast m.in. z tych względów klub Koalicji Obywatelskiej nie będzie popierał zmian z druku nr 1086. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Anna Maria Żukowska, klub Lewica. Wysoka Izbo! Tak jak mówiłam wcześniej, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewica postrzega te propozycje jako propozycje ujednolicające, techniczne, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku depozytów sądowych. Nie wietrzymy tutaj podstępu. Trudno tutaj doszukiwać się jakiejś kwestii pożyczkowej, jeżeli chodzi o budżet państwa, dlatego że te pieniądze nadal pozostają prywatne.

Jeżeli chodzi o to, kto jest ich dysponentem, to w ustawie rzeczywiście jest przepis, który mówi, że dysponentami są prokuratury okręgowe.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z wielką uwagą przypatrywałem się dzisiaj przebiegowi prac komisji nad tym projektem. Muszę się przyznać, że czekałem na jakąś refleksję i autopoprawkę ze strony autorów tego projektu, które zmierzałyby do uszczegółowienia tej ustawy, do tego, aby jasno określić status tych środków, które będą gromadzone na rachunku ministra finansów.

Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050.

Bardzo proszę się zgłosić. Dobrze, dobrze. Bardzo proszę. Ja ustąpię. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Powtórzę raz jeszcze: Koło Parlamentarne Polska 2050 popiera zamiar uregulowania zarządzania depozytami uzyskanymi w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę, w szczególności pochodzącymi z zabezpieczeń majątkowych oraz z wpłat poręczeń majątkowych. Zgadzamy się, że intuicyjne postępowanie z zabezpieczonymi depozytami, wzorowane na postępowaniu z depozytami sądowymi, warto zastąpić dobrą regulacją. Takie techniczne zmiany są potrzebne, i to podkreślaliśmy, aby depozyty przechowywać, jak to mówią sami prokuratorzy, w sposób cywilizowany. Koło Parlamentarne Polska 2050 ocenia jednak negatywnie projekt w zakresie tego, by to minister finansów miał uprawnienia do czasowego zarządzania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach depozytowych. Panie pośle, to nie polityka i nie demagogia, to po prostu obawy. Naszym zdaniem jest to bowiem źródło pożyczkowania zgromadzonych na rachunkach niepublicznych środków. Nie widzimy konieczności przekazywania ministrowi finansów uprawnienia do dysponowania tymi środkami. Złożyliśmy w związku z tym poprawkę. Niestety została ona odrzucona, staje się wnioskiem mniejszości. Mamy nadzieję, że zostanie on przyjęty przez Wysoki Sejm i pan poseł sam zmieni zdanie, a także namówi do tego swoich kolegów. Dzisiaj podczas posiedzenia komisji, po złożeniu przez nas poprawki, pan minister stanowczo zaprotestował. Pan minister śpi? Nie. Stwierdził pan, że przyjęcie tej poprawki jest jednoznaczne z głosowaniem przeciw tej ustawie. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Koło Konfederacja jest przeciwko tej ustawie. Krótko to uzasadnię.

Dlatego też jestem przeciwko przekazywaniu tego centralnie i będziemy głosowali przeciwko tej ustawie. Dziękuję. Zgłosili się posłowie do zadania pytania. Jako pierwszy pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo! Proponowana regulacja, dodanie w tym brzmieniu art. 53 ustawy o prokuraturze wydaje się zasadne, gdyż obecnie art. 53 stanowi, że dochody i wydatki powszechnych jednostek prokuratury stanowią w budżecie państwa drobną część. Brak było rozwiązań o charakterze finansowym dających narzędzie techniczne jednostkom prokuratury do przechowywania zabezpieczonych środków finansowych. W konsekwencji prowadzenie tych środków pod egidą ministra finansów jest zbieżne z dotychczasowymi rozwiązaniami obejmującymi sądownictwo i egzekucje komornicze. Ustawodawca proponuje jednak zmianę polegającą na zwolnieniu prokuratora z ponoszenia kosztów wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Nie sposób się, panie ministrze, z tym zgodzić, albowiem forma zabezpieczenia majątkowego zaczęła być w postępowaniach przygotowawczych wręcz nadużywania w stosunku do osób podejrzanych, w tym także do tych, którym nie przedstawiono jeszcze zarzutów (Dzwonek) w formie postanowienia, a więc wobec tych, którzy formalnie nie zaczęli być stroną postępowania przygotowawczego. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Michała Wosia o udzielenie odpowiedzi. Wysoka Izbo! Krótko odpowiem na jedno pytanie. Mianowicie nie można stosować zabezpieczenia wobec kogokolwiek innego niż ktoś, kto ma status podejrzanego. Wobec czego ta informacja przedstawiona przez pana posła nie jest prawdziwa w świetle obowiązującego prawa. Natomiast co do istoty projektu, pozwoli Wysoki Sejm, że w dwóch zdaniach się odniosę. Istotą tego projektu nie jest centralizacja depozytów, bo zgodnie z prawem o prokuraturze to, czy depozyty będą oddawane, czy te poręczenia w jakiś sposób są wykonywane, jest cały czas w kompetencji szefów poszczególnych prokuratur. Projekt ma charakter techniczny i polega li tylko na tym, że prokuratury poszczególne nie będą sobie otwierały różnych rachunków bankowych w różnych komercyjnych bankach, tylko będzie otwierany ten rachunek przez ministra finansów dla poszczególnych dysponentów będących szefami poszczególnych prokuratur - przez ministra finansów, który nie ma żadnego wpływu na to i zapewnia, że te pieniądze, te środki, które są w ramach złożonych depozytów, mają być dostępne w każdym momencie zgodnie z decyzjami poszczególnych szefów prokuratur, którzy pozostają dysponentami tych środków. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu przewodniczącego komisji finansów i swoim własnym chcę podziękować za konstruktywną dyskusję nad projektem - wczoraj było pierwsze czytanie, dzisiaj pracowaliśmy w komisji sprawiedliwości - za wszystkie uwagi zgłoszone do tego projektu. Mam nadzieję, że Wysoka Izba ten potrzebny projekt uchwali, bo, tak jak pan minister powiedział, jest to w tym momencie niezbędne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Czekamy na posła

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1114 i 1200) Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług zawartym w druku nr 1114 (sprawozdanie: druk nr 1200) Komisja Finansów Publicznych w dniu wczorajszym rozpatrzyła projekt ustawy.

Chodzi więc o rozwiązania, które są bardzo potrzebne, szczególnie w okresie pandemii koronawirusa. Przedkładam zatem projekt ustawy w sprawozdaniu komisji zawartym w druku nr 1200. Komisja wnosi o uchwalenie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawienia pozytywnego stanowiska Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1114. Konieczność zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT-u w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Tyle, proszę państwa, niejako suchych faktów. Rzeczywiście pracowaliśmy wczoraj kilka godzin nad bardzo istotną materią dotyczącą szeroko pojętego handlu internetowego. Pamiętajmy o tym, że Polska, ale również wszystkie inne państwa Unii Europejskiej są zobligowane do tego, aby chronić swoich producentów, ale również swoich przedsiębiorców w nierównej konkurencji, często w odniesieniu przede wszystkim do towarów, które napływają do nas szerokim łukiem poprzez funkcjonowanie wszelkiego rodzaju platform sprzedażowych czy też rynków, przede wszystkim azjatyckich, ale też i amerykańskich. Potrzeba nowelizacji i zmiany tej ustawy w zakresie VAT jest niezbędna, bo z roku na rok, szanowni państwo, udział w rynku tych towarów coraz bardziej rośnie, a pamiętajmy o tym, że towary, które nie będą obłożone choćby podatkiem VAT, tak jak w przypadku Unii Europejskiej stanowią, bez dwóch zdań, zdecydowanie lepszą ofertę dla konsumenta końcowego, w której po prostu jest pomijany ten podatek. Tym samym, szanowni państwo, klub Prawa i Sprawiedliwości, jak najbardziej, jeszcze raz powtórzę, będzie głosował za tym rozwiązaniem, które, jesteśmy przekonani, że przyniesie nie tylko dodatkowe wpływy w poszczególnych państwach europejskich, ale również doprowadzi do sytuacji, w której konkurencyjność polskiego czy też europejskiego biznesu będzie dużo większa w stosunku do pozostałej części świata, przede wszystkim azjatyckiego. Bardzo proszę, pan poseł Dariusz Wieczorek, Lewica.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Lewicy przedstawić opinię odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Tak jak mówiliśmy w imieniu klubu Lewicy w pierwszym czytaniu, jest to bardzo skomplikowana materia. Zastanawialiśmy się, dlaczego rząd nie realizował tych zapisów dyrektyw unijnych wcześniej, bo przypomnę, że dyrektywy pojawiły się w roku 2017, później w roku 2019.

Nasze obawy okazały się słuszne, biorąc pod uwagę to, co powiedział pan przewodniczący i mój szanowny przedmówca w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie jest chyba normalne, żeby w ustawie, którą przedkłada rząd, nagle w trakcie posiedzenia komisji pojawiało się kilkadziesiąt różnych poprawek. Legislatorzy mają poważne zastrzeżenia dotyczące konkretnych zapisów. To wszystko jest robione w trakcie. To świadczy niestety o tym, że ta ustawa nie była dobrze przygotowana już na szczeblu rządowym i mam wrażenie, że to wszystko się działo w wielkim pośpiechu wynikającym pewnie z tego, że ktoś przespał, że te przepisy po prostu trzeba do prawa polskiego implementować. To dla jakości stanowionego prawa niestety nie wróży nic dobrego, ale myślę, że poważniejszym problemem jest to, że te wszystkie zapisy i te poprawki są tak skomplikowane, że może być wielki problem z egzekwowaniem tego prawa i też wielki problem z interpretacją dla podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność gospodarczą. Poza dyskusją jest kwestia dotycząca tego, że tę sprawę trzeba uregulować. Biorąc pod uwagę wielki handel z krajów azjatyckich i towary z krajów azjatyckich, które pojawiają się na polskim rynku, czy towary ze Stanów Zjednoczonych, czyli generalnie spoza Unii Europejskiej, bo na to przedsiębiorcy zwracali uwagę, że to jest ewidentne łamanie konkurencji, bo te towary z natury rzeczy już na wejściu są o 23% tańsze ze względu na to, że nie pobiera się podatku VAT.

Jest tylko pytanie, czy przy tym całym pośpiechu i przy tym, co się działo, rzeczywiście uwzględniliśmy wszystkie rzeczy i zastrzeżenia, które pojawiały się, szczególnie w dokumencie, który w ramach analizy tego projektu ustawy był do naszej dyspozycji, a więc stanowiska małych i średnich przedsiębiorców, którzy przedstawili te zastrzeżenia w piśmie swojego rzecznika.

W imieniu klubu Lewicy chcę powiedzieć, że klub Lewicy będzie ten projekt ustawy wspierał. Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

Największy problem stwarza rozwój handlu internetowego z krajami trzecimi, z krajami spoza Unii, gdzie infrastruktura handlowa w obszarze finansowym nie zapewnia pełnej przejrzystości, transparentności całego procesu wymiany. Stąd rozwiązania zawarte w omawianej ustawie są związane z rozliczaniem VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich, ale nie tylko.

Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich, firm. Ustawa ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w Internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w jednym okienku w państwie swojej siedziby, i to państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafia przesyłka, co oszczędzi firmom wielu kosztów i formalności. Interesująca dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe jest planowana zmiana w zakresie rozliczenia VAT od sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów w innych krajach unijnych. Do tej pory każde państwo członkowskie miało określony przez siebie próg dla tzw. sprzedaży wysyłkowej, po którego przekroczeniu następował obowiązek rejestracji sprzedawcy do celów VAT w kraju konsumpcji, co wiązało się dla niego z dodatkowym obciążeniem, np. obowiązkiem składania deklaracji VAT i prowadzenia ewidencji VAT zgodnie z lokalnymi wymogami.

Ma również doprowadzić do zmniejszenia kosztów realizacji obowiązku VAT w związku z transakcjami transgranicznymi. Nastąpi pełniejsza realizacja zasady opodatkowania towarów i usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT będą zasilać budżety państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru bądź danej usługi.

Osobiście mam przekonanie, że wiedza, kompetencje, umiejętności polskich firm w zakresie handlu zrobiły postęp, a więc jestem dobrej myśli, że polskie firmy poradzą sobie z tym złożonym, bardzo trudnym od strony technicznej, wdrożeniowej procesem. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska.

Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Ja nie będę tak słodzić jak pan poseł Siekierski, który mówi, że to będzie konkurencyjność. Ja powiem o problemach, których nie rozwiązaliśmy, i o tym, za co dodatkowo zapłacą Polacy. Wczoraj, w trakcie pierwszego czytania, mówiłam o handlu transgranicznym, o pakiecie VAT e-commerce, o terminie, w którym Unia Europejska w związku ze swoimi przepisami nałożyła na nas obowiązek implementacji. Mówiliśmy o tym, że m.in. nasze towary w tym zakresie powinny być konkurencyjne, jako że w zupełnie innej formule będziemy handlować. Albo przychodzące towary z innych obszarów poza Unią Europejską. Mija 6 lat.

Czy przez te 6 lat udało się im ten VAT obniżyć? Ależ nie! Bo każdego roku państwo od nas z kieszeni pobierali 8 mld zł, nie realizując swojego zapewnienia przedwyborczego. Jeżeli mówimy i porównujemy: będziemy płacili stawkę podstawową VAT - jako że od wszystkich towarów, nawet tych dotychczas zwolnionych, których wartość była niższa niż 22 euro, będziemy płacili VAT - to proszę sobie zobaczyć: Polak zapłaci 23%, Niemiec zapłaci 16%. Będzie stawka podstawowa. A zatem nasze państwo nas obłupi. Nasze państwo nas obłupi. Ale można było - bo można było - wymyślić w tym projekcie, że VAT e-commerce płacimy w jakiejś innej stawce. Można było.

Można było? Bo nasze towary, tak jak i inne, będą wchodzić i będą opodatkowane w innych krajach europejskich. Miejmy nadzieję, że nasi przedsiębiorcy z tego skorzystają. Proszę powiedzieć albo zgadnąć, panie ministrze, jaka jest dzisiaj sensacyjna informacja. Jesteśmy na drugim miejscu w krajach Unii Europejskiej. Z jakiego powodu jesteśmy tak wysoko? Ano inflacja. No właśnie, panie pośle, wygrał pan dzisiejszy teleturniej. I jakoś tak cicho, jakoś nie wiedzę pana premiera Morawieckiego, ministra finansów, który by wystąpił i powiedział: z waszych kieszeni wyciągamy najwięcej w Europie, jak się da. Przed nami tylko Węgrzy. A zatem jeśli mamy poważnie rozmawiać o tym, jak ma wyglądać Nowy Ład, jak mają być wykorzystywane pieniądze europejskie, to przecież rozmawiajcie z Polakami porządnie, poważnie, a nie zaskakujcie albo nie. Chwalicie się tym, czego normalny Polak nie może sprawdzić, ale wierzcie, że o tej inflacji, idąc do sklepu, każdy będzie wiedział, że po prostu naciągacie go na dodatkową zapłatę podatku. Też wyciągniecie ją z kieszeni Polaków, też jako dodatkowe pieniądze wyciągniecie to z kieszeni Polaków. Wy po prostu każdego dnia im zabieracie. Jeszcze jedno powiem: skandaliczne procedowanie, 18 poprawek, co najmniej kilkanaście naruszeń konstytucyjnych trzech czytań, w podatku PIT, w COVID-zie, zmniejszając darowizny, [[Dzwonek]] wprowadzając zewnętrzny system lokalizacji, dając drobne pieniądze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w zakresie ulgi, którą mogą stosować samorządy. Samorządom dajecie. Oni mogą dać ulgę w zapłacie podatku, a wy kasujecie, kasujecie z naszych kieszeni ciężko zarobione pieniądze. Bo to jest dyrektywa, ale nie róbcie tak, nie idźcie tą drogą.

Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, po przedstawieniu sprawozdania komisji ujętego w druku nr 1200. Jak już zostało tu wielokrotnie powiedziane, pakiet e-commerce dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań, które są rozwiązaniami wspólnotowymi i odpowiadają na potrzebę pewnego ujednolicenia podejścia do opodatkowania podatkiem VAT handlu elektronicznego. Wszyscy rozumiemy, że dynamika związana z rozwojem handlu elektronicznego, którą obserwujemy od wielu, wielu lat, a zwłaszcza - myślę - w ostatnim okresie, spowodowała, że rynek jest pod presją różnego rodzaju impulsów, które mogą zaburzać konkurencję.

Oczywiście wszystko ma swoje wady i zalety. Ostateczną decyzję podejmuje konsument, natomiast trudno ignorować sytuację, w której firmy spoza terenów wspólnoty zyskują dochód, klienta, ale nie płacą na terenie wspólnoty - również w Polsce - podatków.

Tutaj należy wspomnieć. Poprawianie niektórych elementów trwało bardzo długo, a wynikało to tylko i wyłącznie z niedbałości w procesie przygotowywania tego projektu ustawy. Otóż rzeczywiście rozwiązania są wspólnotowe, natomiast do dyspozycji państw członkowskich pozostał choćby element dotyczący dokumentowania sprzedaży. Okazuje się, że zgodnie z pomysłem rządu Prawa i Sprawiedliwości nasze firmy będą miały niestety bardziej rygorystyczne warunki dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość niż firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Nasz rząd postanowił, że dokumentowanie będzie możliwe tylko za pomocą dwóch dokumentów. To jest zaskakujące o tyle, że w podobnym przypadku, czyli w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, te dokumenty są niejako wprost stosowane z przepisów dyrektywy, dzięki czemu ich katalog jest szerszy.

Chcemy, żeby nasze firmy były traktowane dokładnie tak samo, żeby nie miały gorszych warunków niż inne firmy z terenu całej Unii Europejskiej. Proponujemy, aby rozszerzyć katalog dowodów, którymi będzie można wykazać, że dostawa została wykonana. Inne firmy w innych państwach Unii mają łatwiej. Naprawdę apeluję do rządu, żeby nie komplikować dodatkowo życia polskim przedsiębiorcom, polskim firmom, polskim pracownikom i przyjąć tę poprawkę. Ona będzie bardzo dobra. Dziękuję bardzo, panie pośle.

One są pozytywne z punktu widzenia interesów obywateli, ale tworzą chaos prawny. W tym momencie chciałbym zaapelować do rządu, aby nie robić takich rzeczy, nie tworzyć chaosu prawnego, zwłaszcza jeżeli (Dzwonek) właściwe ustawy nowelizowane idą przez parlament, a tak jest w tym przypadku. Dziękuję bardzo i proszę o skierowanie projektu do komisji celem wypracowania lepszej propozycji. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Na początku sprostujmy fałszywe założenia tej dyskusji, bo prawdopodobnie ta ustawa z punktu widzenia Polski aż tak wiele nie zmieni.

Polska zapewniła sobie już wcześniej razem z Francją wyłączenie z tego, żeby sprawniej, lepiej łupić obywateli.

Niemal na pewno czekają nas jeszcze kolejne odcinki tego serialu, w którym Unia i Polska będą bohatersko rozwiązywać trudności wynikające z tego, że Unia i Polska systematycznie dewastują własną gospodarkę durnymi przepisami i podatkami. Unia i Polska na wyścigi wymyślają regulacje, które powodują, że wyprodukowanie czegokolwiek na miejscu jest zbyt drogie, że trudno jest wejść na rynek, wskutek czego jest mniejsza konkurencja i wydłużają się łańcuchy dostaw, że przerzuca się na ludzi produktywnych koszty utrzymywania ludzi nieproduktywnych.

Skutkiem tego jest stała ucieczka produkcji za granicę. Taniej jest, jak się okazuje, uszyć majtki na drugim końcu świata, spakować, przepakować, transportować, dostarczać, omijać przepisy, kombinować niż wyprodukować na miejscu. I to jest dramat, tu jest problem. Mówiąc obrazowo, ta presja regulacyjno-podatkowa wytwarza ogromną różnicę ciśnień między obszarem Unii Europejskiej, w którym produkcja jest droga, ale jest ciągle kapitał i bogaty rynek zbytu, a obszarami, w których produkcja bez tych głupich regulacji podatków jest znacznie tańsza. Produkcja ucieka z obszarów droższych do obszarów tańszych, a towary w drugą stronę - z obszaru tańszego do droższego. Żeby temu przeciwdziałać, Unia Europejska próbuje tworzyć bariery zewnętrzne, zamykać się w fortecy. Oczywiście ta różnica ciśnień i tak ciągle się rozładowuje przez jakieś nieszczelności i stąd właśnie sukces AliExpress, który powoduje, że konsumenci w Europie kupują towary, omijając drapieżne łapska swoich urzędów skarbowych.

Nic się nie dzieje. To pokazuje, że te wszystkie regulacje są po prostu zbędne, a ludzie niezależnie od tego, jak głosują w wyborach, tak naprawdę wolą kupić tanio i bez tych unijnych regulacji niż drogo i z pieczątką unijną. Jakieś prześwietlanie przesyłek, arbitralne naliczanie podatku, potem odwoływanie się przez podatników, rozpatrywanie tych odwołań - to wszystko to ogromny wysiłek, który trzeba podjąć tylko po to, żeby państwo mogło z nas zedrzeć więcej podatków.

Oczywiście to jest niesprawiedliwe, że jedni płacą VAT, a drudzy go nie płacą, to jest nieuczciwa konkurencja, ale sprawiedliwość należy wyrównywać w tę stronę, żeby ulżyć tym, co mają za ciężko, a nie dołożyć tym, którzy mają za lekko. Powinniśmy pilnie zmniejszyć VAT, a skoro nie możemy go zupełnie znieść, to możemy próbować zrównoważyć to w inny sposób, np. zmniejszając inne podatki, dochodowe, zdejmując różne ciężary regulacyjne, uproszczając przepisy, rezygnując z wyśrubowanych, absurdalnych regulacji, które zwiększają koszty w Europie i w Polsce. A my co robimy? Ano właśnie, odwrotnie.

Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie sprawimy, że produkcja w Polsce będzie się opłacać bardziej niż import z Chin, to walka z tym importem będzie skutkowała tylko tym, że na miejscu jednej załatanej dziury w murze powstaną trzy kolejne, a jeśli nawet uda się skutecznie opodatkować ten import, to po prostu będziemy musieli kupować drożej i będzie nas stać na mniej. Jeśli opodatkujemy to naszym VAT-em, to będę miał tylko telefon, a kilkaset złotych trafi do rządu, który wykorzysta to na budowanie (Dzwonek) mostów wzdłuż rzeki albo budowę i rozbieranie kolejnych elektrowni w Ostrołęce.

Na koniec: uzależnienie od Chin jest skutkiem nie wolnego handlu, tylko braku wolności gospodarczej w Europie. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się do zadania pytania? Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Przyznam szczerze, że nie mam żadnej. W swojej naiwności nie będę aż takim optymistą. Trzy czytania, proszę państwa, były pomyślane w ten sposób, żeby projekty ustaw były dobre, a nie po to, żeby były one przepychane kolanem na jednym posiedzeniu Sejmu. Natomiast w dniu wczorajszym zadałem konkretne pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi. Proszę o udzielenie odpowiedzi również na piśmie. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowna Pani Marszałek!

Co przez ten czas zrobił polski rząd? nic nie zrobił. Teraz mamy 2 tygodnie na przeprowadzenie wszystkich zmian, które pozostałe kraje Unii Europejskiej przygotowywały przez 3 lata.

Pozostałe kraje robiły to przez 3 lata. Najprawdopodobniej wpadniemy w pułapkę podwójnego opodatkowania, bo jest pytanie, czy nasza administracja skarbowa jest przygotowana do obsługi transakcji importowych zawieranych (Dzwonek) przez osoby fizyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Pamiętam, jak kiedyś kupiłem sobie buty do koszykówki w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce jest ich bardzo mało, koszykówka jest mało popularnym sportem. Zapłaciłem za nie prawie 500 zł. W ciągu tygodnia przyleciały do Polski, następnie spędziły 3 tygodnie w odprawie celnej, a przy odbiorze dowiedziałem się, że muszę dopłacić 100 zł cła za to, że śmiałem przysłać sobie ze Stanów Zjednoczonych buty, które w Polsce były niedostępne.

Szanowni Państwo! To jest tak zagmatwane, że tego się nie da zrozumieć. Powinniście iść w stronę uproszczenia (Dzwonek), obniżenia, likwidacji, a nie wprowadzania kolejnych mechanizmów. To wy powinniście uczyć Unię Europejską, jak powinna to prawo prowadzić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Warto zadać sobie pytanie, co spowodowało, że akurat teraz Unia zaczęła naciskać na ten podatek.

Po drugie, warto zadać sobie pytanie, co robił człowiek, który sprzedawał długopisy, kiedy długopisy chińskie były tańsze.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica.

Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! W uzasadnieniu do projektu ustawy jest informacja, że od 2022 r. przez najbliższe 10 lat w wyniku implementacji tychże rozwiązań trafi do polskiego budżetu co roku kwota 1157 mln zł. Chciałbym zapytać w takim układzie, jak zdaniem resortu finansów wpłynie to na cenę końcową usług i towarów u odbiorców. Druga kwestia dotyczy rozwiązań, o których mówił poseł sprawozdawca, że zostały przyjęte jako poprawki w drugim czytaniu. Dotyczy to podatków od osób fizycznych, od osób prawnych, zryczałtowanych, dotyczy możliwości odliczenia określonych zakupów. Jest pytanie: Jak w trakcie drugiego czytania można wprowadzać tak zasadnicze rozwiązanie? Jakie skutki finansowe będą po wprowadzeniu tychże rozwiązań dla budżetu państwa? Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Wiesław Buż, Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałbym zwrócić uwagę na następującą kwestię: Jak rząd zamierza kontrolować i ewidencjonować obroty w zakresie usługi przewozu osób? Jak wiemy, w Polsce, na terenie całego kraju, prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na pośrednictwie w przewozie osób przez podmioty zagraniczne. Usługa zamawiana jest za pośrednictwem aplikacji internetowej. Klient zamawia usługę przewozową i dokonuje zapłaty z chwilą jej zamówienia. Aplikacja oczywiście jest spięta z kartą płatniczą. Wartość za przejazd wędruje więc w całości na rachunek operatora zagranicznego i zapewne na zagraniczny rachunek podmiotu gospodarczego. Wykonawca usługi, polski podmiot gospodarczy, otrzymuje zwrot od operatora usługi umowną wartość za wykonaną usługę. Czy te transakcje są kontrolowane i opodatkowane podatkiem VAT? Czy nie zachodzi w tym przypadku unikanie fiskalnych czynności? Wiemy, że rynek krajowy w wyniku świadczonej usługi przewozu osób w systemie taxi ma ogromne kłopoty z tak zorganizowaną nieuczciwą konkurencją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. W końcowej części swojego wystąpienia mówiłem o mojej pozytywnej opinii co do stanu przygotowania polskich firm, systemu skarbowego, możliwości tych wszystkich przesyłów elektronicznych, jeśli chodzi o wdrożenie implementacji ustawy. Jednak wypowiedzi pani poseł Skowrońskiej i kolegów zmuszają mnie do skierowania wprost zapytania do pana ministra, jak resort ocenia stan przygotowania do wdrożenia tej ustawy. Bo jednak stoją za tym określone pieniądze.

Następuje powoli, ale następuje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Na zakończenie, pani marszałek, swojego wystąpienia w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej nie powiedziałam, że będziemy głosowali za, albo nie wybrzmiało to odpowiednio. Mówimy o tych niedoróbkach, o tym przekraczaniu przepisów i niekonstytucyjnych poprawkach, które zostały w komisji rozpatrzone.

U nas tego nie ma. Co w tym zakresie państwo rozważacie w przyszłości?

Z tego tytułu są przychody.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Właśnie to jest pytanie, które powinno padać za każdym razem, kiedy debatujemy na temat nowelizacji ustawy o VAT.

Wielokrotnie przegłosowywaliście ustawy, które utrzymywały wysokie stawki. Panie Ministrze! Proszę tu przyjść i powiedzieć, kiedy wreszcie skończycie mydlić Polakom oczy i obniżycie stawki podatku VAT.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Zaczynając od pytań pani poseł Skowrońskiej dotyczących prac nad ustawą, chciałbym przypomnieć, że wszystkie informacje dotyczące zawartości pakietu e-commerce Polska dostała na przełomie listopada i grudnia 2019.

Co do obniżki VAT-u, chciałem państwu przypomnieć, że w zeszłym roku, w lipcu 2020 r. miała miejsce jedna z największych obniżek VAT-u w ciągu ostatnich lat. Został zmniejszony VAT na owoce, pieczywo, pieluszki dla dzieci i wiele artykułów pierwszej potrzeby.

Pani poseł musiała nie usłyszeć.

To jest tzw. mały CIT-owiec.

Przepraszam bardzo, panie pośle.

Mamy świadomość, że w czasach popandemicznych - pandemia pokazała wrażliwość łańcuchów dostaw i to, że odległość geograficzna staje się coraz większym zagrożeniem dla firm, również dla wielkich producentów - wiele globalnych firm rozważa przeniesienie produkcji bliżej ostatecznego konsumenta.

Może nie będą robić. Bardzo dziękuję. Na inne pytania odpowiemy na piśmie. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (druki nr 1128 i 1146) Proszę pana posła Sławomira Skwarka o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, druk nr 1128.

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego krótkiego, składającego się z dwóch artykułów projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. wnosi: Wysoki Sejm uchwalić raczy projekt ustawy z druku nr 1128 bez poprawek. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak powiedział przed chwilą pan poseł sprawozdawca, to krótki dokument, ale szanowni państwo, jakże ważny z punktu widzenia Bydgoszczy, z punktu widzenia całego regionu kujawsko-pomorskiego, ale także i szerzej, z punktu widzenia nauki polskiej.

Dość powiedzieć, że wśród uczelni technicznych zajmuje czołowe miejsce, a jej absolwenci znani są w Polsce i poza granicami kraju. Zasiadają oni także w tej Izbie parlamentarnej, również i w tej kadencji. I pamiętam jak duża była satysfakcja, jak duża była radość, kiedy zmieniano nazwę tej uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Pamiętam, jak uczestniczyłem w uroczystościach nadania uczelni tej nowej rangi, nowej nazwy.

I oto wchodzimy w kolejny etap rozwoju uczelni.

Uczelnia z nawiązką spełnia kryteria, które są niezbędne właśnie do osiągnięcia statusu politechniki. Warto podkreślić, że to umożliwi dalsze, lepsze kształcenie przyszłych absolwentów, a także prowadzenie ważnych, niezbędnych badań naukowych w regionie kujawsko-pomorskim i w samej Bydgoszczy.

Jeszcze jedno słowo, pani marszałek. Chciałem pogratulować władzom uczelni. Chciałem także docenić wkład rządu, a szczególnie pana ministra Schreibera, który pilnował tej sprawy, myślę, w imieniu rządu, a także wszystkich parlamentarzystów regionu kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 28 kwietnia br. wpłynął do Sejmu druk nr 1128 o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. 11 maja na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży odbyło się pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy. Projekt został jednogłośnie przyjęty bez poprawek. Temat powołania politechniki poruszany był od wielu lat wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Rektor uczelni podjął decyzję o przeprowadzeniu ogólnouczelnianego referendum, które odbyło się z początkiem lutego br., i 83% głosujących pracowników opowiedziało się za zmianą nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską. Referendum było jednym z elementów procesu konsultacyjno-decyzyjnego w sprawie zmiany nazwy uczelni. Poparcie dla inicjatywy wyraziły zarówno senat, jak i rada uczelni. Inicjatywę zmiany nazwy uczelni wspierają władze samorządu lokalnego, jak również regionalnego. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła jednogłośnie specjalne stanowisko popierające powstanie politechniki. Wniosek Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego spełnia wszystkie wymagania formalne konieczne do tego, aby przemianować nazwę uczelni na: Politechnika Bydgoska. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora aż w ośmiu dyscyplinach, w których pięć należy do nauk inżynieryjno-technicznych. Bydgoska uczelnia stała się Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w 2006 r., wcześniej funkcjonowała jako Akademia Techniczno-Rolnicza, a jeszcze wcześniej jako Wyższa Szkoła Inżynierska. Obecnie w strukturze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jest siedem wydziałów: budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, hodowli i biologii zwierząt, inżynierii mechanicznej, rolnictwa i biotechnologii, technologii i inżynierii chemicznej, telekomunikacji, informatyki i elektrotechniki oraz zarządzania. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy to największa uczelnia techniczna w regionie, która w swojej 70-letniej historii - rok 2021, nadmienię, jest rokiem jubileuszowym - wykształciła ponad 70 tys. inżynierów. Zmiana w politechnikę pozwoli uczelni pozostać konkurencyjną, utrzymać prestiż, zwiększyć potencjał naukowo-badawczy oraz poszerzyć ofertę kierunków inżynierskich. Uczelnia stale się rozwija i podąża za najlepszymi uczelniami technicznymi w Polsce. Rozbudowuje swoje obiekty dydaktyczne i uczestniczy w innowacyjnych projektach, m.in. w pracach nad prototypem prostego respiratora, który pomyślnie przeszedł testy po podłączeniu do sztucznego płuca. Cieszy mnie ogromnie fakt proponowanego projektu ustawy dotyczącego zmiany nazwy uczelni i powołania do życia Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Tym bardziej cieszy mnie ten fakt jako posłankę z okręgu bydgoskiego [[Dzwonek]] i ziemi bydgoskiej. Klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za projektem ustawy. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Lewicy mam zaszczyt zarekomendować Wysokiej Izbie poparcie projektu ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jest największą i najstarszą w Bydgoszczy uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedynym w regionie uniwersytetem integrującym nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze i ekonomiczne. W ciągu 70 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad 60 tys. absolwentów, a wśród nich uznani w Polsce i za granicą projektanci, architekci, inżynierowie różnych specjalności, budownictwa, mechaniki, architektury, inżynierii środowiska, hodowli i biologii zwierząt, rolnictwa, biotechnologii, inżynierii chemicznej, telekomunikacji i informacji i elektrotechniki. Obecnie na siedmiu wydziałach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach doktoranckich i podyplomowych kształci się ponad 8 tys. studentów. Wysoko oceniane jest kształcenie nowoczesnych kadr inżynieryjno-technicznych, uruchamianie nowych potrzebnych regionowi, krajowi i gospodarce kierunków studiów, budowanie i rozszerzanie indywidualnego toku edukacji, elastyczność procesu kształcenia, wdrażanie systemów umożliwiających studentom odbywanie części studiów na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Uczelnia zajmuje wysokie miejsca w rankingach wyższych uczelni, zwłaszcza w tych, w których oceniane jest przygotowanie absolwentów do zdobycia pracy. Wysoka Izbo! Zmiana nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy następuje na wniosek rektora uniwersytetu wsparty pozytywnym stanowiskiem senatu i rady uczelni oraz wolą pracowników wyrażoną w referendum. Koalicyjny klub Lewicy będzie zawsze wspierał zasadę autonomii wyższych uczelni i zawsze będzie przeciwstawiał się politykom i rządom, którzy mają zapędy do narzucania uczelniom i pracownikom naukowym tego, jak mają myśleć i jak mają działać naukowo.

Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Właściwie moje wystąpienie będzie również kolejną laudacją na cześć tej słynnej bydgoskiej uczelni, jaką jest bez wątpienia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W imieniu klubu Koalicja Polska, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści mam przyjemność przedstawić naszą opinię na temat projektu zmiany nazwy tego uniwersytetu na: politechnika.

W 2006 r. nadano jej miano Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Przez te lata też zmieniał się bardzo mocno profil uczelni - najpierw był to profil techniczny, następnie od lat 70. aż po XXI w. silnie zdominowany przez nauki rolnicze i przyrodnicze.

Edmund Obiała czy też znany kryptolog prof. Józef Pieprzyk. Wielu jej absolwentów, tak jak wspomnieli moi poprzednicy, zasiadało i zasiada nadal w tej Izbie czy też pełniło bardzo ważne funkcje ministerialne. Bydgoska uczelnia jest jedną z najlepszych szkół technicznych w kraju. Współpracuje z wieloma firmami, m.in. ze słynną bydgoską Pesą, i kształci doskonałych specjalistów pożądanych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Spełnia również wszystkie warunki ustawowe do używania nazwy „politechnika”, ponieważ posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach, z których pięć należy do dziedzin z zakresu inżynierii i techniki. Projekt, nad którym w tej chwili procedujemy w Sejmie, był bardzo szeroko dyskutowany i konsultowany w ramach bydgoskiej uczelni i trzeba dodać, że ponad 80% jej pracowników opowiedziało się właśnie za zmianą nazwy na „politechnika”

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja.

Wysoka Izbo! Oczywiście poprzemy to, jest to zmiana techniczna i wymagana też przez lokalną społeczność uniwersytecką, tak że Politechnika Bydgoska stanie się faktem - i dobrze.

Państwo nie powinno też mieć możliwości wydawania pozwoleń na to, żeby uczelnie istniały. Chociaż oczywiście to popieramy, to jednak chciałoby się, żeby społeczność uczelni bydgoskiej mogła sama zdecydować o tym, jak uczelnia się nazywa, a najlepiej, żeby zdecydowała o tym rada właścicieli, spółka prowadząca albo coś w tym stylu. Troszkę żałuję, że przy okazji nie rozmawiamy o jakości kształcenia, bo niestety nasze uczelnie wyższe, nasze polskie uczelnie wyższe nadal pojawiają się gdzieś w okolicy 400. miejsca w rankingu najlepszych uczelni na świecie. To jest temat, a zamiana techniczna nazwy to jest coś zupełnie pobocznego. Przejdźmy przez to, poprzyjmy to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów chce jeszcze zadać pytanie? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy pytanie zadaje pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W zasadzie trudno tu zadawać jakiekolwiek pytania, można jedynie złożyć oświadczenie co do powstania nowej uczelni w sensie nazwy - starej nowej uczelni. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy jest zdecydowanie największą uczelnią techniczną w województwie kujawsko-pomorskim i spełnia wymogi formalne, aby stać się politechniką. Ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w ośmiu dyscyplinach, w tym pięciu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Co ważne, w tym roku obchodzony jest jubileusz 70-lecia istnienia uczelni, zatem jest to idealna okazja i odpowiedni czas do podjęcia przełomowych decyzji, tak ważnych dla rozwoju bydgoskiej uczelni, miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zmiana nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego na Politechnikę Bydgoską to ogromny prestiż. Nowa nazwa przyczyni się do jeszcze większej rozpoznawalności uczelni, a to z pewnością będzie kluczowym argumentem przy (Dzwonek) wyborze uczelni wyższej przez absolwentów szkół średnich. Taka zmiana daje także możliwość poszerzenia współpracy z wieloma gałęziami gospodarki, zwiększa możliwość badań naukowych, a także daje szansę na otwarcie nowych kierunków inżynierskich. Uczelnia będzie też z pewnością poszerzała zakres współpracy z innymi politechnikami, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Istnienie pierwszej w Bydgoszczy politechniki rozbudza nadzieje mieszkańców na zwiększanie potencjału bydgoskiego środowiska akademickiego i oczekiwania przedsiębiorców na nowe efekty w zakresie kształcenia specjalistycznych kadr dla różnych dziedzin gospodarczych i społecznych. W związku z powyższym mam dwa pytania. Na jaką kwotę i na jakie cele może liczyć w 2021 r. i w najbliższych latach Politechnika Bydgoska ze środków Narodowego Planu Rozwoju oraz środków tzw. Polskiego Ładu? W związku z blokowaniem przez polityków PiS ustawy o powołaniu Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy jak długo jeszcze mieszkańcy Bydgoszczy będą czekać na możliwość podjęcia przez Politechnikę Bydgoską współpracy naukowej z nowym, autonomicznym Uniwersytetem Medycznym w Bydgoszczy w celu kształcenia [[Dzwonek]] kadr w zawodach medycznych, tak bardzo potrzebnych w Polsce nie tylko w czasie pandemii? Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Ewa Kozanecka, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy ma na celu zmianę nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na: Politechnika Bydgoska. Ta zmiana jest niezwykle ważna, niezwykle oczekiwana zarówno przez społeczność uczelni, jak i przez mieszkańców nie tylko Bydgoszczy, ale i całego województwa, przyszłych studentów i obecnych studentów z naszego województwa oraz tych, którzy do nas przyjeżdżają.

Panie ministrze, mam pytanie w związku z tą zmianą nazwy. Jak w praktyce zmiana nazwy wpłynie na rozwój uczelni i kształcenie studentów? Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chcę skorzystać z okazji, żeby raz jeszcze podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego awansu, bo tak to traktuję, i tego zasłużonego docenienia osiągnięć dotychczasowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a już niedługo politechniki. Szkoda, że nawet taką rzecz, co do której wszyscy się zgadzamy, niektórzy próbują jakoś upolitycznić i ubrać w jakąś polityczną narrację. To bardzo niedobrze, że próbuje się tutaj mieszać pewne piękne rzeczy, z których wszyscy się cieszmy, z jakąś niepotrzebną narracją, która nie powinna tu mieć miejsca. Dziękuję bardzo. Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pana Wojciecha Murdzka o udzielenie odpowiedzi.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o pytanie pana posła Szopińskiego, trudno odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ponieważ poruszył tematy niezwiązane wprost z tematem tej ustawy. Ale pragnę zapewnić, że środki i krajowe, i unijne na rozwój szkół wyższych są sukcesywnie zwiększane i te możliwości wzrastają. Natomiast pan poseł zdaje sobie sprawę, że zarówno w Krajowym Planie Odbudowy, jak i w Polskim Ładzie nie ma tego etapu, gdzie by były wskazywane konkretne instytucje, podmioty, niezależnie od dziedziny, w związku z tym nie ma również wskazań konkretnych uczelni. A ponieważ też jakby bez związku z tematem pan poseł poruszył kwestię uniwersytetu medycznego, to przy okazji dobra wiadomość dla wszystkich szkół wyższych kształcących lekarzy, pielęgniarki, że w Krajowym Planie Odbudowy jest wyjątkowo dużo środków na ten cel - będziemy to podejmować i koordynować wspólnie z ministrem zdrowia - a mianowicie tam jest kwota 770 mln euro przewidziana na rozwój tego obszaru szkół wyższych, czyli wyjątkowo dużo, adekwatnie do tych potrzeb, które pandemia objawiła. Odpowiadam na pytanie pani poseł Ewy Kozaneckiej. Niewątpliwie celem tej zmiany jest nie tylko kwestia nazwy, ale właśnie kwestia otwarcia perspektywy umożliwiającej intensywny rozwój, rozpoznawalność w regionie, rozpoznawalność międzynarodową, a bez współpracy międzynarodowej trudno sobie wyobrazić dynamiczny i pożądany rozwój szkoły wyższej. Oczywiście jednoznaczne identyfikowanie jako uczelni politechnicznej w regionie, ale nie tylko w regionie, niewątpliwie będzie uatrakcyjniało uczelnię, co, mam nadzieję, zaowocuje przysporzeniem kolejnych studentów, a docelowo absolwentów. Tak sobie pomyślałem, że absolwenci tej nowej uczelni, jeśli chodzi o nazwę, będą w tym rozdaniu środków zewnętrznych, unijnych, w Krajowym Planie Odbudowy, w projektach Horyzont Europa już uczestniczyć jako absolwenci, bo przecież w 2027 r. kończy się ta perspektywa, czyli już pracujemy na rzecz mądrego, dobrego wydawania tych środków, które są przed nami. To też jest droga do wzmacniania pozycji i roli szkoły wyższej, jaką jest politechnika, bo myślę, że przy tym jednoznacznym poparciu taki będzie finał. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej (druki nr 1101 i 1147) Bardzo proszę pana posła Tomasza Zielińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej, druk nr 1101.

Projekt ustawy zakłada utworzenie Akademii Zamojskiej w miejsce funkcjonującej obecnie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i historycznie nawiązuje do uczelni założonej przez Jana Zamoyskiego. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tomasz Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawiam stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej, druk nr 1101. Projekt ustawy zakłada utworzenie Akademii Zamojskiej w miejsce działającej obecnie Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Akademia Zamojska była pierwszą prywatną uczelnią wyższą w I Rzeczypospolitej, zaś do jej powstania i organizacji przyczynił się Szymon Szymonowic. Dewizą akademii zawartą w akcie fundacyjnym z dnia 5 lipca 1600 r. była słynna dzisiaj sentencja Jana Zamoyskiego: „Takie są Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Akademia w początkowym okresie swojego istnienia była ważnym punktem na mapie edukacji Polski, ośrodkiem myśli naukowej. Przez wiele lat zajęcia w akademii prowadzili wybitni profesorowie i naukowcy, m.in. Melchior Stefanides, pierwszy rektor Jan Niedźwiecki-Ursinus, Adam Burski, Tomasz Drezner czy Stanisław Staszic. Po pierwszym rozbiorze uczelnia w 1784 r. została zlikwidowana przez Austriaków, a w jej miejsce utworzono liceum. Przez wiele lat środowiska naukowe oraz samorządowe Zamojszczyzny dążyły do reaktywowania Akademii Zamojskiej, jednak próby te okazywały się zawsze nieudane. Obecnie zgłoszony przez grupę posłów projekt ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej uzyskał bardzo mocne poparcie społeczne, widoczne w szeregu deklaracji administracji samorządowej i rządowej z terenu województwa lubelskiego. Wśród nich należy podkreślić deklarację wsparcia inicjatywy powołania akademii przez prezydenta Zamościa, marszałka województwa lubelskiego czy wojewodę lubelskiego. Projekt ustawy przewiduje zachowanie ciągłości funkcjonowania w Zamościu szkoły wyższej. Mienie dotychczasowej uczelni stanie się mieniem akademii, która przejmie wszelkie prawa i obowiązki uczelni.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc uzyskać do końca 2025 r. kategorię naukową co najmniej B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, biorąc powyższe pod uwagę, będzie głosował za uchwaleniem niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo!

Projekt ma wiele, bardzo wiele fundamentalnych wad i bardzo niewiele słabo umotywowanych zalet. Jest projektem poselskim i to dziwi, bo na posiedzeniu komisji pan minister udzielił mu rekomendacji, zatem powstaje pytanie, dlaczego nie jest to projekt rządowy. Ale można to zrozumieć, gdy czytamy treść.

Ustawa mówi, że nazwa „akademia” przynależy i może być nadana i używana tylko w stosunku do jednostek posiadających co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnia obecnie nie spełnia tego warunku, lecz w strategii jej jest zapisane, że ma osiągnąć te uprawnienia jak najszybciej. Ta niecierpliwość nie jest niczym uzasadniona. Mamy świadomość, że kierunek powołania takiej uczelni jest słuszny dla miasta takiego jak Zamość. Jest słuszny pod warunkiem jednakże, że będzie to uczynione zgodnie z prawem. Rzecz druga: ustawa nie była konsultowana na poziomie projektu przede wszystkim ze środowiskiem akademickim, a dobry obyczaj wymaga tego, aby takie konsultacje się odbyły, nie spotkania, ale konsultacje. To, że były konsultacje samorządowe, to naprawdę za mało. Są negatywne opinie: po pierwsze, Biura Analiz Sejmowych, Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wreszcie Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, które wręcz mówią, że swego rodzaju zaborem mienia jest fakt - to jest w stanowisku - jeśli w ustawie, w art. 4 ust. 1 jest zapisane, że mienie obejmujące własność i inne prawa majątkowe uczelni, obecnej uczelni, czyli Uczelni Państwowej im. I drugi artykuł, który może dziwić, a może nawet przestraszać. Art. 5 ust. 3 mówi, że umowy z pracownikami wygasną 3 miesiące po wejściu w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy. W tej sprawie zgłosimy poprawkę (Dzwonek), bowiem nie możemy się pogodzić z faktem, że pracownicy po 16 latach, a wielu jest takich pracowników. To jest w najwyższej mierze upokarzające dla całego zespołu, dla całej społeczności akademickiej. Przed kilkoma dniami Reuters doniósł, że Viktor Orbán robi reformę szkolnictwa wyższego polegającą na tym, że powstaną fundacje, które będą zarządzały majątkiem uczelni. Chciałabym spytać wnioskodawców, czy byli na specjalnym szkoleniu u Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Dziękuję. I bardzo proszę, pan poseł Marcin Kulasek, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Lewica chce zrównoważonego terytorialnie rozwoju Polski, wspierania miast średniej wielkości, w tym również dawnych stolic wojewódzkich. Jednym z takich miast, które na skutek reformy rządu AWS-UW utraciło status stolicy województwa, jest Zamość. Pierwsze lata po reformie Buzka były dla takich miast jak Zamość bardzo trudne. Dlatego działania zmierzające do budowy lub wzmocnienia instytucji państwowych, w tym instytucji naukowych w miastach średniej wielkości zasługują na poparcie. Niestety uzasadnienie projektu budzi wątpliwości i zaniepokojenie. Jest raczej dalekie od tradycji renesansowego humanizmu, dalekie od wizji Polski otwartej na Europę, prowadzącej dialog z Zachodem. Nie rozumiem, dlaczego projekt ustawy tworzącej nowe uczelnie nie jest inicjatywą rządową. Dlaczego nie przeszedł rządowej ścieżki legislacyjnej z właściwymi jej konsultacjami społecznymi? Czy rząd nie popiera tego projektu? Dlaczego tego projektu nie popiera Polska Akademia Nauk? Dlaczego nie popiera go Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich?

Wszyscy jej pracownicy mają stracić pracę i poddać się weryfikacji dokonanej przez ludzi pana ministra Czarnka. A kto wskaże rektora nowej uczelni? Oczywiście pan minister Czarnek. Zamiast kroku w stronę zrównoważonego rozwoju Polski mamy skok na istniejącą uczelnię wyższą. Zamiast nawiązania do pięknych tradycji Akademii Zamojskiej mamy zapowiedź czystek i próbę utworzenia posad dla swoich. Dlatego w imieniu klubu Lewicy zgłaszam dwie poprawki, tj. wykreślenie przepisu wyrzucającego z pracy pracowników Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica oraz wykreślenie przepisu dotyczącego procedury wskazania rektora. Przyjęcie tych poprawek warunkuje poparcie Lewicy dla dalszych losów poselskiego przedłożenia. Dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł Jan Łopata, Koalicja Polska.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska pragnę przedstawić naszą opinię odnośnie do projektu ustawy ustanawiającej Akademię Zamojską. Wysoki Sejmie! Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli” To słynne i prawdziwe zdanie wypowiedział hetman wielki koronny kanclerz Jan Zamoyski, wielce zasłużony oczywiście dla Zamościa, dla Rzeczpospolitej założyciel Akademii Zamojskiej. A generalnie należy zauważyć i podkreślić z uznaniem, że tradycje akademickie Zamościa i regionu były i są bardzo żywe. Wprawdzie dawna Akademia Zamojska założona w 1594 r. funkcjonowała niespełna dwa wieki do 1784 r., ale jej ogromny dorobek i miastotwórcza funkcja nie zostały zapomniane i przeradzały się w wiele inicjatyw społecznych mających na celu powrót Zamościa do elity miast akademickich. Ziściło się to dopiero w roku 2005, kiedy to Rada Ministrów Rzeczypospolitej podjęła decyzję o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Uczelnia, co warto podkreślić, dysponowała wówczas zaledwie dwoma pomieszczeniami w historycznym gmachu Akademii Zamojskiej. Obecnie, dzięki mozolnej, efektywnej pracy uczelnia dysponuje znaczącym majątkiem. Trzeba zauważyć ten rozwój i dać satysfakcję należną władzom i społeczności uczelni. Ponieważ trudno przejść obojętnie wobec stanowiska społeczności akademickiej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, która ma być przekształcana, które to z żalem informuje, że są za reaktywowaniem Akademii Zamojskiej, ale z poszanowaniem prawa i godności pracowników, którzy od 16 lat budują w Zamościu akademickość tego miasta. Stawiają oni zarzut braku konsultacji, a nawet braku wiedzy o propozycjach ustawy. Stawiany jest również poważny zarzut mówiący o tym, że projekt ustawy podważa autonomiczność i łamie statut. Z takim stanowiskiem zgadza się również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi na interpelację jesienią ubiegłego roku. Podziela to również Polska Akademia Nauk, KRASP.

Biorąc te opinie pod uwagę, a nade wszystko uznając, że został uczyniony gwałt na żywej tkance organizmu uczelni, stwierdzam, że klub Koalicji Polskiej jest za reaktywowaniem Akademii Zamojskiej, ale z poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa i logiki obiektywnego działania. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Pani Marszałek! Tak jak w przypadku poprzedniej dyskusji o Politechnice Bydgoskiej była dosyć duża jasność, tak tutaj niestety niejasności jest ogrom.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc nie posiada statusu uczelni akademickiej.

Szanowni Państwo! Jeżeli jest tyle wątpliwości i jeżeli te wszystkie ciała poza pomysłodawcami tej ustawy są przeciwne temu ruchowi, to należy zadać pytanie, o co chodzi. O co chodzi?

A w związku z tym, że niestety w systemie, o którym mówimy, nie żyjemy, będziecie właśnie decydować siłowo, wbrew decyzji wszystkich istniejących tutaj, wymienionych na stronie sejmowej, ciał. Nie wiem, dlaczego w to brniecie, ale właśnie jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, może chodzić o pieniądze, może chodzić o stanowiska. Dziękuję bardzo, panie pośle. Wysoka Izbo! Mieszkańcy Zamościa i Zamojszczyzny! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Poselskiego Kukiz’15 - Demokracja Bezpośrednia w sprawie sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Akademia Zamojska jest trzecią uczelnią wyższą w Polsce. Funkcjonowała 190 lat i została zlikwidowana przez zaborcę austriackiego w 1784 r. Od wielu lat wskazuje się na potrzebę reaktywowania Akademii Zamojskiej. W III RP zamysł jej wskrzeszenia w 2000 r. znalazł wyraz w uchwale senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, co spotkało się z poparciem kilkunastu regionalnych organizacji, m.in. „Solidarności”, Batalionów Chłopskich, Dzieci Zamojszczyzny, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej czy Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Stosowne uchwały w tym względzie podjęła Rada Miasta Zamość już w 2003 r., a kolejne - w 2004 r., w 2005 r. i w 2019 r. Powołana w 2005 r. wyższa szkoła zawodowa była zobowiązana do działań na rzecz powstania na jej bazie Akademii Zamojskiej.

Z tych też powodów, dzięki wsparciu prezydenta miasta Zamościa Andrzeja Wnuka, w 2019 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zamość.

Obecny ekstraordynaryjny sposób powołania Akademii Zamojskiej jest obowiązkiem parlamentarzystów w celu zadośćuczynienia wieloletnim staraniom władz miasta Zamościa i przedstawicieli strony społecznej, którzy włożyli wiele wysiłku w proces reaktywacji Akademii Zamojskiej. Jest to również spełnienie marzenia ostatniego ordynata hrabiego Jana Zamoyskiego, który już w latach 80. rozmawiał z władzami o reaktywacji Akademii Zamojskiej.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Jeżeli nie, rozpoczynamy pytania. Jako pierwszy pan poseł Jan Szopiński, Lewica.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W projekcie założono, że utworzenie akademii będzie musiało powodować dostosowanie się jej do wymogów określonych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, a więc akademia musi uzyskać kategorię naukową co najmniej B do 2025 r. Mam pytanie adresowane osobiście do pana ministra Czarnka: Czy pozostałe polskie uczelnie zawodowe będą mogły liczyć na taką życzliwość wyrażoną przez pana ministra: z jednej strony jako posła, a z drugiej strony jako ministra? Czy od dzisiaj wszystkie polskie uczelnie zawodowe mogą stać się akademiami? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jan Łopata, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo!

Gdyby się nie dostosowała, to w ust. 2 mówi się, że traci możliwość posługiwania się nazwą: akademia. I podejrzewam, że taki będzie efekt, oczywiście przy innej kadrze, przy innej obsadzie personalnej, ale efekt będzie taki. Czyli innym słowy: Janów Podlaski będzie w Zamościu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Pod pozorem uszczęśliwienia mieszkanek i mieszkańców Zamojszczyzny przeprowadza się zamach na polską naukę i polskie szkolnictwo wyższe. To projekt, który mami przyszłych studentów, kandydatów na studia tym, że będą studiowali na akademii, kiedy uczelnia nie ma takich uprawnień ani nie ma takich możliwości. Sejm łamie wprost ustawę o szkolnictwie wyższym, Sejm doprowadza do tego, że niekonstytucyjne, niezgodne z prawem ustawy są procedowane tylko po to, żeby panowie z PiS, z panem ministrem Czarnkiem na czele, ministrem podpisanym pod projektem ustawy poselskiej, mogli przejąć uczelnie. Jest to niezgodne z prawem, niezgodne z dobrym obyczajem i niesprawiedliwe. Przy okazji jeszcze robią oni czystki na uczelni, wyrzucając pracowników, tylko po to, żeby te uczelnie przejąć. Proszę o odpowiedz na piśmie: Czy to jest tak, [[Dzwonek]] że za chwileczkę okaże się, że jeden z polityków PiS będzie rektorem, a inny kanclerzem? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo!

Zatem pytam: Czy rozwiązania jednostkowe to takie, które są niezgodne z prawem?

Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Czy Zamość zasługuje na akademię? Z pewnością tak. Czy zasługuje na to, żeby tę Akademię Zamojską tworzyć w ten sposób? Absolutnie nie. Proszę państwa, ten projekt ustawy, projekt poselski, jest procedowany wbrew stanowisku społeczności uczelni, przy negatywnej opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wreszcie przy negatywnej opinii Polskiej Akademii Nauk, która wskazuje, że na dziś uczelnia nie spełnia wymogów określonych w Prawo o szkolnictwie wyższym, bowiem nie posiada statusu uczelni akademickiej. Proszę państwa, przeczytam tylko fragment tego uzasadnienia Polskiej Akademii Nauk: Z zaskoczeniem przyjęto uzasadnienie przekształcenia szkoły zawodowej w akademię oraz jej główny cel. W ocenie Polskiej Akademii Nauk jest to sprzeczne z konstytucją, zasadą wolności uprawiania nauki, swobodą dyskutowania i poglądów, wolnością poszukiwania i dochodzenia do prawdy.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Czas, jaki został zaproponowany w projekcie ustawy na spełnienie wymogów z

Moje pytanie do ministra: Jakie dodatkowe pieniądze będą skierowane do Akademii Zamojskiej, aby było możliwe spełnienie wymogów? A pana posła wnioskodawcę prosiłbym o ujawnienie, w oparciu o jakie kierunki Akademia Zamojska spełni wymogi (Dzwonek) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Magdalena Łośko, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proces zmiany nazwy Państwowej Uczelni im. Szymona Szymonowica na Akademię Zamojską jest w drastycznie odmiennym położeniu aniżeli punkt wcześniejszy związany z politechniką.

Apeluję od odstąpienie od siłowych rozwiązań. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki pana Wojciecha

Wysoka Izbo!

W związku z tym podpis pana ministra jest jak najbardziej zasadny. Wydaje się, że kwestionowanie tego jest daleko idącym przedsięwzięciem. Oczywiście w moim komentarzu mówiącym o rozwiązaniu niesystemowym miałem na myśli, i dalej jest to prawdziwe, że inicjatywa posłów nie dotyczy zmiany systemu, tylko dotyczy jednej uczelni, konkretnej uczelni. W tym sensie nie jest to rozwiązanie systemowe.

Oczywiście nie jest tak, że zmiana nazwy jest powiązana z innym sposobem liczenia subwencji, z jakimiś dodatkowymi środkami. Oczywiście poparcie władz lokalnych, regionalnych może zaowocować taką aktywnością. Natomiast zmiana kategorii uczelni na uczelnię akademicką powodowałaby zmianę algorytmu liczenia.

Natomiast oczywiście uczelnia może składać wnioski w tych przestrzeniach, gdzie takie możliwości są stworzone. Nie mamy żądanych sygnałów, żeby takie prace trwały. Dziękuję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt.

Szanowni Państwo Posłowie! To jest normalne w demokracji.

Jeżeli pani poseł pozwoli, to chętnie do przepisów prawa dojdę. Szanowni Państwo! Rozmawiamy o projekcie ustawy, na który czekają mieszkańcy Zamojszczyzny, na który czekają samorządy, ponad 60 samorządów ponad podziałami politycznymi, które wiedzą o tym, że taka uczelnia się temu regionowi należy.

które się, pani poseł, zjednoczyły w Społecznym Komitecie Reaktywacji Akademii Zamojskiej.

Natomiast jeżeli chodzi o prawo, szanowni państwo, zachęcam posłów do tego, żeby.

Jest to taki sam projekt.

To nie jest łamanie konstytucji, reguł nauki. To nie jest łamanie ustawy w sensie systemowym, tak jak powiedział pan minister.

Bo są deklaracje zaangażowania się i finansowego, i poprzez zachęty dla młodzieży.

W związku z tym wydaje mi się, że ten problem jest inaczej ukształtowany. Dziękowałem osobiście rektorowi uczelni państwowej w Zamościu, który powiedział, że misja uczelni, która jest zapisana w projekcie ustawy, jest dokładnie realizowana w tej uczelni.

A teraz jest podnoszony taki problem.

Proszę o zagłosowanie jednak za tą ustawą. Dziękuję. To bardzo ciekawe, że jednostkowe łamanie konstytucji nie jest niczym złym, tylko jednostkowym łamaniem konstytucji. Myślałam, że to jest po prostu łamanie zasad naszego najważniejszego dokumentu. Jakby pan zaczekał chwileczkę, tobym panu wyjaśniła, bo widać, że pan nie zrozumiał, że żyje pan w innym otoczeniu prawnym, niż żył pan w 2016 r. Otóż w tym czasie pojawiła się nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, którą również pan minister Murdzek, obecny tutaj na sali, na pewno panu chętnie przybliży, która zmieniła także zasady dotyczące powoływania uczelni i uprawnień, które mogą mieć. Może się pan powoływać na to, co się działo w 2012, 2003, 1750 r., ale żyjemy w 2021 r., a wy próbujecie oszukać ludzi na Zamojszczyźnie. To, co proponujecie, to jest granda i hucpa. Pomijając, że to jest wstęp do niekonstytucyjnych działań dotyczących obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, to jest to zwykłe oszukanie ludzi, którym mówicie: będziecie na akademii, podczas gdy na akademii nie będą.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk nr 1125) Proszę sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta panią Małgorzatę Paprocką o przedstawienie uzasadnienia projektu.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie inicjatywę ustawodawczą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy: projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Proponowana przez pana prezydenta zmiana Kodeksu cywilnego polega na dodaniu art.

Od wielu lat w praktyce obrotu, ale także w orzecznictwie sądów powszechnych ujawniają się w tym zakresie rozbieżności. Należy pamiętać, że zagadnienie to dotyczy sytuacji bardzo poważnych, przypadków śpiączki pozaurazowej czy stanów wegetatywnych. Po stronie członków najbliższej rodziny poszkodowanego powstaje zatem silna i długotrwała trauma. Na przestrzeni ostatnich lat w orzecznictwie sądów powszechnych ukształtowało się przeważające stanowisko, że tego rodzaju krzywda podlega naprawieniu przez zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Podstawą zasądzania był albo art. 448 Kodeksu cywilnego, albo art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, ale konieczna była dla takiego zasądzenia albo rozszerzająca interpretacja tych przepisów, albo zastosowanie ich w drodze analogii. W praktyce zatem prowadziło to również do sytuacji takiej, kiedy sądy odmawiały zasądzenia zadośćuczynienia.

Ich utrata w następstwie czynu niedozwolonego, np. w wyniku wypadku drogowego, w ocenie prezydenta powinna podlegać naprawieniu przez zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia. W omawianych przypadkach krzywda osoby najbliższej jest niewątpliwie zbliżona do krzywdy, której normatywną podstawę odnajdujemy w art. 446 Kodeksu cywilnego, tj. krzywdy związanej bezpośrednio ze śmiercią poszkodowanego.

Z uwagi na charakter roszczenia oraz ujawnioną rozbieżność w orzecznictwie w ocenie pana prezydenta zasadna jest szybka i adekwatna reakcja ustawodawcy polegająca na jednoznacznym przesądzeniu tej kwestii i ustanowieniu normatywnej podstawy tego typu roszczeń. Proponowane rozwiązanie zagwarantuje przede wszystkim poszanowanie zasady równości wobec prawa, a także spowoduje, że w podobnych stanach faktycznych będzie zagwarantowane rozstrzyganie spraw w analogiczny sposób. Prawo do zadośćuczynienia będzie dotyczyć szczególnie dramatycznych sytuacji, gdy w następstwie ciężkiego i trwałego uszczerbku na ciele lub rozstroju zdrowia dochodzi do niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Zakres podmiotowy zgodnie z propozycją pana prezydenta określony jest w sposób analogiczny do obowiązujących już przepisów Kodeksu cywilnego i dotyczy najbliższych członków rodziny poszkodowanego. Z uwagi na dotychczasową praktykę, ale też zawiłość spraw sądowych pan prezydent proponuje, aby nowe przepisy miały zastosowanie do zdarzeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i w dniu jej wejścia w życie jeszcze nieprzedawnionych.

Pani Marszałek! W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy uprzejmie proszę o poparcie przedstawionego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani minister. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Wysoka Izbo!

Projekt bowiem przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym zapisów, zgodnie z którymi najbliższej rodzinie poszkodowanego, który wskutek wypadku doznał trwałego uszkodzenia ciała, przysługiwać będzie odszkodowanie za naruszenie więzi rodzinnej. W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należy podkreślić, że więzi rodzinne stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania rodziny i podlegają ochronie prawnej - art. 18 i art. 71 konstytucji i art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ich utrata w następstwie czynu niedozwolonego, np. w wyniku wypadku drogowego, powinna podlegać naprawieniu przez zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za zerwane w dramatycznych okolicznościach więzi.

O zerwaniu więzi rodzinnej można mówić jedynie w okolicznościach wyjątkowych, w których doszło nie do zaburzenia, zakłócenia lub pogorszenia więzi, lecz do faktycznej niemożności nawiązania lub utrzymania kontaktu właściwego dla danego rodzaju stosunków, w szczególności więzi łączącej dzieci i rodziców, z powodu ciężkiego i głębokiego stanu upośledzenia funkcji życiowych w następstwie stanu śpiączki pourazowej poszkodowanego lub stanu wegetatywnego, stanu związanego z uszkodzeniem mózgu lub innego głębokiego stanu upośledzenia funkcji życiowych. Chciałbym tu podkreślić, że są to okoliczności, w których doszło nie do zaburzenia, zakłócenia lub pogorszenia więzi, lecz do faktycznej niemożności nawiązania lub utrzymania kontaktu właściwego dla danego rodzaju stosunków osób najbliższych z powodu ciężkiego stanu zdrowia. Ocena wszystkich przesłanek zadośćuczynienia będzie dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy, których obowiązek wskazania będzie spoczywał na dochodzącym zadośćuczynienia. Ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała w takich przypadkach powoduje niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Po stronie członków najbliższej rodziny poszkodowanego powstaje silna i długotrwała trauma. W tego rodzaju tragicznych sytuacjach skutek zerwania więzi rodzinnych jest podobny w zakresie do śmierci bliskiej osoby, a cierpienie najbliższego członka rodziny związanego z takim chorym jest dominujące w dłuższym okresie, zaś intensywność poczucia braku nadziei jest nie mniejsza niż trauma związana ze śmiercią. Ze względu na wagę społeczną przedmiotu regulacji Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera przedstawiony projekt ustawy z druku nr 1125. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Jaśkowiak, Koalicja Obywatelska.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Katarzyna Ueberhan, Lewica.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W dniu wypadku Katarzyna J. miała 17 lat. Była licealistką. We krwi miał morfinę i amfetaminę. Doznała rozległych obrażeń, jej stan lekarze ocenili jako wegetatywny. Od tamtego czasu wymaga całodobowej opieki w każdym aspekcie życia, a szanse na poprawę są nikłe. Edyta B. Od chwili wypadku drogowego, w wyniku którego doznała ciężkiego urazu mózgu, znajduje się w stanie głębokiego wyłączenia świadomości, w stanie wegetatywnym. Nie ma możliwości nawiązania z nią kontaktu. W dniu wypadku miała 34 lata. Była mężatką, matką 6-letniego syna, pracowała jako lekarka, dermatolożka, pisała pracę doktorską. Jest jedynym dzieckiem swoich rodziców. Młoda matka samotnie wychowująca dzieci w wieku 3 i 4 lat na skutek błędu medycznego doznaje obrzęku mózgu, a następnie pozostaje w utrwalonym stanie wegetatywnym. W świetle opinii biegłych strata matki destrukcyjnie wpływa na rozwój psychiczny dzieci, prowadząc do trudności adaptacyjnych, emocjonalnych i uczuciowych. To tylko parę historii, ludzkich tragedii, w których przypadku sąd musiał rozstrzygać o przyznaniu lub odmowie zadośćuczynienia bliskim ofiar przestępstw. Postępowania trwały latami, a rozstrzygnięcia bywały różne. Nie trzeba i nie można czekać. Nie trzeba czekać na wybudzenia osoby w śpiączce, by stwierdzić, że ona i jej najbliżsi cierpią. Nie trzeba i nie można czekać, by za to cierpienie zadośćuczynić. Członkowie rodziny, których bliscy zapadają w śpiączkę pourazową czy w stan wegetatywny, cierpią często niemniej niż w momencie, gdy ich bliska osoba umiera. Przyznanie zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego ma być możliwe w przypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które skutkuje zerwaniem lub niemożnością nawiązania więzi rodzinnych. Wprowadzenie takiej zmiany proponuje niniejsze przedłożenie, prezydencki projekt nowelizujący Kodeks cywilny zawarty w druku sejmowych nr 1125. Proponowana zmiana przepisów ma pomóc w rozstrzygnięciu rozbieżności orzeczniczych, które pojawiły się w ostatnich latach, i to zarówno na poziomie sądów powszechnych, jak i na poziomie Sądu Najwyższego. Obecnie w Kodeksie cywilnym wprost umożliwia się sądowi przyznanie najbliższym członkom rodziny odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jedynie w przypadku osoby bliskiej zmarłej wskutek czynu niedozwolonego.

Członkowie rodzin, których roszczenia nie zdążą się przedawnić, również mogliby zwrócić się o zapłatę zadośćuczynienia, jeśli spełniliby wymienione kryteria. Ze względu na znaczenie społeczne problemu nowelizacja ma wejść w życie w ciągu miesiąca od jej ogłoszenia.

Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Byłem przed chwilą na posiedzeniu Komisji Zdrowia, na której był projekt ustawy. Wszyscy posłowie Lewicy, PO prześcigali się, żeby tej grupie dołożyć, tej dołożyć, tej dołożyć, tamtej dołożyć, oczywiście z kieszeni tych ludzi, którzy nie mają pieniędzy na pomoc swojej krewnej, która uległa ciężkiemu wypadkowi. A ci z kolei nie mają pieniędzy, bo poszło na nią. Gdyby państwo odbierało ludziom jakieś uprawnienia, to byście wrzeszczeli. Ale jeżeli państwo odbiera im konieczność płacenia na coś czy utrzymania czegoś, to się mówi, że to bardzo dobrze, że państwo zdejmuje ciężar. Tym samym jednak zdejmuje również odpowiedzialność. Znika poczucie więzi rodzinnej, człowiek uważa, że to nie on ma się opiekować kalekim członkiem rodziny, tylko że od tego jest państwo. Państwo, które odpowiada za wszystko, ma również wszelkie prawa. Jeżeli odpowiada za wszystko, to ma prawo pobierać podatki na to, żeby to wszystko robić.

Ten koszt społeczny spada na całe społeczeństwo. Gdy się popłacze trochę nad tym, da 5 czy 10 przykładów ludzi, którzy cierpią i nie mają pomocy, można spowodować, że Sejm zechce się przychylić i wydać pieniądze podatnika, nie widząc, że być może te pieniądze są babci, która dzięki temu zje tylko jedną bułkę, bo na drugą już jej nie będzie stać.

Tak że niestety dobre serce to jest na Lewicy, prawica ma rozum. Prawica nie kieruje się dobrym sercem, bo dobrym sercem to można tylko doprowadzić kraj do ruiny. Jeżeli dobry tatuś daje synkowi wszystko, o co synek prosi, to doprowadzi go do ruiny, zdemoralizuje. To samo dotyczy rządu, który tak traktuje społeczeństwo. Tak że to dotyczy sprawy pryncypialnej, ta sprawa jest drobna, ale jest niesłychanie charakterystyczna. Godząc się na to, powodujemy kolejny drobny rozrost państwa, uznajemy odpowiedzialność państwa, a więc też prawo państwa do zajmowania się wszystkimi i wszystkim, uznajemy, że państwo odpowiada za wszystkich. Jest to klasyczny ustrój niewolniczy. W ustroju niewolniczym pan odpowiadał za swojego niewolnika i musiał go leczyć.

I dla zasady będę głosował przeciwko. Dlatego że - powtarzam jeszcze raz - ważne są zasady, a nie poszczególne przypadki. Musimy patrzeć, jak działa prawo, ale również na to, jak to prawo oddziałuje na społeczeństwo.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050. Pni Marszałek! Wysoki Sejmie! A ja uważam, że to dobrze, że pojawia się propozycja prawnego rozwiązania zapłaty zadośćuczynienia, kiedy najbliższy członek rodziny dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu, który skutkuje niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Projektodawca ma na myśli szczególnie dramatyczne sytuacje, kiedy w następstwie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest już możliwe występowanie więzi rodzinnej. To mogą być stany śpiączki pourazowej, panie pośle, uszkodzenia mózgu. Trudno jednak o dokładne wymienienie zdarzeń, w wyniku których można będzie występować o takie zadośćuczynienie. Istotne będzie jednak określenie, co jest więzią rodzinną i między kim ona rzeczywiście występuje. Bo przecież warte odnotowania jest to, że przepisy prawa cywilnego posługują się pojęciem osoby bliskiej, osoby najbliższej, ale w kodeksach nie znajdziemy dokładnych definicji tych pojęć. Eksperci prawni Koła Parlamentarnego Polska 2050 sygnalizują, by w projekcie określenie „najbliższy członek rodziny” zastąpić pojęciem „najbliższa osoba” Nie pędźmy z tym projektem, jak to często bywa w tym Sejmie. Dyskutujmy, dopuśćmy do głosu ekspertów, w tym przypadku weźmy pod uwagę różne opinie prawne, bo przecież w doktrynie dyskusyjna jest możliwość przyznania odszkodowania konkubentom, wychowankom zmarłego, narzeczonym czy innym osobom niepozostającym w relacji pokrewieństwa, powinowactwa czy w przysposobieniu.

Są też i tacy przedstawiciele doktryny, którzy uważają, że do rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego należy też zaliczyć wychowanków, narzeczonych, konkubentów, jeżeli ich związek ma charakter dostatecznej trwałości i cechuje się dostatecznie silną wspólnością gospodarczą. Koło Parlamentarne Polska 2050 popiera ten projekt, bo uważamy za słuszne przyznanie zadośćuczynienia, ale rzeczywiście osobom najbliższym poszkodowanemu, z którym nie występuje już więź. Zgadzamy się z panią minister. Pamiętajmy w tym przypadku o poszanowaniu i równości wobec prawa. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. 1 minuta na zadanie pytania. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na wstępie, panie pośle, z całym szacunkiem do pana, tu państwa nie będzie. Nie podejrzewam ludzi, którzy uczestniczą w wypadkach drogowych, że chcą mieć wypadek. Jest to zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne. Tu będzie tylko orzeczenie sądu, który wreszcie uporządkuje sprawę bardzo ważną dla wielu, wielu ludzi. A teraz przejdę do pytania, które poniekąd pan poseł Zimoch już zadał, a mam podobny tok myślenia. Mamy osobę, która jest jedynym żywicielem rodziny, ale jest osobą najbliższą dla tychże osób, czyli nie jest rodziną w myśl kodeksu. Doznaje ona wypadku: Czyli kto będzie generalnym beneficjentem projektu? Kto skorzysta na ustawie? Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Prezydencie! Panie Ministrze! Chciałbym serdecznie podziękować panu prezydentowi za ten bardzo ważny projekt ustawy. Projekt bardzo krótki, bo zaledwie kilkuzdaniowy, ale jakże niezwykle ważny z punktu widzenia, znaczenia społecznego, z punktu widzenia doniosłości tego projektu. Rzeczywiście tak jest, że ta potrzeba nowelizacji wynika właśnie z tej rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Ta dominująca linia orzecznicza mówi o tym, że rzeczywiście są zasądzane przez sądy zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny poszkodowanego za krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej, ale dobrze wiemy, jak to również w tej dyskusji zostało zaprezentowane, że zdarzają się przypadki odmawiania przez sądy tego odszkodowania. Więc raz jeszcze dziękuję za tę kolejną inicjatywę (Dzwonek) ustawodawczą pana prezydenta. Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny to z całą pewnością dobra inicjatywa, potrzebny akt prawny, który zmierza do rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie przyznawania zadośćuczynienia wypłacanego najbliższym. Chciałbym za pośrednictwem pani minister zwrócić się do pana prezydenta o to, aby w swojej aktywności częściej przedstawiał tego typu projekty, częściej działał, tak jak oczekują tego rodacy, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją, bo niestety dotychczasowa praktyka była zupełnie inna. Poczytuję ten projekt ustawy jako zwrot w dobrym kierunku. Pani poseł Monika Falej, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związku z przedłożonym projektem ustawy przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy - Kodeks cywilny chciałabym uzyskać konkretne informacje. Może akurat macie państwo takie dane. Ile osób, ile rodzin osób poszkodowanych przestępstwem, w wyniku którego osoby poszkodowane zapadły w śpiączkę pourazową czy trwały stan wegetatywny, otrzymało do tej pory czy otrzymuje średniorocznie i w jakiej wysokości zadośćuczynienie? Ile osób otrzymuje zadośćuczynienie na podstawie obowiązujących obecnie przepisów w wyniku pozytywnych rozstrzygnięć postępowań sądowych, a ile takich rozstrzygnięć oddalono czy średniorocznie się oddala?

Jak wiele spraw o zadośćuczynienie dla rodzin osób poszkodowanych przestępstwem zawieszono (Dzwonek), a ile nie zostało rozstrzygniętych na podstawie obecnych przepisów, a miałoby to do nich zastosowanie obecnie proponowane rozwiązanie. Na jakiej wysokości zadośćuczynienie mogą liczyć rodziny w konsekwencji przyjęcia i stosowania proponowanego rozwiązania ustawowego? Dziękuję i poproszę informację na piśmie. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Więzy rodzinne stanowią fundament prawidłowego funkcjonowania rodziny i podlegają ochronie prawnej. Ich utrata w następstwie czynu, np. w wyniku wypadku drogowego, powinna rzeczywiście podlegać naprawieniu przez zapłatę odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Słuszny jest tego typu kierunek rozumowania. Tego typu rozwiązanie jest m.in. niezbędne do realizacji konstytucyjnej ochrony rodziny, o której mowa w art. 18 konstytucji, oraz zasady równości wobec prawa.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta panią Małgorzatę Paprocką.

Pani Marszałek! Na wstępie chciałam bardzo uprzejmie podziękować za wyrazy poparcia dla projektu pana prezydenta. Tak naprawdę wszystkie pytania sprowadzają się do kwestii definicyjnej i kręgu beneficjentów. Projekt pana prezydenta odwołuje się do dzisiejszej siatki pojęciowej w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego i dla spójności systemu prawnego posługuje się kategorią najbliższych członków rodziny.

Dziękuję bardzo, pani minister. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Romanowskiego. Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam przyjemność zaprezentować podstawowe elementy projektu stanowiska rządu, który jest na końcowym etapie procedowania. Jest również jednoznacznie pozytywny co do celu tej regulacji. Będziemy proponować, rekomendować projekt do dalszych prac legislacyjnych z pewnymi drobnymi uwagami do rozważenia w trakcie procesu legislacyjnego, ponieważ zasadniczo propozycja zasługuje na aprobatę. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego regulacji, która będzie jednoznacznie przesądzała o przysługiwaniu osobom najbliższym bezpośredniego poszkodowanego roszczenia o przyznanie zadośćuczynienia z tytułu wspomnianej krzywdy, która wynika z pozostawania bezpośredniego poszkodowanego w stanie powodującym niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, jest rzeczywiście potrzebna. To wprowadza pewność prawa, usuwa stany niepewności wynikającej z dotychczasowego orzecznictwa i oczywiście uzasadnia konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, a także zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez niego prawa. Bo rzeczywiście jest tak też, poniekąd odpowiadając na również na uwagę pana posła Korwin-Mikkego, że mamy do czynienia z roszczeniem, które jest kierowane nie do państwa, tylko do sprawcy tej szkody o zadośćuczynienie, czyli na zasadzie sprawiedliwości wyrównawczej, a nie sprawiedliwości dystrybutywnej czy rozdzielczej. Zwracamy uwagę na kilka kwestii, które niewątpliwie mogą być rozważane w trakcie dalszych prac legislacyjnych, niewątpliwie należałoby zwrócić uwagę na zwiększenie ilości spraw w sądach. Poniekąd też sygnalizując, mówimy o następujących liczbach. Nie ma niestety pełnych danych, które można by wskazać, ile osób może skorzystać z zadośćuczynienia, ponieważ statystyki sądowe mówią łącznie o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach.

Oczywiście na tym tle to będą tylko szacunki, ile spraw na podstawie tego nowego roszczenia może znaleźć się w sądach. Wskazujemy też oczywiście do rozważania kwestię retroaktywności - nie tylko ze względu na cel, co również zawsze jest ważne, ale również co do konstrukcji.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu na podstawie art. 87 ust. 2, w związku z art. 90 ust. 1 regulaminu Sejmu, kieruje przedstawiony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, zawarty w druku nr 1125, do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Ogłaszam 3 minuty przerwy.

Wznawiam obrady. Obecnie przystąpimy do stwierdzenia kworum. Bardzo proszę wszystkich państwa posłów o naciśnięcie dowolnego przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Bardzo proszę.

Stwierdzam kworum. Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu 24. Powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 1139 i 1151) Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1185, 1174, 1175 i 1166. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1182, 1178, 1197 i 1177. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 1204 i 1205. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1208. W związku z tym na podstawie art. 74 regulaminu Sejmu podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wznowienia „Wiadomości” Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z druku nr 1171. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 1171, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wznowienia „Wiadomości” Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1127. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1127, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku. Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1162. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1162, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1122-A. Proszę pana posła Bolesława Piechę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo!

W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy w całości oraz poprawkę.

Tym samym, zgodnie z zasadami legislacji, poprawka również uzyskała rekomendację negatywną. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1122. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu wniosek o odrzucenie projekty ustawy w całości oraz poprawkę, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Obecnie pod głosowanie poddam zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowodowuje bezprzedmiotowość pozostałej propozycji. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w całości. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce nacisnąć

Sejm wniosek odrzucił. W jedynej poprawce wnioskodawcy proponują inne brzmienie art. 9a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę odrzucił. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1122, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1149-A. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Wiesława Szczepańskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W czasie drugiego czytania do tej ustawy wpłynęło osiem poprawek. Komisja w dniu wczorajszym rozpatrzyła zgłoszone poprawki i rekomenduje odrzucenie poprawki od 1. do 4. i przyjęcie poprawki od 5. do 8. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1149. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Wszystkie poprawki zgłoszone zostały do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Komisja wnosi o ich odrzucenie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił.

Komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy.

Sejm poprawkę przyjął. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Głosujemy.

W 8. poprawce wnioskodawcy proponują nowe brzmienie pkt 5 w załączniku do ustawy w części Kategoria A. Głosujemy.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1149, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1150-A. Proszę pana posła Mieczysława Baszkę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W drugim czytaniu zgłoszono dwie poprawki. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 19 maja rozpatrzyła poprawki. Natomiast komisja przyjęła rządowy projekt ustawy i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Z poprawką tą łączy się poprawka 2. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Głosujemy.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1150, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1148-A. Proszę panią poseł Beatę Strzałkę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, druki nr 1015 i 1148. Sejm na posiedzeniu w dniu 19 maja, zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia dwóch poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja po rozpatrzeniu poprawek na wczorajszym posiedzeniu wnosi, aby Wysoka Izba poprawki odrzuciła, a tym samym przyjęła projekt ustawy bez poprawek. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1148. Komisja przedstawia również wnioski mniejszości oraz poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. We wnioskach mniejszości 1., 3., 4. i 5. wnioskodawcy proponują m.in., aby świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwały niezależnie od dochodu rodziny. Nad tymi wnioskami mniejszości będziemy głosować łącznie.

Sejm wnioski mniejszości odrzucił. W 2. wniosku mniejszości do art. 5 pkt 1 lit. b wnioskodawcy proponują coroczną waloryzację kwoty dochodu uprawniającej do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 1. poprawce do art. 5 pkt 1 lit. b wnioskodawcy proponują m.in. coroczną waloryzację kwoty dochodu uprawniającej do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. W 2. poprawce do art. 18 ust. 1, 2 i 4 wnioskodawcy proponują m.in., aby pierwsza waloryzacja kwoty dochodu uprawniającej do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego została przeprowadzona w 2022 r. Głosujemy.

Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1148, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1169-A. Proszę panią poseł Elżbietę Dudę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1145 i 1145-A. Sejm na 30. posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1169 do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Poprawki od 1. do 7. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. poprawki wraz z konsekwencją, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki wraz z konsekwencją, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę przyjął.

Głosujemy.

W 8. poprawce wnioskodawcy proponują dodać do projektu ustawy nowelizującej art. 1a zawierający zmiany do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Z tą poprawką łączy się poprawka 11. Głosujemy. Kto jest przeciw?

W 10. poprawce wnioskodawcy proponują dodać do projektu ustawy nowelizującej art. 2a zawierający zmiany do ustawy o działach administracji rządowej. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 12. poprawce wnioskodawcy proponują dodać do projektu ustawy nowelizującej art. 3a zawierający zmianę do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Proszę państwa, anulujemy to głosowanie, ponieważ państwo mówią, że jest zła informacja, zły opis.

Tak, tak, nasi też, panie pośle, tak że okej.

Proszę nie brać pod uwagę numeru głosowania, tylko numer poprawki pod spodem. Poprawka 13. - to jest już

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Sejm poprawkę przyjął. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1169, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1184. Komisja przedstawia jednocześnie wnioski mniejszości, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Głosujemy.

W 2. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują, aby pozostawić w obowiązującym brzmieniu art. 3 i 4. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

W 4. wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują, aby uchylić art. 9. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. wniosku mniejszości, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek mniejszości odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1184, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie zagranicznej. Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1117. Komisje przedstawiają jednocześnie wniosek mniejszości, nad którym głosować będziemy w pierwszej kolejności. W jedynym wniosku mniejszości wnioskodawcy proponują, aby w art. 53a

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1117, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 1200-A. Proszę pana posła Henryka Kowalczyka o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym w czasie drugiego czytania do ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT zgłoszono jedną poprawkę. Komisja Finansów Publicznych po jej rozpatrzeniu nie rekomenduje przyjęcia tej poprawki i rekomenduje przyjęcie całej ustawy. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1200. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu poprawkę, nad którą Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1200, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 1128. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1128, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm uchwalił ustawę o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1154 i 1185) Proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1154. Marszałek Sejmu skierowała w dniu 17 maja br. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w dniu 19 maja br. wnosi, by Wysoki Sejm raczył odrzucić poprawkę Senatu. Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W punktach porządku dziennego dotyczących rozpatrywania poprawek Senatu głosować będziemy nad wnioskami o odrzucenie poprawek Senatu. W jedynej poprawce do art. 7 ustawy o dowodach osobistych Senat proponuje dodanie ust. 4. Głosujemy.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1152 i 1182) Proszę pana posła Tomasza Zielińskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1152. Połączone komisje na posiedzeniu w dniu 18 maja rozpatrzyły cztery poprawki Senatu i wnoszą, aby Sejm wszystkie poprawki odrzucił. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów.

Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1155 i 1174) Proszę pana posła Witolda Czarneckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywała uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz innych ustaw. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie wszystkich poprawek. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.

jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy.

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk.

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Senat proponuje zmianę w części wspólnej. Głosujemy.

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1157 i 1178) Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1157.

Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. W uchwale Senat proponuje odrzucić ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1156 i 1175) Wysoka Izbo! Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Senat zaproponował 23 poprawki. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich poprawek Senatu. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Senat zgłosił do art. 1 ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy - Prawo energetyczne.

Głosujemy. Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął.

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 1153 i 1197) Proszę pana posła Grzegorza Matusiaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odrzucono uchwałę Senatu dotyczącą odrzucenia ustawy o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przypominam, że Sejm odrzuca uchwałę Senatu odrzucającą ustawę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeżeli Sejm nie odrzuci uchwały Senatu odrzucającej ustawę, uważa się ją za przyjętą. Głosować będziemy nad wnioskiem o odrzucenie uchwały Senatu. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej ustawę z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1160 i 1166) Proszę pana posła Krzysztofa Lipca o przedstawienie sprawozdania komisji.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo Mam przyjemność w imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tej uchwały stwierdza, że Senat wprowadził do wymienionej ustawy trzy poprawki.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Głosujemy. Kto jest przeciw?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 3. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 1158 i 1177) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z druku nr 1158 Senat uchwalił 16 poprawek.

Wszystkie wymienione poprawki mają charakter redakcyjny i legislacyjny. Zwłaszcza poprawka 2. rodzi podejrzenie niekonstytucyjności, ponieważ skutkuje tym, że takie same podmioty w takich samych warunkach będą traktowane w inny sposób. Nabywcy, którzy będą wpłacać środki na otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, będą traktowani inaczej niż nabywcy korzystający z zamkniętych mieszkaniowych rachunków powierniczych. Poprawki 7. i 9. głosowane łącznie także należy odrzucić.

Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. Przystępujemy do głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy.

10 - za, 440 - przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto jest przeciw?

Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 11. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

450

Sejm poprawkę przyjął. Z poprawką tą łączy się poprawka 14. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 12. i 14., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 13. poprawki, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 15. i 16., zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm odrzucił poprawki bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23. porządku dziennego: Wybór uzupełniający sędziego-członka Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 1124 i 1168)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ustaliła kandydatkę na stanowisko sędziego-członka Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Lipca w celu przedstawienia sprawozdania komisji.

Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie listy kandydatów na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Pani marszałek stosownie do przepisów regulaminu Sejmu i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przedstawiła komisji dokument w sprawie wyboru kandydata sędziego na członka Krajowej Rady Sądownictwa wskazanego przez Klub Parlamentarny w druku nr 1124.

Ta lista zawiera jedną pozycję, jedno nazwisko. Kandydatem do Krajowej Rady Sądownictwa jest pani sędzia Katarzyna Ewelina Chmura. W imieniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka proszę o zatwierdzenie tej listy, a więc wskazanie na wybór pani sędzi Katarzyny Eweliny Chmury. Dziękuję. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Otwieram dyskusję. Proszę.

Wysoka Izbo! Dzisiaj politycy PiS będą wybierali sędziowskiego członka Krajowej Rady Sądownictwa. My jako klub nie przyłożymy do tego ręki. Jest to na wskroś niezgodne z polską konstytucją. Art. 187 mówi jasno o tym, że Sejm ma prawo wybrać czterech członków przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, czterech i ani jednego więcej. Wysoka Izbo! Wszyscy na tej sali wiedzą, że wybór sędziowskich członków do Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Wiedzą to posłowie, wiedzą to także kandydaci, ale wiedzą to też wszyscy prawnicy w Polsce. Proszę spojrzeć, z 10 tys. sędziów w Polsce do instytucji cieszącej się niegdyś szacunkiem, poważaniem, stojącej niegdyś na straży niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości kandydują dzisiaj zaledwie trzy osoby. Są to dwie nikomu nieznane panie i człowiek, o którym media pisały, że miał być określany mianem herszta w grupie mającej stać za kampanią hejtu. I nawet oni są popierani w większości tylko przez sędziów, którzy coś od tej władzy otrzymali. Pod ich listami poparcia podpisali się w większości sędziowie, którzy coś tej władzy zawdzięczają, czy to awans, czy funkcję prezesa, czy coś innego. Wysoka Izbo! To, co jest najgorsze, to to, że obecna władza, stojąc nad przepaścią prawną, zamiast zrobić krok wstecz, robi krok do przodu. Wiecie, że wybierając w Sejmie sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa, łamiecie regułę praworządności. Wiecie, że na szali leżą miliardy złotych z budżetu unijnego, z funduszów pomocy. Ale robicie to mimo wszystko, szkodząc sobie, szkodząc Polkom i Polakom, a wszystko to, byle tylko zaspokoić jakieś szaleńcze wizje Ziobry od 6 lat niszczącego niezależność wymiaru sprawiedliwości. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Jako prawnik, ale i obywatel, najzwyczajniej w świecie mam poczucie uczestnictwa w jakiejś koszmarnej procedurze, w której jak gdyby nigdy nic partia rządząca wystawia kandydatkę do Krajowej Rady Sądownictwa, która w świetle konstytucji, uchwał Sądu Najwyższego, orzecznictwa sądów międzynarodowych nie spełnia podstawowego kryterium, czyli kryterium niezależności, oraz kryterium działania na podstawie solidnego prawa. Mam poczucie najwyższego zażenowania i to moje poczucie najwyższego zażenowania podzielają nie tylko członkowie i członkinie klubu Lewicy, ale i setki tysięcy obywateli i obywatelek, którzy od lat angażują się w obronę niezawisłych sędziów i niezależności sądów. Dzisiaj partia rządząca, zasłaniając się bezprawnymi przepisami, udaje, że kandydatką do KRS-u jest przedstawicielka środowiska sędziowskiego. A tak naprawdę wbrew wymogowi konstytucyjnemu jest kandydatką władzy ustawodawczej. 2017 r. - Sejm dokonuje największego zamachu na niezależność sądową, jakim jest wygaszenie kadencji sędziów KRS. 2020 r., styczeń - bezprecedensowa uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego, cywilnej, karnej, pracy i ubezpieczeń społecznych, które stwierdziły co? Czego jeszcze potrzebujemy, aby stwierdzić, że mamy do czynienia z farsą demokracji? Wysoka Izbo! Lewica nie będzie uczestniczyła w tej farsie, bo niby-wybór do niby-KRS byłby zdradą obywateli. Nie wpiszemy się w zakłamany scenariusz i nie przejdziemy nad tym głosowaniem, udając, że uzupełniamy skład konstytucyjnego organu. KRS wydaje zatrute owoce. Nominuje sędziów, którzy potem wydają wyroki, które można obalać z uwagi na fakt, że wydawali je niesędziowie. Lewica nie przyłoży ręki do pogłębiania chaosu prawnego w naszym kraju.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Prawo i Sprawiedliwość w ramach procesu wieloletniego już dewastowania polskiego wymiaru sprawiedliwości zamieniło konstytucyjny organ obdarzony szacunkiem, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej, jakim była Krajowa Rada Sądownictwa, w siedlisko prymitywnych hejterów internetowych, którzy skupiają się - do niedawna jeszcze było o tym głośno - na tym, jak najwięcej kasy wyciągnąć za tzw. diety, nawet za czytanie literatury, zdaje się, w czytelniach czy w bibliotekach.

Ale dla obywateli polskich najważniejsze jest to, że już wiedzą po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, całkiem niedawno wydanym, że sędziowie, którzy orzekają w takich w sądach po powołaniu przez Krajową Radę Sądownictwa... że takie wyroki mogą być podważone. Mogą być skutecznie podważone nie przez organa Unii Europejskiej, tylko przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, organizację, która stoi na straży praworządności krajów członkowskich, ma siedzibę w Strasburgu i nie ma wiele wspólnego z Unią Europejską. Warto o tym przypomnieć. Dlatego, podzielając poglądy klubów opozycyjnych, wypowiedziane tutaj wcześniej. klub Koalicji Polskiej będzie jednak w tym głosowaniu uczestniczył, oczywiście głosując przeciwko tej kandydaturze.

Wysoki Sejmie! Szkoda, że poseł sprawozdawca dokładniej nie powiedział, jak przebiegało posiedzenie komisji sprawiedliwości. W tej sprawie właściwie należałoby milczeć, wyjąć karty i wyjść z sali plenarnej. Popieranie jakichkolwiek kandydatów do tak wadliwie ukształtowanej i tak nieprawidłowo funkcjonującej neo-KRS byłoby wspieraniem działania instytucji, która działa wbrew swej konstytucyjnej misji i przyczynia się do pogłębiania chaosu prawnego w Polsce. Przyczynia się do pogłębiania chaosu, ale także osłabia standard prawa człowieka do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, o czym, jak już mówiliśmy na posiedzeniu komisji sprawiedliwości, mówi art. 45 konstytucji. Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z.

Przedmiotem w tej chwili będzie wybór uzupełniający sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa. a trybunał już się wypowiedział na temat zgodności działania z konstytucją Krajowej Rady Sądownictwa. W tej sytuacji oczywiście Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za kandydaturą pani Katarzyny Chmury.

W przypadku niedokonania wyboru członków rady we wskazanym wyżej trybie Sejm, zgodnie z art. 11d ust. 6 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, wybiera członków rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując ponownie na tę samą listę kandydatów ustaloną przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem pani Katarzyny Eweliny Chmury na stanowisko sędziego - członka Krajowej Rady Sądownictwa, zechce nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm większością 3/5 głosów wybrał panią Katarzynę Ewelinę Chmurę na stanowisko sędziego-członka Krajowej Rady Sądownictwa. Zarządzam 5 minut przerwy.

Wznawiam obrady. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk nr 1090) Proszę panią poseł Barbarę Bartuś o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawczej przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawarty w druku sejmowym nr 1090. Projektowana ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r., stwierdzającego niezgodność art. 156 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 156 § 2 k.p.a. w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 konstytucji. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu przypomniał, że możliwość stwierdzenia nieważności decyzji jest wyjątkiem od zasady poszanowania trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej. Jednocześnie podniósł, że brak wyłączenia dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej z przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. po znacznym upływie czasu skutkuje destabilizacją porządku prawnego, jeżeli decyzją przyznano stronie ekspektatywę nabycia prawa, z której zamierza ona skorzystać. W tym kontekście Trybunał zwrócił uwagę, że ustawodawca określając przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji oraz zakres ich zastosowania, powinien brać pod uwagę wszystkie zasady mieszczące się w klauzuli państwa prawnego przewidzianej w art. 2 konstytucji, a odstępstwa od zasady trwałości decyzji ostatecznej nie powinny naruszać wynikających z art. 2 konstytucji zasad bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. W konkluzji swego wyroku Trybunał podniósł, że stabilizacja stanów faktycznych, po upływie określonego czasu, leży w interesie porządku publicznego. Ponadto, zważywszy na tło faktyczne sprawy P46/13, podkreślił, że z czasem wzrasta ryzyko prawne polegające na możliwości wykształcenia się odmiennej linii orzeczniczej zarówno w stosunku do norm materialnych i procesowych, które legły u podstaw wydanej decyzji, jak i samej przesłanki rażącego naruszenia prawa. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jako dotyczący tzw. pominięcia prawodawczego, a przy tym mający formułę zakresową, nie doprowadził do delegowania art. 156 § 2 k.p.a. z porządku prawnego. Dlatego też Trybunał w swoim orzeczeniu podkreślił, że stwierdzenie niekonstytucyjności w zakresie pominięcia prawodawczego nakłada na ustawodawcę obowiązek rozszerzenia unormowania art. 156 § 2 k.p.a., przewidującego ograniczenia możliwości stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ustawodawczej proponuję, aby wszelkie wady kwalifikowane jako rażące naruszenie prawa były objęte 30-letnim terminem przedawnienia.

Oceniając zarzuty kasacyjne w przedmiotowej sprawie, stwierdził, że w ocenie NSA okres, po którym niedopuszczalne byłoby stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, powinien być znacząco dłuższy niż w przypadku innych przyczyn. Przypomnę, że co do zasady jest to 10 lat. NSA nawiązał do przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zasiedzenia. Z art. 172 § 2 k.c. wynika, że po upływie 30 lat posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. W przepisach przejściowych proponujemy, aby do postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosować przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Naszym zdaniem jest to wystarczający czas, który umożliwi tak organom stosującym prawo, jak i adresatom decyzji zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwsza pani poseł Barbara Bartuś w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W ocenie Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca ma wręcz obowiązek kształtowania regulacji prawnych, które będą sprzyjały wygaszaniu wraz z upływem czasu stanu niepewności. Niezbędne jest zatem ustanowienie odpowiednich granic dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji. Trwałość decyzji organów władzy publicznej nie może być pozorna. Taka pozorność występowałaby nie tylko, jeżeli ustawodawca nie przewidywałby ograniczeń wzruszalności ostatecznych decyzji, ale również jeżeli ograniczenia te nie byłyby wystarczające dla zachowania zasady zaufania obywatela do państwa i zasady pewności prawa. Ustawodawca nie może z jednej strony deklarować trwałości decyzji z uwagi na jej ostateczność, a z drugiej strony przewidywać nieograniczoną terminem możliwość wzruszania decyzji, na podstawie której strona nabyła prawo lub ekspektatywę. W szczególności następuje to w razie powołania się na otwartą i nieostrą przesłankę rażącego naruszenia prawa.

Tam Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że możliwość stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, mocą której nastąpiło nabycie prawa lub ekspektatywy nabycia praw, ograniczona jest terminem 10 lat, liczonych od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Uwzględniając zasadę nadrzędności konstytucji, art. 8 ust. 1, a ponadto zasady demokratycznego państwa prawnego, art. 2 konstytucji, oraz legalizmu, art. 7 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy podkreślić, że działanie organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa oznacza przede wszystkim działanie zgodnie z konstytucją, a w razie wątpliwości co do jej zgodności - z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny w tym orzeczeniu, w składzie rozpoznającym skargę na orzeczenie WSA, zajął stanowisko, iż możliwość stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, mocą której nastąpiło nabycie prawa lub ekspektatywy nabycia praw, ograniczona jest terminem 10 lat, liczonych od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. I takich wyroków naczelnego sądu jest więcej.

Chciałam tu podkreślić, że Komisja Ustawodawcza w swoim projekcie tak naprawdę tylko wykonywała orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego, tak jak powiedziałam na wstępie, opowiadamy się za skierowaniem tego projektu do dalszych prac. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Zwiefka, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyrażam duże zadowolenie z powodu faktu, iż nastąpiło przedłożenie ze strony Komisji Ustawodawczej projektu w tak istotnej kwestii jak uznanie i konsekwentne wdrożenie legislacyjne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. w sprawie, która jest istotna dla wielu indywidualnych obywateli, ale także dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących w naszym kraju. To już trzecie podejście, trzecia próba załatwienia tej kwestii. Pierwsza miała miejsce w roku 2016, kiedy Komisja Ustawodawcza polskiego Senatu podjęła prace w tej właśnie kwestii, ale one niestety nie zakończyły się powodzeniem. Później była próba generalnego podejścia do reformy Kodeksu postępowania administracyjnego - również zakończona niepowodzeniem. I tym razem - mam nadzieję, że zgodnie ze staropolskim powiedzeniem: do trzech razy sztuka - po raz trzeci tym razem Sejm podejmuje prace, by wypełnić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Orzeczenie, które tak naprawdę nie zmienia niczego w istniejącym porządku prawnym, wskazuje wszakże na lukę, która w nim się znajduje, mówimy tutaj o art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. W zasadzie w pełni mogę zgodzić się z uzasadnieniem, które zostało przedłożone przez Komisję Ustawodawczą. Natomiast z wnioskami, które zostały wyciągnięte w tej kwestii - już niekoniecznie.

Przywołane wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego oczywiście są istotne. Brakuje mi wszakże opinii tegoż sądu. Nie wiem, czy zwróciliśmy się o taką opinię, czy też powinniśmy to zrobić w najbliższej przyszłości, kontynuując prace nad tym projektem.

Ale po to, by znaleźć właściwe rozwiązanie, niezbędne są dalsze prace. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że nie do końca mogę się zgodzić z propozycją, aby sprawy, które są już w toku, ale nie zakończyły się ostateczną decyzją, były po wejściu w życie tej ustawy rozstrzygane w oparciu o te nowe przepisy. Zatem sugerowałbym, abyśmy te nowe przepisy odnieśli do spraw, które rozpoczną się po wejściu w życie ustawy bądź które nie zostały rozpoczęte przed jej wejściem w życie. Pani poseł Bartuś stwierdziła, że ten krótki okres kilkutygodniowy jest wystarczający. Wydaje się, że aby właściwie przygotować się do stosowania tego nowego przepisu, lepszy byłby jednak okres kilkumiesięczny (Dzwonek), przynajmniej 3-miesięczny, by wszyscy rzeczywiście zdążyli się z tym nowym prawem zapoznać. To także pozwoliłoby ewentualnie osobom zainteresowanym, które mogłyby sprawę rozpocząć. Już kończę, panie marszałku, przepraszam bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska chciałbym prosić o przekazanie tego projektu do nadzwyczajnej komisji kodyfikacyjnej celem kontynuowania prac nad tym projektem. Teraz pani poseł Magdalena Biejat, klub Lewicy. Wysoka Izbo! Reprywatyzacja od lat jest źródłem tragedii tysięcy obywateli. Utrudnia życie lokatorom, posiadaczom i kupującym nieruchomości, rujnuje budżety samorządów i łamie życiorysy zwykłych ludzi. Przez ostatnie ćwierć wieku na tej sali wypowiedziano na ten temat ocean słów, ale nie zrobiono właściwie nic. Art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego jest źródłem tragedii ofiar reprywatyzacji, ale także bolączką wszystkich obywateli, którzy nie mogą w pełni zaufać decyzjom, które zapadają w ich sprawach. Odwracanie decyzji administracyjnych po kilkudziesięciu latach od ich wydania, które jest istotą reprywatyzacji, bulwersuje społeczeństwo, bo dotyka elementarnego poczucia sprawiedliwości i praworządności. Z jednej strony stoi zasada legalizmu, która wymaga korygowania decyzji wydanych ze znaczącym naruszeniem prawa. Z drugiej strony są decyzje sprzed 60 lat, które dziś uznaje się za wadliwe, ale dzięki którym podniesiono z gruzów stolicę, wybudowano setki szkół i budynków użyteczności publicznej, mieszkania komunalne i socjalne, mamy parki, po których spacerują ludzie, w których bawią się dzieci, mamy utrwalony przez ponad 60 lat porządek społeczny i prawny. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że możliwość unieważniania decyzji administracyjnych wydanych z rażącym naruszeniem prawa, od których wydania upłynęło wiele lat, a decyzja była podstawą nabycia praw lub ekspektatywy, którą umożliwia obecnie art. 156 k.p.a., jest niezgodna z konstytucją. Trybunał zobowiązał tym samym ustawodawcę do zmiany tego przepisu. Niestety, mimo upływu 6 lat rządów PiS, mimo wcześniejszych zapewnień Patryka Jakiego, że uporacie się ze sprawą warszawskiej i nie tylko warszawskiej reprywatyzacji, mimo tego że podobno cenicie sobie porządek prawny - realnie nie zrobiliście nic. Ustawy reprywatyzacyjnej jak nie było, tak nie ma, ciągle cofane są decyzje, które zapadły ponad 60 lat temu, a ludzie nadal tracą dach nad głową. Na tym, że brakuje jasnych i ostatecznych przepisów regulujących to, jak zwracane są przejęte przez Polskę Ludową grunty, cierpią przede wszystkim lokatorzy, ale cierpi też cała reszta społeczeństwa. Na mocy art. 156 k.p.a. reprywatyzowane są szkoły, domy kultury, budynki użyteczności publicznej, zabytki i parki, likwidowane są bazary, tak jak ostatnio na warszawskiej Sadybie, samorządy tracą tereny przewidziane pod usługi publiczne, nagle w gruzach legną plany powstania szkół czy przychodni zdrowia. Dlatego nieustannie zabiegamy o uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej oraz doprecyzowanie obecnych przepisów. Niestety, ustawa reprywatyzacyjna Lewicy, która kompleksowo i ostatecznie rozwiązuje problem reprywatyzacji, która uniemożliwia zwroty w naturze, która ustala uczciwe wysokości odszkodowań, ustawa, którą stworzyliśmy w porozumieniu z przedstawicielami lokatorów, którą szeroko konsultowaliśmy i która uzyskała aprobatę licznych ekspertów, nadal nie doczekała się uwagi ze strony pani marszałek Sejmu i nie trafiła pod głosowanie. Ale bezczynność Sejmu i koalicji rządzącej nie powstrzymuje dramatów ludzi. Lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych ciągle obawiają się o to, czy nie pojawią się roszczenia do ich domów. Tam gdzie te roszczenia są, ludzie nie śpią po nocach, bojąc się, że wyroki ostatecznie zapadną i będą musieli opuścić domy, w których mieszkają całe życie. Na warszawskiej Pradze ratusz wstrzymuje podłączenie ogrzewania w kamienicach, skazując mieszkańców na niebotycznie drogie ogrzewanie elektryczne, wpędzając ich w nędzę i w choroby. Ciągle przybywa bloków, które zostały wybudowane w latach 60. czy 80. na gruntach, do których dzisiaj znikąd pojawiają się roszczenia. To mieszkania, które ciężko sprzedać i równie ciężko kupić, bo banki nie udzielają na nie kredytów hipotecznych, a spółdzielnie mieszkaniowe, do których należą, nie chcą inwestować w ich remonty i modernizację. Lewica poprze ten projekt, bo jest potrzebny obywatelom, w szczególności zaś mieszkańcom Warszawy, którym nadal zagraża reprywatyzacja. Obecnie k.p.a. przewiduje 10-letni okres na odwrócenie wadliwych decyzji. Z niezrozumiałych przyczyn kodeks przewiduje jednak wyjątki nieopatrzone żadnym terminem. Zaliczają się do nich m.in. decyzje na mocy tzw. dekretu Bieruta. Konstytucyjna zasada pewności prawa, kluczowa dla stabilności państwa, jego autorytetu oraz zaufania społecznego, wymaga, aby przepisy te ujednolicić i uznać, że dla wszystkich decyzji przyjmujemy taki sam, 10-letni okres, po którym uznaje się je za ostateczne i nieodwracalne. Dlatego złożymy stosowną poprawkę. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak podkreślają eksperci, to bardzo ważna zmiana dla administracji publicznej i dla obywateli zainteresowanych decyzjami wywłaszczeniowymi. Gdyby zaczął obowiązywać przepis, który został zaproponowany w projekcie, nieważność wydanych dawniej decyzji zostałaby wyłączona. W świetle dotychczasowych zaniechań ustawodawcy wniesioną obecnie do Sejmu RP inicjatywę ustawodawczą należy ocenić pozytywnie. Należy jednak zapytać, dlaczego musieliśmy taki długo czekać na nowelizację. Od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie mija już przecież 5 lat. Przyjęcie niezwykle długiego, bo 30-letniego terminu przedawnienia, nie znajduje przekonujących podstaw. Przeciwnie, może ono spotkać się z zarzutem zachwiania wewnętrznej spójności regulacji art. 156 k.p.a., braku uwzględnienia współczesnych potrzeb społeczno-gospodarczych, a także niekonsekwencji ustawodawcy wobec przeciwnych tendencji zmian ustawowych obserwowanych w prawie materialnym.

Można bowiem postawić pytanie: czemu decyzja przenosząca prawo własności nieruchomości wydana z rażącym naruszeniem prawa może podlegać stwierdzeniu nieważności przez okres całych 30 lat, a tożsama decyzja przenosząca prawo własności nieruchomości, lecz wydana przez organ oczywiście niewłaściwy w sprawie - już jedynie przez okres 10 lat? Czy rzeczywiście różnica w kategorii wady prawnej decyzji może uzasadniać aż tak daleko idące zróżnicowanie ochrony praw nabytych adresatów decyzji administracyjnej? Wydaje się, że argument z analogii do zasiedzenia nieruchomości nie jest tutaj właściwy. Mógłby on stanowić co najwyżej podstawę do wprowadzenia szczegółowego okresu przedawnienia wzruszalności decyzji przenoszących prawo własności nieruchomości z jakiejkolwiek przyczyny nieważności, nie zaś dla zróżnicowania okresu przedawnienia decyzji w zależności od jej wady prawnej. Konkretne przypadki wad nieważności są na tyle silnie zróżnicowane, że próba gradacji tych wad rodzajowo od najbardziej do najmniej poważnych jest ryzykowna, a już z całą pewnością nie powinna opierać się na intuicji niepopartej żadnymi konkretnymi argumentami. Ze względu na przytoczone argumenty wydaje się, że przedłożony w Sejmie projekt nowelizacji wymaga jeszcze pogłębionej refleksji. Wydaje się, że nowelizacja art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego powinna raczej zmierzać do jednakowego traktowania przedawnienia stwierdzenia nieważności decyzji w odniesieniu do każdej z wad wskazanych w art. 156 § 1 Ewentualne odstępstwa od tej zasady powinny odnosić się do poszczególnych kategorii decyzji, np. wspomnianych w uzasadnieniu projektu decyzji przenoszących prawo własności nieruchomości.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof Tuduj, koło Konfederacji.

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Na tę ustawę czekamy od 2016 r., od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W międzyczasie powstała komisja do spraw reprywatyzacji warszawskich, która zagrzebała trwające kilkadziesiąt lat postępowania w dalszych problemach prawnych. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że większość decyzji reprywatyzacyjnych mogło zostać wzruszonych jedynie na podstawie istniejących już przesłanek k.p.a., tj. m.in. wydania decyzji reprywatyzacyjnych z rażącym naruszeniem prawa skierowanych do osoby niebędącej stroną czy wydania decyzji w wyniku przestępstwa.

Trybunał Konstytucyjny wskazywał już 12 maja 2015 r., że przesłanki do nadzwyczajnego zaskarżenia decyzji, tj. do stwierdzenia nieważności decyzji, powinny obowiązywać znacznie dłużej niż 10 lat dotychczas przewidzianych w kodeksie. Gdyby miał dobrą wolę, by rozwiązać m.in. sprawy dotyczące reprywatyzacji warszawskich, ale także innych, to ten projekt zajmujący zaledwie jedną stronę, pojawiłby się dużo wcześniej, bo na początku rządów PiS-u. W zamian PiS zdecydował się na bardzo drogą kampanię wyborczą w Warszawie, która i tak zapewniła miażdżące zwycięstwo kandydatowi totalnej opozycji. Sprawy dotyczące własności nieruchomości w Warszawie, a które trwają już od dekretu Bieruta, nie zostały rozwiązane i nie zanosi się na to, aby komisja reprywatyzacyjna miała je rozwiązać. Mam nadzieję, że wypłacane poszkodowanym odszkodowania nie będą podważane przez kolejne rządy osób, które będą chciały zamieść pod dywan aferę reprywatyzacyjną. Apeluję z tego miejsca: nie psujcie państwo prawa, częściej zaglądajcie do orzeczeń sądów i trybunałów, które w dużej mierze rozwiązują istniejące problemy. 30-letni termin przedawnienia nawiązuje do uregulowań Kodeksu cywilnego, tj. instytucji zasiedzenia nieruchomości w złej wierze, i jest w tym przypadku naszym zdaniem jak najbardziej prawidłowym rozwiązaniem. Dziękuję za uwagę. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koło Parlamentarne Polska 2050 zasadniczo popiera przedstawiony projekt ustawy jako wykonujący niezwykle doniosły i słuszny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r.

Należy przypomnieć, że zmieniany artykuł dotyczy przypadków nadzwyczajnych, w których organ administracji publicznej może stwierdzić nieważność już wydanej, prawomocnej decyzji administracyjnej pozostającej w obrocie prawnym. Tego typu decyzje są zawsze trudne i mogą być podejmowane z wyjątkową starannością, gdyż eliminacja z obrotu już obowiązujących decyzji zawsze narusza interesy osób, które w oparciu o te decyzje, często w dobrej wierze, podejmowały różne działania i prowadziły swoje, często bardzo ważne, sprawy życiowe. Trybunał orzekał w tej sprawie, odpowiadając na pytanie prawne zadane przez WSA w Warszawie na kanwie sprawy reprywatyzacyjnej. To właśnie w sprawach reprywatyzacyjnych dochodziło bardzo często do wzruszania na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 4 k.p.a. decyzji nacjonalizacyjnych wydanych dziesiątki lat temu, co prowadziło niejednokrotnie do rewolucyjnych zmian w życiu wielu osób, nie tylko nowych beneficjentów reprywatyzacji, ale także np. lokatorów mieszkań w kamienicach komunalnych. Cieszę się więc, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., choć miał charakter interpretacyjny i zakresowy, stał się podstawą setek rozstrzygnięć sądów administracyjnych, które odmawiały wzruszania kolejnych decyzji zapadłych dziesiątki lat temu. Szkoda, że dopiero dziś, po 6 latach od wydania orzeczenia, Sejm proceduje nad ustawą normalizującą w pełni tę kwestię i wykonującą wyrok trybunału. Wydaje się jednak, że projekt ma dwie zasadnicze wady.

Termin 30-letni jest aż trzydziestokrotnie dłuższy od 10-letniego terminu przewidzianego w art. 156 § 2 k.p.a., obowiązującego w wypadku podważania decyzji wydanych z naruszeniem przepisów o właściwości dotyczących spraw już poprzednio rozstrzygniętych inną decyzją ostateczną, skierowanych do osoby niebędącej stroną w sprawie czy zawierających wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. Zawarte w uzasadnieniu odniesienie terminu zasiedzenia nieruchomości w złej wierze do Kodeksu cywilnego należy uznać za błędne. Po pierwsze, jest to termin prawa cywilnego nie zaś administracyjnego, dodatkowo setki tysięcy decyzji administracyjnych wydawanych jest codziennie w bardzo szerokiej gamie spraw, nie tylko dotyczących nieruchomości. Polska 2050 proponuje zatem, aby wprowadzić w tym wypadku termin 10-letni, taki sam jak w przypadku innych przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji z art. 156 k.p.a., o których była wcześniej mowa. Należy zauważyć, że 30-letni termin należy do najdłuższych terminów znanych polskiemu prawu. Wydaje się, że wprowadzenie tak długiego terminu nie wypełnia intencji wyroku TK, który dążył do kompromisu między zasadą legalizmu a zasadą zaufania obywatela do państwa. Termin 30-letni przyznaje ewidentnie w dalszym ciągu zdecydowany prymat zasadzie legalizmu, skoro pozwala wzruszać decyzje zapadłe pokolenie wcześniej. Podważanie takich decyzji niemal zawsze będzie prowadziło do pogłębiania się chaosu prawnego i konieczności kaskadowego unieważniania kolejnych czynności prawnych podejmowanych już wiele lat temu, często przez osoby fizyczne lub nieżyjące, lub osoby prawne nieistniejące. Jednocześnie Polska 2050 nie kwestionuje możliwości zastosowania nowych przepisów do postępowań w toku. Taka możliwość jest uzasadniona faktem obowiązywania już od 6 lat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które jest wykonywane niniejszym projektem ustawy. Uczestnicy obrotu mieli więc od lat świadomość (Dzwonek), że możliwość domagania się wzruszenia decyzji administracyjnych sprzed dziesięcioleci jest przynajmniej prawnie wątpliwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

14-dniowy termin wejścia w życie ustawy może utrudnić organom wydającym decyzje administracyjne oraz adresatom tych decyzji zapoznanie się ze zmianami i zakończenie trwających postępowań administracyjnych. Stąd moje pytanie: Czy zostanie rozważona możliwość wydłużenia tego terminu? Wątpliwości budzi też zapis dotyczący postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Czy autorzy projektu mają świadomość, że może to doprowadzić do takiej sytuacji, że trwające postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych nie będą mogły zostać zakończone i rozstrzygnięte, mimo że zostały wszczęte zgodnie z obowiązującym od lat stanem prawnym? Wysoka Izbo! Wprowadzenie 30-letniego okresu, w którym dopuszcza się możliwość podważenia złej decyzji administracyjnej, może wydawać się celowe i dające gwarancję dochodzenia swoich roszczeń w wydłużonym czasie. Jednak wraz z upływem czasu wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności powodujących nieodwracalność skutków decyzji administracyjnej wydanej z naruszeniem prawa. Mam pytanie do rządu, czy nie obawia się, że sytuacja taka może doprowadzić do rozchwiania systemu prawnego, w którym z jednej strony decyzja administracyjna powinna zostać podważona, a z drugiej strony skutki owej decyzji nie mogą zostać odwrócone. Prowadzi to do powstania sytuacji niejednoznacznych, które przecież chcemy wyeliminować z naszego systemu prawnego. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Projektowana ustawa przewiduje zmianę w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego przez dodanie nowego § 3, zgodnie z którym nie stwierdza się nieważności decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 30 lat, a decyzja ta była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa. Pierwszy to ten długi, 30-letni okres, na który m.in. zwraca również uwagę prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dużym optymizmem przyjąłem informację pani poseł, że ten projekt ustawy będzie jeszcze dopracowywany, [[Dzwonek]] czyli będzie praca w komisjach.

Szanowny Panie Marszałku! Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2015 r. długo leżał, aż wreszcie się doczekał projektu naprawczego w postaci wprowadzenia nowych przepisów w ustawie - Kodeks postępowania administracyjnego. W 2018 r. rzecznik praw obywatelskich pytał ministra spraw wewnętrznych i administracji pana ministra Brudzińskiego o zaawansowanie prac nad rozwiązaniem tego problemu, o którym powiedział Trybunał Konstytucyjny. Rozważano, jakie są orzeczenia sądowe w tej prawie.

Jakie jest państwa stanowisko w sprawie terminu wejścia w życie ustawy? Czy 30-letni okres jest okresem odpowiednim?

Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! To bardzo ważne przedłożenie, które powinno znaleźć się w niedługim czasie w polskim porządku prawnym. To nie tylko wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale kolejny krok, który podjęliśmy w ramach regulacji tego, co poprzednie władze narobiły w zakresie reprywatyzacji w Polsce: wielkie afery, krzywda tysięcy ludzi, niejasny stan prawny. Od razu po przejęciu władzy zaczęliśmy prace w wielu obszarach i dzisiaj krok po kroku wyjaśniamy te wszystkie problemy, które narosły przez kilkanaście lat.

Wiele afer korupcyjnych, jedna nieruchomość pod drugiej, ludzie którzy musieli być eksmitowani przez osoby, które nie miały prawidłowych tytułów prawnych - dzisiaj to wszystko wyjaśniamy, krok po kroku, konsekwentnie. Czas mija, ale nasza ciężka praca daje owoce. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim stronom, wszystkim klubom, które zabrały głos, że popierają kierunek, który jest przyjęty w tym projekcie. Niemniej czuję się w obowiązku odnieść do kilku kwestii dotyczących i tempa proponowania tych przepisów, i ewentualnych zaniechań, które doprowadziły do sytuacji, w której nasz rząd, nasza większość od lat naprawia te patologie, które niestety miały miejsce w wielu miastach w Polsce. Platforma Obywatelska płacze 5 lat, że nie ma wykonania wyroku. Gdybyście nie paraliżowali prac komisji weryfikacyjnej, zapewne byśmy byli w lepszym miejscu niż dzisiaj. Tylko przypominam: to wy ponosicie odpowiedzialność, że ta afera w ogóle wybuchła. tę większość parlamentarną, która wzięła się za to, wypaliła gorącym żelazem te patologie i dzisiaj konsekwentnie blokuje ścieżki powrotu tych wszystkich mechanizmów, gdyby - nie daj Boże - Platforma wróciła do władzy. A co wy robiliście w koalicji z Platformą, kiedy Hanna Gronkiewicz Waltz i podlegli jej urzędnicy doprowadzili do tej wielkiej afery?

Rozumiem, że może nie pani osobiście, ale mówię o ugrupowaniu politycznym, które pani reprezentuje. Otóż zrobiono. Mieszkańcy nie są wyrzucani z domów. Zabezpieczyliśmy poprzednio w ustawie o UGN niemożność reprywatyzacji takich nieruchomości. Mieszkańcy pokrzywdzeni dostali odszkodowania.